Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Paulinę Matysiak, Aleksandrę Szczudło, Konrada Frysztaka i Daniela Milewskiego. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Aleksandra Szczudło i Daniel Milewski. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Aleksandra Szczudło i Konrad Frysztak. Proszę panią poseł sekretarz o odczytanie komunikatów.

W dniu dzisiejszym odbędzie się również wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Elektromobilności i Energetyki Prosumenckiej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce - godz. 14. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Przystępujemy do pierwszego pytania.

Bardzo proszę, panie pośle, o pierwsze pytanie. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 2 minuty, dlatego też bardzo szybko - argumenty przemawiające za tym, żeby sołectwo Mścice zostało w gminie Będzino, bo dzisiaj o tym mówimy. Mieszka tam prawie 2 tys. mieszkańców, co stanowi aż 20% mieszkańców całej gminy. Na 244 zarejestrowane działalności gospodarcze w gminie 133 znajdują się tam, czyli 55% wszystkich działalności gospodarczych to jedno sołectwo. Mścice to osobna jednostka osadnicza oddzielona od Koszalina 4-kilometrowym lasem i w żaden sposób niepołączona z miastem Koszalinem. Rolnicy i jeden z wiodących ośrodków hodowli zarodowej w Polsce po włączeniu w granice administracyjne Koszalina stracą możliwość korzystania z PROW-u - linia demarkacyjna nie pozwoli im korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co rolnicy zrobili, aby tak ich karać?

Co ważne, do tych placówek oświatowych uczęszcza wiele dzieci z innych miejscowości w gminie Będzino, które mają do Mścic blisko, ale też te jednostki budowane były wysiłkiem całej społeczności gminy, aby służyły tej społeczności. Szanowny Panie Ministrze! Kilka lat wcześniej, za rządów PO, do miasta Koszalina zostały włączone Jamno i Łabusz. Myśli pan, że one mają dzisiaj podgrzewane chodniki? Nic się nie zmieniło, panie ministrze. I mam nadzieję, że (Dzwonek) to doświadczenie spowoduje, że jednak tego nie zrobimy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiany w podziale terytorialnym państwa stopnia gminnego, w tym dotyczące zmian granic gmin, następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i z uwzględnieniem zasad i procedur określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach. Zgodnie z ww. przepisami wnioskodawcą w sprawie zmian w podziale terytorialnym państwa na szczeblu gminnym może być zainteresowana rada gminy. Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stosowny wniosek winien być poprzedzony przeprowadzeniem przez daną radę konsultacji z mieszkańcami, opatrzony uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku. Powyższy przepis wymaga również opinii rad gmin objętych wnioskiem poprzedzonych przeprowadzonymi przez te rady konsultacjami z mieszkańcami, zaś w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granicę powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw. Rada gminy występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem właściwego wojewody, w terminie do 31 marca. Wojewoda zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Chciałbym zwrócić uwagę, że wniosek, o którym mówił pan poseł, nie jest procedowany z urzędu przez Radę Ministrów, nie jest także na wniosek Rady Ministrów podejmowany. Jest to wniosek podejmowany przez miasto Koszalin i dotyczy włączenia do obszaru miasta Koszalina obszaru trzech sołectw. Jest on w tej chwili analizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Także kwestie, o których mówił pan poseł, są analizowane.

Wniosków w skali kraju jest więcej.

Myślę, że także w tym roku tak będzie. Zaplanowane już jest posiedzenie zespołu komisji wspólnej rządu i samorządu, który będzie opiniował ten wniosek zgodnie z zasadami. I ta decyzja zgodnie z procedurą zostanie podjęta. Dziękuję bardzo. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Jarosław Rzepa. Panie Marszałku!

Dopytam jeszcze w takim razie o Sianów i o Łazy. To kolejny wniosek. Kolejny wniosek, bo gmina sobie wymyśliła, że chce mieć dostęp do morza - dostęp do morza kosztem gminy Mielno. Ludzie powiedzieli: nie, wojewoda, choć niejednoznacznie, też. Rady gmin zarówno w Będzinie, jak i w Mielnie powiedziały stanowcze ˝nie˝ I mam nadzieję, panie ministrze, że wreszcie się z nimi pan spotka, bo oni pana proszą, zarówno Mścice, jak i Mielno. Nie chce się pan z nimi spotkać. Widzę, że panu zależy na tym, żeby jednak ta procedura przeszła cicho.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan minister Paweł Szefernaker. Ja bym prosił jednak, żeby z mównicy sejmowej nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Po pierwsze, mieszkańcy gminy Mielno, bo pan ten wątek także tutaj podjął. Wielokrotnie w moim biurze poselskim rozmawialiśmy na ten temat, bo jest grupa osób, która chce, prosi, złożyła wniosek, podpisała, o to, aby. Ten wniosek jest procedowany. To, że pan tego nie widział, nie znaczy, że nikt tego nie widział. To po pierwsze.

Po trzecie, proszę nie mówić, że ja nie chcę się spotkać, ponieważ zorganizowałem spotkanie z panią burmistrz Mielna, na które nie przyszła. Więc bardzo proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Po czwarte, są zorganizowane kolejne spotkania z mieszkańcami, które - myślę - pozwolą Radzie Ministrów przyjąć taką opinię, która będzie do zaakceptowania. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Ja rozumiem, że pan po prostu poczuł, że jest tutaj możliwość zadania pytania, trochę zakręcenia.

Proszę, panie pośle, naprawdę nie warto tutaj kłamać. Proszę również wziąć pod uwagę, panie pośle.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Grzegorz Lorek, Krzysztof Kozik, Barbara Bartuś, Mariusz Trepka i Marek Polak kierują pytanie do ministra finansów. Pierwsze pytanie zadają posłowie Grzegorz Lorek i Marek Polak. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Panie i Panowie!

To dane lepsze od oczekiwań. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji z przewodniczącą Komisji Europejskiej powiedział: Polska rozpoczęła już realizację KPO, gdyż nie możemy czekać po pandemii z tak ważnymi inwestycjami. Panie Ministrze! Czy obecne rozstrzygnięcia w zakresie Polskiego Ładu mają znaczenie we wzroście gospodarczym naszego kraju? Jeżeli tak, to jakie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku!

Ale ze zdumieniem odczytuję wyniki Eurostatu, które wskazują, że takie państwa jak Włochy, Niemcy czy Hiszpania nie osiągnęły do dziś przedpandemicznego poziomu. Chciałbym zapytać, z czego wynika fakt, że państwa strefy euro są aż tak daleko w tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Piotr Patkowski. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o wpływ Funduszu Inwestycji Strategicznych, funduszu Polski Ład na wzrost PKB, to do tej pory odbyły się dwie edycje, zostały rozstrzygnięte dwie edycje z tym związane i edycja związana z funduszem wsparcia dla gmin, w których znajdowały się PGR-y.

Możemy szacować wstępnie wpływ tego programu na PKB, biorąc pod uwagę następującą metodologię, czyli uwzględniając, jak PKB by się kształtowało, gdyby te środki nie znalazły się w budżetach samorządów i nie zostały wydane na inwestycje. Patrząc na to już szczegółowo, warto zauważyć, że główne inwestycje samorządów będą w roku 2023 r. i w latach kolejnych, biorąc pod uwagę okres, który jest potrzebny samorządom od przyznania promes i rozstrzygnięcia konkursów do rozpoczęcia regularnych prac i dokonania w związku z tym płatności, które też będą miały wpływ na gospodarkę.

Proszę wziąć również pod uwagę, że szacunki uwzględniają te dwa nabory, które zostały rozstrzygnięte, i nabór PGR-owy, natomiast nie bierzemy jeszcze pod uwagę kolejnych naborów, które przecież mogą zostać ogłoszone i pewnie będą ogłoszone i rozstrzygnięte.

Warto także wziąć pod uwagę, że to będzie wpływało na PKB w bardzo istotnym jego aspekcie, a mianowicie we wzroście stopy inwestycji w relacji do PKB.

A więc te zamówienia będą trafiały przede wszystkim do małych bądź średnich polskich firm. Warto też zwrócić uwagę na to, że struktura jakościowa tych inwestycji będzie się głównie koncentrowała nie na dużych miastach, nie na metropoliach i nie będzie realizowana przez największe firmy, ale przez małe polskie mikroprzedsiębiorstwa, co powoduje, że ten wzrost PKB będzie podwójnie dobry jakościowo. Po pierwsze, będzie wpływał na wzrost stopy inwestycji, a po drugie, będzie realizowany przez mikro- i małe przedsiębiorstwa czy średnie z polskim kapitałem. Co do samego PKB innych państw członkowskich, to tak jak już tutaj pan poseł zwrócił słusznie uwagę, rzeczywiście Polska osiągnęła stopę PKB wyższą, niż to było przed COVID-em. Wiele państw, szczególnie zachodniej Europy, jeszcze tego nie osiągnęło. Wynika to z wielu przyczyn, m.in. tego, że w Polsce ten spadek PKB w roku 2020 był relatywnie niski w stosunku do takich państw jak Francja czy Belgia, ale też Polska zastosowała bardzo aktywną odpowiedź na sytuację gospodarczą związaną z kryzysem, z COVID-em, m.in. bardzo mocną politykę napędzającą i pobudzającą inwestycje i aktywną politykę prospołeczną, dzięki której obroniliśmy miejsca pracy i mamy jeden z trzech najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej, ale też mamy jedną z bardziej proaktywnych polityk gospodarczych wspomaganą środkami publicznymi, dzięki czemu ten wzrost PKB rzeczywiście jest jednym z najwyższych na terenie Unii Europejskiej, jednocześnie przy jednym z niższych deficytów, jeśli chodzi o rok 2021, konkretnie szósty najniższy deficyt na poziomie Unii Europejskiej. Czyli połączyliśmy aktywną politykę gospodarczą ze zrównoważonymi finansami publicznymi. Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Barbara Bartuś. Bardzo proszę. Dziękuję. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! To dodatkowe pytanie rozpocznę jednak od podziękowań. Od podziękowań za to, że te pieniądze na Polski Ład są przeznaczane, że ministerstwo jednak jest w tym, stoi na stanowisku, że te pieniądze idą na inwestycje, na inwestycje w takie regiony jak mój, daleko od ośrodków, centrów dużych miast, że ten zrównoważony rozwój jest przez to realizowany, że inwestycje są realizowane w moim powiecie gorlickim, na Sądecczyźnie, w miejscach, w których dawniej o takich pieniądzach samorządy w ogóle nie mogły marzyć. Panie Ministrze! Pytanie.

Jeszcze jedno. Analiza pod kątem inflacji, bo jeżeli jest podaż, jeżeli można tyle inwestycji realizować, są pieniądze, to i ceny idą w górę w przypadku tych inwestycji. Dziękuję bardzo. Ponownie odpowiedzi udziela podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Piotr Patkowski. Wysoka Izbo! Zacznę od kwestii ewentualnego wpływu na inflację programu Polski Ład - tutaj właściwie ten efekt powinien być pomijalny. Zwróćmy uwagę, że to są środki przeznaczane głównie na programy inwestycyjne, czyli wzmacniające także produktywność gospodarki, i w dłuższym, ale nie tylko w dłuższym, bo też w średnim okresie wyższa dynamika inwestycji, tak jak wspomniałem, to jest nawet 0,5 punktu procentowego w roku 2023 dodatkowego wygenerowanego wpływu i wzrostu gospodarczego, będzie zwiększała przede wszystkim możliwości podażowe gospodarki oraz obniżała jednostkowe koszty pracy, co powinno też obniżać presję na wzrost cen. Więc zwróćmy uwagę na to, o czym też mówiłem w pierwszej części wystąpienia, na ten jakościowy, bardzo jakościowy wpływ programu Polski Ład na poziom inwestycji. Jeśli chodzi o wpływ na same gminy i samorządy, to zwróćmy uwagę, że często one trafiają - ale nie tylko, bo praktycznie każda gmina, niezależnie czy mała, czy największa metropolia złożyła poprawny wniosek, otrzymała te środki - zwróćmy uwagę, że one mają szczególną wartość właśnie w tych gminach, które ze względu na często bardzo niskie dochody bieżące nie mają tej możliwości wygenerowania przestrzeni finansowej na pobudzanie inwestycji. Więc o ile często w średnich i większych miejscowościach jest to po prostu dodatkowa przestrzeń na kolejne inwestycje, o tyle w najmniejszych miejscowościach jest to jedyna szansa na to, żeby poszczególne inwestycje mogły być zrealizowane, w związku z czym są to też jedyne szanse na to, żeby przedsiębiorstwa, które znajdują się na tych terenach, mogły realizować przedsięwzięcia inwestycyjne na tym terenie. Dość trudno jest oszacować, jaka jest skala takich gmin i jaki jest tego dokładny poziom, natomiast można spokojnie powiedzieć, że w zdecydowanej większości gmin wiejskich jest to program, który nie tylko rozszerza bazę potencjalnych inwestycji przez nie realizowanych, ale przede wszystkim daje często pierwszą szansę, żeby inwestycje, które do tej pory były tylko planowane, mogły się rzeczywiście odbyć. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do następnego pytania. Jest ono kierowane do ministra spraw zagranicznych, a zadają je posłowie Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk i grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Jako pierwszy pan poseł Sławomir Nitras. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Panie ministrze. Ja przepraszam, bo nie dostrzegłem pana. Sprawa jest niezmiernie poważna. Jak wiemy, w przyszłym tygodniu od wtorku będzie szczyt NATO w Madrycie i będą poruszane dwie najważniejsze kwestie, czyli kwestia obecności, zwiększenia obecności wojsk NATO-wskich na wschodniej flance NATO i budowa nowej koncepcji strategicznej sojuszu, w której, jak rozumiem, wschodnia flanka NATO ma być kwestią najistotniejszą, czyli wyzwaniem najpoważniejszym. Myślę, że w tej kwestii w Polsce nie powinno być jakiegokolwiek sporu, tzn. od lewa do prawa w Polsce wszyscy powinni wspierać w tej materii działania rządu w Madrycie i dobrze by było, żeby nie było wątpliwości co do tego, jakie są zamierzenia rządu. Dobrze by było, żeby te kwestie nie budziły jakichkolwiek wątpliwości w Polsce. I chciałbym, panie ministrze, żeby pan bardzo precyzyjnie odpowiedział na moje pytanie, a nie mówił generalnie o strategii. Powołuję się na wypowiedź pana kolegi, ministra Jabłońskiego, wiceministra spraw zagranicznych, z 5 czerwca z ˝Rzeczpospolitej˝ Zapytany przez dziennikarza, to jest cytat, czy szczyt NATO pod koniec czerwca powinien podjąć decyzję o rozmieszczeniu amerykańskiej broni jądrowej na flance wschodniej w Polsce, pan minister Jabłoński odpowiada: Zdecydowanie warto o tym rozmawiać. Rosja ma na wyposażeniu swoich sił zbrojnych środki masowego rażenia, nie ma więc żadnego powodu, aby państwa najbardziej zagrożone takim scenariuszem nie posiadały symetrycznych środków. Moje pytanie, panie ministrze, brzmi: Z czym państwo jedziecie do Madrytu? Czy jest jakiś pomysł, urodził się w rządzie, na obecność broni masowego rażenia, broni jądrowej w Polsce? Czy to jest stanowisko przedyskutowane z kimś?

Dziękuję. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Marcin Przydacz. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście to będzie bardzo ważny szczyt w Madrycie. To będzie pierwszy formalny szczyt NATO-wski, który powinien podejmować konkretne decyzje dotyczące także adaptacji Sojuszu wobec sytuacji, która wydarzyła się na Ukrainie. Ma pan rację, panie pośle, wskazując, że głównym efektem szczytu będzie przyjęcie nowej koncepcji strategicznej.

Koncepcja strategiczna będzie publicznym dokumentem wskazującym główne kierunki działania, rozwoju NATO w perspektywie następnych kilku lat. Dla nas priorytetem jest, aby nowa koncepcja odzwierciedlała diametralną zmianę bezpieczeństwa euroatlantyckiego, jaka nastąpiła w wyniku pełnoskalowej agresji Rosji. Zabiegamy o to, aby odpowiednio opisać zagrożenie, jakim jest Rosja, a także kierunki odpowiedzi Sojuszu na jej działania. Oczekujemy, i to jest częściowa odpowiedź na pańskie pytanie, że obrona kolektywna zostanie w koncepcji wskazana jako absolutnie kluczowe zadanie Sojuszu. W związku z tym konieczne będzie długoterminowe wzmacnianie działań z zakresu odstraszania i obrony NATO, w tym w szczególności na wschodniej flance Sojuszu. Staramy się jednocześnie urealnić podejście do ewentualnych kontaktów NATO z Rosją w przyszłości. W nowej koncepcji strategicznej po raz pierwszy znajdą się także odniesienia do wyzwań stawianych przez Chiny. Dla Polski istotne jest, aby problematyka chińska jednak nie dominowała w działaniach NATO nad największym i bezpośrednim zagrożeniem dla obszaru euroatlantyckiego, jakim jest Rosja. Drugim elementem, równie ważnym, dotyczącym koncepcji strategicznej będzie pakiet szczegółowych decyzji dotyczących długoterminowego wzmacniania, odstraszania i obrony.

Jeśli chodzi o broń masowego rażenia, to są to oczywiście decyzje sojusznicze, ale są to także decyzje podejmowane w kanałach bilateralnych, w rozmowach amerykańskich.

Natomiast to, co jest dla nas kluczowe, i to podkreślę, to wzmacnianie obecności sojuszniczej, wzmacnianie obecności amerykańskiej na wschodniej flance NATO, nie tylko w Polsce, ale także w państwach bałtyckich, tych, które są najbardziej zagrożone, również w państwach na południu wschodniej flanki. To jest dla nas absolutnym priorytetem.

To wsparcie jest realizowane przede wszystkim w kontaktach dwustronnych.

Dodatkowo oczywiście odbędzie się dyskusja nad wsparciem innych naszych partnerów, Gruzji, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny. Będziemy rozmawiać czy pan prezydent reprezentujący Polskę będzie rozmawiał także z państwami like-minded tzw. wolnego świata - czyli przedstawiciele Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei Południowej - o wyzwaniach już natury globalnej. Będzie oczywiście także prowadzona dyskusja na temat rozszerzenia NATO. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że Finlandia i Szwecja zadeklarowały gotowość i chęć wejścia w ramy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja będzie trwała, mamy nadzieję, że konkluzywnie zakończy się w perspektywie przyszłych miesięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę. Panie Marszałku!

Wiceminister spraw zagranicznych mówi: warto rozmawiać. Więc chciałbym zapytać, czy może najpierw warto by było też porozmawiać z Polakami, bo mi się wydaje, że taka dyskusja w Polsce się nie odbyła, a ona w tym przypadku jest bardzo konieczna. Pan dzisiaj mówi wprost, że na pewnym etapie, że być może. Znaczy, każdy, kto nas dzisiaj słucha, może mieć ewidentnie wrażenie, że pan po prostu kręci. Ja bym chciał wiedzieć, jakie jest stanowisko rządu. Czy rząd zabiega o to, żeby w Polsce była broń masowego rażenia, bo takie stanowisko musi być uzgodnione nie tylko z Wysoką Izbą, ale przede wszystkim z Polakami. My mamy różne wątpliwości i bardzo ograniczone zaufanie do państwa. Mamy pewne zastrzeżenia i cała Polska powinna mieć te zastrzeżenia.

Jak czytamy, jego sklep z paletkami i błazenkami nazywał się ˝Idolek˝ Największa w NATO fabryka trotylu. Więc wszystkie pytania, które tu padają, mają głębokie uzasadnienie w tym, co już za waszych czasów przeżyliśmy. Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Marcin Przydacz. Bardzo dziękuję. Miałem nadzieję na poważną dyskusję, taką, jaką proponował pan poseł Nitras. Jeśli chodzi o obecność amerykańską, panie pośle, to nie wiem, czy akurat pańska opcja polityczna ma jakikolwiek mandat do dyskutowania o obecności, o odstraszaniu. To 2016 r., to szczyt w Warszawie, to zabiegi prezydenta Dudy i rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do obecności NATO-wskiej w Polsce. Coś, co nie udawało się przez kilkanaście lat, stało się faktem po 2016 r. Tysiące żołnierzy sojuszniczych przyjechało do Polski. Dziś jesteśmy dużo bardziej bezpieczni, mając wojnę - tak naprawdę za granicami naszego państwa - poprzez obecność sojuszniczą amerykańską, rozbudowywaną także i za czasów kontaktów prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem. Dziś rozmawiamy z prezydentem Bidenem o zwiększeniu tej obecności w ramach sił konwencjonalnych, w ramach polityki odstraszania. Ten parasol ochronny sojuszników może być realizowany niekoniecznie, panie pośle, poprzez obecność na danym terytorium. Jasne jest, że naszym przeciwnikiem, i to w koncepcji strategicznej będzie wskazane, jest Rosja. Rosja, która jest również posiadaczem broni masowego rażenia. I o tym mówię, że warto rozmawiać na temat tego, jak potencjalnie może Rosja zachować się w przyszłości i jak będzie reagował Sojusz. Obecność sojusznicza w naturalny sposób będzie wzmacniać naszą obronę. A rozmawiać warto nawet z panem posłem o tej tematyce, tak żebyśmy rzeczywiście dobrze się rozumieli.

Bardzo dziękuję za tę możliwość. Chciałbym tylko przypomnieć, że historia Rzeczypospolitej nie zaczęła się w roku 2015 i żołnierze amerykańscy byli tu już wcześniej. Byli za ministra Klicha, za poprzedniego prezydenta. Więc chciałbym, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że nasze rządy, to, co dzieje się w naszym kraju, to pewna sztafeta. Akurat wszystkie siły polityczne - i to wielka zasługa w ogóle całej klasy politycznej - zabiegały o to, żeby wojska amerykańskie i wojska NATO-wskie były w Polsce.

Jako pierwszy pan poseł Robert Obaz. Bardzo proszę.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polski Ład i jego rozwiązania są dobre dla każdego z nas, szczególnie dla tych najmniej zarabiających. Przy tej inflacji, która jest, każda złotówka więcej w portfelu Polaków to ważna rzecz.

Usługi, szczególnie jeśli chodzi o usługi publiczne, organizacja transportu, edukacji - te wszystkie rzeczy kosztują ogromnie dużo. Na ostatnim posiedzeniu komisji słyszeliśmy, że rząd nie finansuje edukacji, tylko przyznaje subwencję, a resztę musi zrobić samorząd. Podobne subwencje są zapowiadane do inwestycji, ale to tylko dodatek. Więc pytanie, jakie się nasuwa, to jak rząd zamierza zrekompensować samorządom ubytki w podatkach.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przede wszystkim chciałbym zacząć od wyników finansowych za rok 2021. Dla jednostek samorządu terytorialnego te wyniki były wyjątkowo dobre, były to dane najlepsze, jeżeli chodzi historię jednostek samorządu terytorialnego.

To były historycznie najlepsze wyniki budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego obecnie otrzymują równe udziały w podatkach dochodowych co miesiąc i tak będzie również po 1 lipca, czyli w tym roku jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od zmian ustawowych w każdym miesiącu do końca roku będą miały takie same wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie uzupełnienia ubytków z tytułu obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych już w 2021 r. został wprowadzony mechanizm zabezpieczający jednostki samorządu terytorialnego przed utratą tych ubytków, a mianowicie wprowadzono pojęcie kwoty referencyjnej waloryzowanej nominalnym PKB i do tej kwoty referencyjnej CIT-u i PIT-u. Jeżeli ta kwota referencyjna okaże się wyższa niż to, co wynika z prognoz budżetowych, to w budżecie państwa będzie musiała się znaleźć odpowiednia część subwencji ogólnej, czyli subwencja rozwojowa, którą jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać na podstawie algorytmu opartego w głównej mierze o liczbę ludności. Niezależnie od tego zwracam również uwagę na dużą kwotę środków przekazywanych z funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład - to już w zakresie rozstrzygniętych przetargów kwota ponad 53 mld zł, więc myślę, że środków dla jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza w obszarze inwestycyjnym, jest naprawdę dużo.

Tam również zapadły decyzje, że wraz ze stroną samorządową będziemy wypracowywać rozwiązania legislacyjne, które umożliwią elastyczną politykę budżetową jednostek samorządu terytorialnego jeszcze w tym roku, by sprostać wyzwaniom wzrostu cen usług komunalnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Polskie samorządy cały czas szukają sposobu, jak sprawnie, zgodnie z prawem i przede wszystkim bezpiecznie wypełniać swoje obowiązki, ale też móc realizować wszystkie zadania, które zostały im powierzone, bo niezwykle ważne jest, by miały za co je realizować. Niestety ten udział w PIT i CIT nie jest wystarczający. Lewica złożyła konkretne propozycje dotyczące zwiększenia udziałów PIT i CIT dla samorządów, ponieważ takie mamy postulaty ze strony samorządowej i takie też jest oczekiwanie w stosunku do strony rządowej, żeby zwiększyć ten udział, ponieważ samorządy mają obecnie oczekiwania od nauczycieli, muszą też zadbać o kadrę medyczną w szpitalach, gdzie obecnie pielęgniarki proszą o to, żeby zwiększać im udział w zarobkach, również służby niemedyczne tego oczekują. Dziękuję. Ponownie na pytania odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Sebastian Skuza. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tak jak przed chwilą wyjaśniałem, w miejsce ubytków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wejdzie część subwencji ogólnej, tzw. subwencja równoważąca, która będzie dzielona algorytmicznie na podstawie obiektywnych kryteriów. Co do zwiększenia udziałów w podatku od osób fizycznych, to zwracam uwagę tutaj na rzecz następującą, że dla niektórych jednostek samorządu terytorialnego takie rozwiązanie może nie przynieść efektów. Z jakie względu?

Tam baza podatkowa z tytułu podatku od osób fizycznych zmniejszy się diametralnie. Jeden z wójtów przedstawił sytuację w swojej jednostce samorządu terytorialnego i powiedział, że w jego gminie za rok 2021 drugi próg podatkowy przekroczyło tylko łącznie z nim 27 osób, więc zwiększenie udziałów PIT w takiej gminie po znacznej redukcji bazy nic nie da. Dlatego zostało wprowadzone narzędzie subwencji rozwojowej, która równomiernie będzie uzupełniać ubytki z tytułu obniżenia stawek podatkowych i podwyższenia kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konkluzji chciałbym dodać takie pytanie: Czym lepiej dysponować: 1% od miliardów czy 100% od niewielkiej bazy lub nawet od zera? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.

Jako pierwsi pytanie zadają Waldemar Andzel i Jarosław Krajewski. Panie Marszałku! Polacy w trakcie pandemii bardzo ochoczo zaczęli korzystać z mobilnych i elektronicznych rozwiązań dla obywateli. Tymczasem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o projekcie ustawy o aplikacji mObywatel i o utworzeniu cyfrowego portfela na dokumenty. Bardzo proszę o przedstawienie szczegółów proponowanych zmian, od kiedy miałyby one wejść w życie i ilu Polaków korzysta obecnie z aplikacji mObywatel. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Jarosław Krajewski. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kontynuując te pytania, które przedstawił pan poseł Waldemar Andzel, zwracam się do pana ministra z takim konkretnym pytaniem. W związku z tym, że jak przepisy proponowane przez kancelarię premiera wejdą w życie, będziemy mogli mówić o zrównaniu pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w ramach aplikacji mObywatel z tymi dokumentami w wersji tradycyjnej, to będzie to duże ułatwienie dla milionów Polaków. Chciałbym w związku z powyższym zapytać pana ministra, czy planowana jest kampania informacyjna w tej sprawie, która będzie popularyzowała aplikację mObywatel i która będzie prowadziła nas do jak największego upowszechnienia tej aplikacji, możliwości korzystania z niej, ponieważ tak jak wspomniałem, ona zdecydowanie ułatwi życie milionom Polaków. Jeżeli tak, to jakie środki będą przekazane na tę akcję informacyjną, kampanię społeczną? Czy planowana jest również rola mediów publicznych w popularyzacji bardzo dobrych rozwiązań dla obywateli? Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Natomiast uznaliśmy jako osoby odpowiedzialne za kwestię cyfryzacji w naszym państwie, że jeśli proponujemy Polakom tak popularne rozwiązanie, jakim jest aplikacja mObywatel, która przecież zawiera w sobie szerokie komponenty, również te umożliwiające w wielu miejscach potwierdzanie własnej tożsamości, jak chociażby komponent mObywatel, mPrawo jazdy, dostępne są legitymacje studenckie, uczniowskie, które potwierdzają naszą tożsamość, to chcielibyśmy, żeby rzeczywiście obywatele, którzy korzystają na co dzień z tej aplikacji, mogli wszędzie na równi z dowodem osobistym tą przecież bezpieczną aplikacją potwierdzać swoją tożsamość w każdej sytuacji w naszym kraju.

Pierwsza kluczowa zmiana - aplikacja mObywatel będzie traktowana w polskim państwie na równi z dowodem osobistym, wyłączając kwestie przekraczania granic. Druga niezwykle ważna zmiana to jest również wprowadzenie transakcyjności w aplikacji mObywatel, za pośrednictwem której obywatele będą mogli płacić za usługi publiczne, czyli jeśli w danym urzędzie obywatel załatwia daną sprawę i musi uiścić opłatę, będzie mógł to spokojnie zrobić z poziomu aplikacji, z poziomu telefonu, nie będzie musiał szukać oddzielnie kasy, żeby uiścić opłatę, tylko będzie mógł to robić za pośrednictwem mObywatela. Sama ustawa, która zrównuje prawnie aplikację z dowodami osobistymi, mamy nadzieję, że wejdzie w życie jeszcze w tym roku, pod koniec tego roku. Taki jest nasz cel obecnie.

Będziemy tam dodawać kolejne dokumenty, jak chociażby mLegitymacja emeryta i rencisty. Mamy już mKartę Dużej Rodziny, z czego korzysta kilkaset tysięcy Polaków, mamy też mLegitymację szkolną, studencką, mamy również dokumenty dla kierowców: mPojazd, mPrawo jazdy.

Odpowiadam na pytanie pana posła Jarosława Krajewskiego. To jest bardzo cenne pytanie. Absolutnie musimy rozpocząć dużą kampanię informacyjną. Takie plany oczywiście są, panie pośle.

Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za tę wyczerpującą wypowiedź. Aplikacja mObywatel jest jedną z kilkuset dostępnych e-usług publicznych zlokalizowanych na różnych platformach rządowych. Administracja publiczna w Polsce wciąż przechodzi dynamiczną transformację. Proszę o udzielenie informacji, jak rozwijają się pozostałe usługi zlokalizowane na portalach obywatel.gov.pl i biznes.gov.pl. O ile wzrosła liczba użytkowników tych portali od początku pandemii COVID-19? Które województwa, ewentualnie miasta, powiaty, dominują, jeśli idzie o zainteresowanie mieszkańców e-usługami publicznymi? Dziękuję bardzo. Ponownie odpowiedzi udziela sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pan Adam Andruszkiewicz. Szanowny Panie Marszałku! Panie Pośle!

Temu służy chociażby profil zaufany, z którego na co dzień korzysta 14 mln Polaków, załatwiając wiele swoich spraw urzędowych.

Takie propozycje z pewnością będą realizowane. Jeśli chodzi o konkretne dane, o które pytał pan poseł, szczegółowo odpowiemy panu posłowi na to pytanie na piśmie, ponieważ to było takie szczegółowe pytanie, nawet do poziomu powiatów.

Średnia z miesiąca to jest ponad 15 mln odsłon na portalu, co wydaje się dość dobrym wynikiem. To jest cały szereg projektów. Mam nadzieję, że szanowni państwo będziecie te projekty wspierać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że Polska naprawdę staje się państwem cyfrowym. Osiągamy coraz lepsze wyniki w wielu międzynarodowych rankingach. To nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że to będzie przez państwa jak najbardziej docenione, ponieważ to hasło: nowoczesna Polska, innowacyjna Polska, szeroki, bezpłatny dostęp do Internetu w szkołach, rekordowe zakupy, jeśli chodzi o sprzęt dla uczniów w szkołach do nauki zdalnej, wyposażenie samorządów w nowoczesne narzędzie innowacyjne - to się dzieje. Te nakłady pod rządami Prawa i Sprawiedliwości są nieporównywalnie większe, jeśli chodzi o porównanie z opozycją, z czasami Platformy Obywatelskiej, kiedy te nakłady były, można powiedzieć, tylko symboliczne. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, jak budować innowacyjne, nowoczesne, przyjazne dla naszego obywatela państwo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego pytania. Panie posłanki Monika Wielichowska i Joanna Jaśkowiak, a także grupa pań posłanek z Koalicji Obywatelskiej kierują pytanie do ministra aktywów państwowych. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Są w Polsce spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, które do celów ogrzewania i podgrzewania wody nabywają energię cieplną od przedsiębiorstw energetycznych, w których paliwem do produkcji energii cieplnej jest gaz ziemny, a które zostały wykluczone z rekompensat, bo rząd wdrożył ustawę niesprawiedliwą społecznie, wadliwą i przede wszystkim dziurawą. Mówiłam o tym z tego miejsca dokładnie 4 miesiące temu. Za mną są złożone interpelacje, spotkanie z prezesem URE i udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. 25 lutego br. w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska do laski marszałkowskiej złożyłam projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Nowelizacja zrównoważy prawo do rekompensat, do ciepłego mieszkania, umożliwi pomoc wykluczonym ze wsparcia gospodarstwom domowym. To bardzo oczekiwana nowelizacja prawa przez tysiące mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w całej Polsce. 23 marca marszałek Sejmu skierowała ten poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, zawarty w druku nr 2111, do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych do pierwszego czytania. Projekt do dziś leży w komisyjnej zamrażarce. Minęły znowu 4 miesiące. Na co, panie ministrze, czekacie? Projekt jest gotowy, więc korzystajcie. Nie czekajcie na ludzkie dramaty.

Ona zrównoważy prawa wszystkich obywateli. Co pan minister zrobił, by projekt był procedowany? Dlaczego rząd (Dzwonek) nie przedstawił swoich rozwiązań, jeśli nie chcecie korzystać z rozwiązań przygotowanych przez nas? Dziękuję. Dziękuję. Na pytanie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan Maciej Małecki. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd od początku kryzysu energetycznego wywołanego przez Władimira Putina, pomimo kompletnie naiwnej, oderwanej od rzeczywistości polityki europejskich elit, prowadzi działania ograniczające wzrost cen energii.

Wsparcie tym dodatkiem obejmuje blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. To jest wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin, które najmocniej dotknął wzrost cen energii. 29 stycznia weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Czyli cena rynkowa jest trzykrotnie wyższa niż ta, którą płacą odbiorcy indywidualni w domach jednorodzinnych, we wspólnotach, w spółdzielniach mieszkaniowych i odbiorcy wrażliwi - szpitale, szkoły, przedszkola, hospicja, ochotnicze straże pożarne itd.

Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że przy okazji tej ustawy można było objąć ochroną odbiorców wykorzystujących gaz do celów bytowych: gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspomnianych przeze mnie odbiorców wrażliwych. Klucz do rozwiązania tego problemu leży nie w Warszawie, ale w Brukseli. To przepisy unijne nie pozwalają na rozszerzenie wsparcia polegającego na dopłatach do cen gazu dla przedsiębiorców takich jak ciepłownie, które produkują ciepło komercyjnie.

Te przepisy unijne nie pozwalają na objęcie ochroną taryfową prezesa URE przedsiębiorców produkujących ciepło. Kwestia taryf dla przedsiębiorców wykorzystujących gaz do produkcji ciepła została poruszona też w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 września 2015 r. w sprawie Komisja przeciw Polsce, który doprowadził do konieczności przyjęcia nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne. Wtedy do polskiego prawa zaimplementowano przepisy dyrektywy gazowej liberalizujące rynek gazu w Polsce w zakresie taryfowania przedsiębiorców energetycznych działających na rynku paliw gazowych. Te zmiany zniosły nadzór prezesa URE nad taryfami na sprzedaż gazu do odbiorców hurtowych oraz na sprzedaż gazu do odbiorców końcowych, którzy dokonują zakupu paliwa w punkcie wirtualnym lub w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. 1 października 2017 r. na mocy tych przepisów zniesiono zatwierdzanie przez prezesa URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.

Przestańcie awanturować się w polskim Sejmie i załatwcie to w Brukseli. Bo tam rządzicie, tam jesteście większością i to jest miejsce, które może odblokować obniżenie cen paliw, cen ciepła dla odbiorców nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. Dodatkowe. Niech pani nie krzyczy, na Boga, no!

Pani poseł, bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wczoraj Sejm zajmował się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Z danych GUS-u z 2020 r. wynika, że tych gospodarstw jest 5 mln. Chciałam zapytać pana ministra, co proponuje pan pozostałym 3,5 mln gospodarstw rolnych korzystających z węgla dla celów grzewczych. Co proponuje pan, panie ministrze, osobom korzystającym np. z oleju opałowego? Bo inaczej tym pozostałym osobom zostanie tylko chrust, a może go braknąć w lesie. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Na tym posiedzeniu Sejmu jest procedowana ustawa obniżająca cenę węgla dla odbiorców indywidualnych i na cele bytowe we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt przewiduje rekompensaty dla sprzedawców, którzy sprzedawali paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny, brykiet, pellet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego po cenie nie wyższej niż 966,60 zł brutto za tonę dla gospodarstw domowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przyznania rekompensaty jest także zarejestrowanie na terytorium Polski przedsiębiorstwa korzystającego z tej rekompensaty. Rekompensata ma wynosić nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego na jedno gospodarstwo domowe.

Pierwsza sprawa to rok 2014 i premier Ewa Kopacz, która. w Radzie Europejskiej zgodziła się na zniesienie jednomyślności państw członkowskich w sprawach klimatycznych.

To hasło ˝drożyzna˝ może pani sobie powiesić w lustrze. bo dzisiaj za drożyznę w Polsce odpowiada Władimir Putin, któremu chcieliście sprzedać Lotos, od którego chcieliście brać gaz do roku 2037. i z którym wasz lider Donald Tusk spacerował prawie pod rękę po sopockim molo.

Wzrosty cen energii elektrycznej, wzrosty cen ciepła, wzrosty cen gazu, które obejmują całą Europę, wynikają z agresji Putina na Ukrainę i z kompletnego oderwania od rzeczywistości europejskich elit, które nie zrobiły nic. żeby zatrzymać ten pochód Putina, które wolały z nim robić interesy takie jak Nord Stream 1, Nord Stream 2. Kiedy Polska szła drogą śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził konsekwentną, ambitną, niezależną politykę klimatyczną, żeby uwolnić nas od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu, wasi patroni polityczni z Europejskiej Partii Ludowej, tacy jak Angela Merkel, ubijali biznesy z Putinem. Dzisiaj trzeba być po prostu skrajnie nikczemnym, żeby atakować polski rząd za inflację wywołaną przez Putina i waszą naiwność jako Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Panie posłanki Barbara Dziuk i Anna Dąbrowska-Banaszek mają pytania do ministra edukacji i nauki. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Był to bardzo trudny czas, kiedy musieliśmy zmierzyć się z gigantycznym problemem społecznym na całym świecie. W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich członków społeczności edukacyjnej, jak i naukowej, zapowiedziało utworzenie nowego portalu: edukacja.gov.pl. To kolejny krok w kierunku cyfrowej szkoły przyszłości. To taki cyfrowy tornister, który nic nie waży.

Moje pytania do pana ministra są następujące: Jak wziąć udział w konsultacjach? Kogo one dotyczą? Jaka jest rola i cel portalu? Dziękuję. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pan Tomasz Rzymkowski. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Odpowiadam na pytania pani poseł. W konsultacjach można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej edukacja.gov.pl. Jeśli chodzi o to, do kogo je adresujemy, kogo mają dotyczyć te konsultacje, to odpowiadam, że konsultacje dotyczą wszystkich uczestników życia edukacyjnego i naukowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oczywiście nauczycieli szkolnych i nauczycieli akademickich, uczniów, studentów, rodziców dzieci szkolnych, dyrektorów szkół, rektorów uczelni wyższych, kuratorów oświaty i innych pracowników oświaty i nauki.

Edukacja.gov.pl ma służyć podniesieniu świadomości w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego uczniów, nauczycieli i wszystkich uczestników życia edukacyjnego w Polsce. Ponadto planowane są funkcjonalności dotyczące ułatwienia kwestii administracyjnych w szkołach i uczelniach wyższych, certyfikacji kompetencji, diagnozy kompetencji i innych umiejętności.

Dodatkowe pytanie zada pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Każda forma rozszerzenia, ułatwienia edukacji jest bardzo potrzebna. Widzimy to teraz. Utworzona platforma m.in. skraca czas potrzebny do kontaktu. To bardzo dobre uzupełnienie dotychczasowej oferty edukacyjnej. Ponad 11 tys. podmiotów, szkół już z tego korzysta. To możliwość zwiększenia praktycznych umiejętności uczniów. Moje pytanie dotyczy kolejnych planowanych działań. Czy są już przewidywane kolejne nowe aktywności na podstawie tego, co już widzimy w ankietach? Ponownie odpowie pan sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, rzeczywiście program ˝Laboratoria przyszłości˝ okazał się wielkim sukcesem.

Te środki trafiły tam na początku tego roku.

Jeśli nie skorzystały, to jest już, jakby to powiedzieć, ich sprawa, bo nie wnioskowali o przyznanie tych środków.

Jeśli chodzi o inne formy wsparcia, to niewątpliwie wielkim sukcesem zakończył się nabór.

Dzięki temu często po raz pierwszy polska młodzież i polskie dzieci mają okazję zobaczyć ważne miejsca z punktu widzenia naszej historii, tożsamości narodowej, ale również ważne miejsca z punktu widzenia nauki, edukacji, z punktu widzenia poszerzania swoich umiejętności.

Dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do następnego pytania. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Andrzej Gawron. Panie Marszałku! 14 czerwca przez przekop Mierzei Wiślanej przepłynęła pierwsza jednostka pływająca. Inwestycja jest już na ukończeniu. W najbliższym czasie kanał żeglugowy połączy port w Elblągu z Zatoką Gdańską. To szansa na rozwój gospodarczy regionu, to szansa na zwiększony ruch turystyczny, a jednocześnie to ogromne przedsięwzięcie, jedno ze strategicznych osiągnięć rządu, które znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa Polski i umocni naszą suwerenność. Widać to szczególnie teraz, gdy na Ukrainie toczy się wojna, a polskie jednostki muszą każdorazowo uzyskiwać zgodę na przepłynięcie Cieśniny Pilawskiej. Przy zaostrzeniu tego konfliktu mogłoby się okazać, że Rosja zablokuje nam Zalew Wiślany. I pomimo tak oczywistych faktów zdarza się, że opozycja poddaje krytyce tę inwestycję. Proszę więc pana ministra o udzielenie informacji, jakie parametry charakteryzują sam przekop Mierzei Wiślanej, ale również tor wodny do portu w Elblągu, a co za tym idzie, jakie jednostki będą mogły korzystać z tego nowego szlaku żeglugowego i jakich korzyści gospodarczych, turystycznych możemy się spodziewać po całkowitym zakończeniu inwestycji. Resztę czasu wykorzystuje pan poseł Aleksander Mrówczyński, również Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sądzę, jestem przekonany, że totalnej opozycji nie trzeba przekonywać - myślę, że nie trzeba, wierzę w to bardzo - co do sensu tego, co robimy, czyli do przekopu Mierzei Wiślanej. Jeśli tak, to tylko powiem, że na pewno wie ona o tym, że dwa plus dwa jest cztery, ale w tym przypadku to będzie pięć, a niekiedy 10. To jest efekt synergii. Panie Ministrze! Proszę powiedzieć tym wszystkim niedowiarkom, proszę przekazać, że 17 września rzeczywiście będziemy mieli wielki dzień i w tym dniu będzie otwarcie przekopu, za co serdecznie dziękuję panu prezesowi, panu ministrowi i wszystkim zaangażowanym. Bardzo dziękuję. Odpowiedzi udziela sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Marek Gróbarczyk. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim na wstępie trzeba opowiedzieć o całym procesie związanym z budową kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Została ona przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana do realizacji. Niestety przez 8 lat u naszych poprzedników nie działo się za wiele w tej materii.

Przy tej samej okazji jedna z pań senator Platformy Obywatelskiej ufundowała pomnik w Kątach Rybackich, przypominający o tym, jak to przekop jest niezbędny, konieczny do realizacji.

Dla nas było rzeczą oczywistą, że realizacja tej inwestycji musi mieć swoją kontynuację. W związku z tym w 2016 r. został przygotowany nowy program wieloletni, który wskazywał konieczność realizacji tej inwestycji i określał środki na jej realizację.

Obejmuje on przede wszystkim budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną, budowę toru żeglugowego przez Zalew Wiślany, budowę i modernizację toru wodnego na rzece Elbląg, budowę mostu w Nowakowie oraz doprowadzenie toru żeglugowego do portu w Elblągu, a dodatkowo będzie budowa sztucznej wyspy i budowa pogłębiarki, która będzie utrzymywała ten tor w należytej kondycji.

Oczywiście zakładamy, że będzie to przede wszystkim port wspierający porty trójmiejskie. W obecnej sytuacji, kiedy mamy ogromne zapotrzebowanie na nowe tereny, jest to doskonała okazja do uruchomienia terenów portowych, przygotowania nowych terenów portowych. W tym zakresie port w Gdańsku prowadzi bardzo intensywne analizy co do inwestycji na tym terenie.

Na pewno będziemy potrzebowali znacznych ilości nowych powierzchni magazynowych i składowych, w związku z tym również dopuszczamy czy zakładamy możliwość budowy nowego terminala w okolicy Tolkmicka, który będzie właśnie pełnił rolę przede wszystkim terminala masowego.

Będzie to przedsięwzięcie w 100% biznesowe, w związku z tym port w Gdańsku przygotowuje rozwiązania. Tutaj zakładamy, że będzie to zwiększenie i zabezpieczenie możliwości przerzutu oraz zaopatrzenia dla pododdziałów 16. Dywizji Zmechanizowanej właśnie z wykorzystaniem drogi morskiej, oczywiście nie mówiąc już o podstawowych elementach związanych ze skróceniem drogi wodnej czy generalnie otwarciem zalewu dla swobodnej żeglugi, dla nowych jednostek. Założenie, że Cieśnina Pilawska mogłaby być kiedyś wykorzystana, jest absolutnie błędne.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Szanowni Posłowie!

Pytanie brzmi: Czy ominięcie cieśniny przyczyni się, i w jakim stopniu, do zwiększenia naszej suwerenności, a tym samym bezpieczeństwa - jakie są tu wskaźniki i przewidywania - być może poprzez nienarażanie naszego kraju na zbędne i niebezpieczne spory, co może być przyczyną agresji ze strony Rosji? Bardzo proszę. Oczywiście tragedia na Ukrainie, która się dzieje, wskazuje na właściwy kierunek tej inwestycji.

A więc jest to rozwiązanie, które tworzy możliwości przekierowania ładunków z obszarów, które do tej pory nie były wykorzystywane. Pojawienie się zupełnie nowych grup towarowych i nowych operatorów jest niezwykle istotne dla rozwoju regionu, przede wszystkim dla rozwoju portu w Elblągu, ale tworzy też inne możliwości rozwojowe.

Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama, Grzegorz Gaża, Jerzy Paul i Bożena Borys-Szopa kierują pytanie do ministra zdrowia. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Pacjenci, a także lekarze pozytywnie oceniają dotychczasowe zmiany w zakresie cyfryzacji otrzymywanych recept oraz e-skierowań. W ślad za tym rozwiązaniem postulowane są kolejne, jak chociażby e-rejestracja do specjalistów. Proces elektronicznej rejestracji powinien umożliwić np. zapisanie się na wizytę do specjalisty kardiologa, na tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny. Dotychczas takiej możliwości jednak nie ma, co wielu pacjentom utrudnia cały proces mimo chęci skorzystania ze świadczenia. Pragnę zapytać, czy ministerstwo podjęło działania, których efektem będzie wprowadzenie usługi e-rejestracji do specjalisty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Maciej Miłkowski. Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest systemowe, kompleksowe pytanie dotyczące przyszłości i rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz wsparcia systemu ochrony zdrowia przez systemy informatyczne, które usprawniają świadczeniodawcom, ale w szczególności pacjentom cały proces leczenia. To kolejna rzecz oczekiwana przez pacjentów po sukcesie e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne, które są już standardem postępowania. Brakuje jednak istotnego elementu zapisania się na konkretne świadczenie zdrowotne i ta e-rejestracja jest bardzo oczekiwana. Faktycznie w Ministerstwie Zdrowia podpisane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 2 czerwca br. w zakresie przygotowania pilotażu odnośnie do elektronicznej centralnej rejestracji na niektóre świadczenia zdrowotne.

To jest porada kardiologiczna, poradnia kardiologiczna oraz dwa świadczenia kosztochłonne w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Ustaliliśmy, że pilotażem będzie objętych 20 podmiotów w dwóch regionach kraju.

Chcemy przetestować bardzo różnorodne techniki, podmioty małe do 500 świadczeń medycznych, jak również duże podmioty, które to realizują. Warunkiem uruchomienia tych ośrodków było posiadanie systemu do e-rejestracji przez te podmioty bądź deklaracja, że te szpitale, te podmioty lecznicze podepną się pod system informatyczny gabinet.gov.pl i całe koszty dostosowania systemu będą kosztami podmiotu.

Założenie jest takie, że to są świadczenia pierwszorazowe. Oczywiście w tomografii, w rezonansie właściwie zawsze to jest odrębny cel leczenia diagnostycznego w przypadku porady, później jest kontynuacja. Na razie kontynuacji nie będziemy obsługiwali, ale w ogóle celem jest przetestowanie, żeby wszedł ten system e-rejestracji centralnej, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje świadczeń zdrowotnych. Zarejestrowanie się do takiego podmiotu leczniczego będzie możliwe w trzech trybach.

Te funkcjonalności, które są testowane, to zapisanie się na wizytę, zarządzanie tymi slotami przez pacjentów, przez podmioty lecznicze, zapisanie się na listę osób oczekujących. Dodatkowe pytanie zada pan poseł Jarosław Gonciarz. Bardzo wyczerpująco odpowiedział pan na moje pytanie. Aby tradycji stało się zadość, chciałbym dopytać: Czy warunki techniczne do przeprowadzenia pilotażu na pewno będą spełnione? Czy po nowym roku, w przyszłym roku, gdybyśmy chcieli objąć szerszy zakres w kraju, również te warunki techniczne będą spełniane? Dziękuję. Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Maciej Miłkowski.

Przy okazji będzie testowane też kilka systemów informatycznych firm prywatnych, które normalnie dostarczają oprogramowanie na rynek.

14 tys. aptek zostało podłączonych w szybkim czasie.

Jak państwo widzą, ten pilotaż i w ogóle cała metodologia przygotowywania projektów centrum zdrowia są takie, że najpierw po cichu, spokojnie wszystko jest testowane.

Przechodzimy do kolejnego pytania. Posłowie Barbara Nowacka, Paweł Poncyljusz i grupa posłów z Koalicji Obywatelskiej kierują pytanie do prezesa Rady Ministrów. Jako Koalicja Obywatelska popieramy zmierzanie Europy do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej, jednak przyjęcie przez rząd PiS części kamieni milowych w ramach KPO wynika z potrzeby opanowania krytycznej sytuacji w Polsce, gdzie nawet własny elektorat oczekuje europejskich pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy. Część polityków obozu Zjednoczonej Prawicy uważa niektóre kamienie milowe za kapitulację wobec Komisji Europejskiej. Przykładem nieprzemyślanej polityki rządu PiS, opartej na zasadzie: jakoś to będzie, jest zgoda na wpisanie do KPO kamieni milowych dotyczących wprowadzenia od 2024 r. opłaty rejestracyjnej od samochodów spalinowych, a po 2 latach - podatku od samochodów spalinowych. Dowodem na to, że rząd nie wiedział, na co się zgadza, są kompromitujące tłumaczenia ministra Budy, że z tym podatkiem to jeszcze nic nie wiadomo, czy prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że to są jakieś bajki. Z tych pokrętnych wyjaśnień wynika, że rząd nie ma i nie miał w czasie negocjacji KPO pomysłu na podatek od samochodów spalinowych. A teraz jeszcze rząd przestraszył swój elektorat, który jeździ samochodami spalinowymi ze względu na pogarszającą się sytuację społeczno-gospodarczą - w czym największe zasługi mają funkcjonariusze PiS, panowie Morawiecki i Glapiński - i nie będzie mógł sobie pozwolić na zakup samochodu elektrycznego obciążonego dodatkowymi podatkami. Stąd pytanie: Jakie były założenia dotyczące stawek podatku od samochodów spalinowych w instrukcji negocjacyjnej przedstawicieli polskiego rządu w negocjacjach na temat KPO z Komisją Europejską? Drugie: Czy nie jest tak, że posiadacze aut spalinowych tymi podatkami zapłacą za budowę fabryki samochodów elektrycznych marki Izera, która ma kosztować co najmniej 5 mld zł? Polacy już zapłacili 70 mln zł za działalność spółki ElectroMobility Poland, która od kilku lat koncentruje się jedynie na opowiadaniu bajek - jak to mówił premier Kaczyński o polskim samochodzie elektrycznym Czy nowy podatek od samochodów spalinowych w KPO to jedyny ślad po tych obietnicach premiera Morawieckiego? Dziękuję bardzo. Ministrów odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan Ireneusz Zyska. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, dzięki któremu zostaną zrealizowane nowe inwestycje, zbudujemy innowacyjną gospodarkę, zwiększymy zatrudnienie. Środki finansowe z tego instrumentu zostaną przeznaczone również na rozwój gospodarczy, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację, zdrowie i - co niesłychanie ważne - rozwój nowoczesnej energetyki, w tym obszar elektromobilności, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, pojazdów wodorowych. Szanowni Państwo! Odpowiadając na pytanie grupy posłów reprezentowanych przez pana posła Pawła Poncyljusza, muszę powiedzieć, że nie było żadnych instrukcji negocjacyjnych, nie było założeń dotyczących wysokości podatków czy też opłat związanych z emisyjnością. Zapis dotyczący kamienia milowego jest bardzo szeroki i nie zobowiązuje do nakładania nowych obciążeń podatkowych zarówno w zakresie emisyjności pojazdów konwencjonalnych, na paliwa konwencjonalne, jak i z tytułu używania takich paliw. Wielokrotnie pan premier Mateusz Morawiecki, ale także inni przedstawiciele rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości informowali opinię publiczną o tym, że nie będziemy nakładać żadnych opłat związanych z użytkowaniem pojazdów konwencjonalnych. Polityka Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości to polityka zachęty, a nie polityka kar i obciążania społeczeństwa, szczególnie tych grup społecznych, których nie stać na to, aby dokonać zakupu urządzeń, jakimi są samochody elektryczne nowych technologii, które są jeszcze drogie, dlatego że każda technologia wchodząca na rynek to technologia relatywnie droga. Chciałbym też przypomnieć państwu posłom, którzy zadają to pytanie, że w ˝Polityce energetycznej Polski do 2040 r.˝ - to jest dokument strategiczny w zakresie miksu energetycznego, transformacji energetycznej w Polsce - wprowadziliśmy podstawowy filar tej polityki, jakim jest sprawiedliwa transformacja. Otóż nie możemy dopuścić do tego, żeby nastąpiło wykluczenie jakiejkolwiek grupy społecznej z tytułu transformacji energetycznej czy też szeroko rozumianej transformacji gospodarczej, która w tej chwili trwa. Nie możemy też doprowadzić do wykluczenia transportowego, wykluczenia komunikacyjnego. Wielu z Polaków użytkuje dzisiaj pojazdy, samochody z napędem konwencjonalnym, jest to zdecydowana większość polskiego społeczeństwa.

Tutaj chciałbym powiedzieć i przypomnieć, że w 2018 r. została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Akt ten zdefiniował ścieżkę budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa zawiera zachęty do zakupu pojazdów zeroemisyjnych m.in. poprzez zwolnienie z akcyzy i limit amortyzacji podwyższony dla pojazdów elektrycznych do 225 tys. zł.

Otóż, szanowni państwo, dzisiaj w Polsce obowiązują przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Samochody, których silniki mają większą pojemność, a tym samym emitują więcej szkodliwych substancji do środowiska, płacą wyższą stawkę podatku akcyzowego.

Panie Ministrze! To kiedy wy kłamiecie? Kłamiecie Komisji Europejskiej czy kłamiecie teraz z mównicy? Zapisaliście wyraźnie w kamieniach milowych, że będzie podatek. Teraz pan mówi: nie będzie podatku. Jak nie wypełnimy kamieni milowych, to pieniądze do ludzi nie trafią. A pan teraz nas informuje, że nie wypełni, i bałamutnie opowiada, że akcyza to nie jest podatek. To się nazywa podatek akcyzowy, panie ministrze, więc bardzo bym prosiła, żeby szanował pan powagę Sejmu i mówił prawdę. Zaplanowaliście podatek. Już dowiedzieliśmy się, że 1 mln samochodów nie ma, nie było i nie będzie. Zgadza się, też byliśmy o tym przekonani, chociaż wiemy, ile zapłacili za to podatnicy. Jak przeciwdziałacie wykluczeniu komunikacyjnemu? Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan Ireneusz Zyska. Wysoka Izbo! Opozycja może tylko i wyłącznie zakrzykiwać rzeczywistość. które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż, proszę państwa, 1 mln samochodów będzie na polskich drogach. Pani poseł, ja mam panią za kulturalną osobę, proszę mi wierzyć.

Dzięki temu polskie miasta zakontraktowały ponad 600 autobusów elektrycznych i blisko 150 autobusów z napędem wodorowym.

870 mln zł rząd przeznaczył na ten cel. To są nowoczesne ładowarki, najnowocześniejsze na świecie, produkowane zresztą przez rodzimą polską firmę. Te ładowarki będą rozmieszczone w dużych aglomeracjach miejskich i przy głównych trasach transportowych, autostradach, drogach ekspresowych. To spowoduje, że w wyniku przyzwyczajenia kierowców do szybkiego przepływu, szybkiej rotacji samochodów, szybkiego tankowania samochodów konwencjonalnych, później elektrycznych skokowo zwiększy się ilość pojazdów elektrycznych na polskich drogach. Myślę, szanowni państwo, że przed rokiem 2030 - w takiej perspektywie według ekspertów z wielu organizacji branżowych, think tanków - na polskich drogach będzie jeździło milion samochodów elektrycznych. Dodatkowo skierowaliśmy ponad 1 mld zł na rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, 4 tys. km linii sieci dystrybucyjnych, które mają zaopatrzyć w dostawy energii 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych, co z kolei spowoduje możliwość bezpiecznego ładowania pojazdów elektrycznych.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Adam Ołdakowski. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

W ramach programu w całej Polsce powstać ma 100 obwodnic o łącznej długości 820 km. Na realizację programu przeznaczono 28 mld zł. Według założeń budowa obwodnic służyć ma poprawie bezpieczeństwa na drogach, poprawie przepustowości sieci drogowej oraz wyprowadzeniu ruchu z zatłoczonych miast. Realizacja inwestycji ma pozytywnie wpłynąć na środowisko, m.in. przyczynić się do poprawy jakości powietrza czy obniżenia poziomu hałasu. Dzięki realizacji programu powstać mają nowe miejsca pracy. Mają być one również impulsem do rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe. W związku z tym, że minął już rok od przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia ˝Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030˝, chciałbym zadać panu ministrowi pytanie o realizację programu. W szczególności chciałbym dowiedzieć się, jaki jest postęp prac w województwie warmińsko-mazurskim. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie zainteresowani tematem inwestycji drogowych, szczególnie programem budowy 100 obwodnic! Ministerstwo Infrastruktury opracowało program budowy 100 obwodnic. Program ten jest na lata 2020-2030 i, jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcony realizacji obwodnic w ciągach dróg krajowych. Już na wstępie trzeba przyznać, że to pierwszy tak gruntowny i kompleksowy program budowy obwodnic zaproponowany przez polski rząd, a konkretnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych. Szacujemy, że łączna długość wyniesie ok. 820 km. Trzeba podkreślić, że budowane przez nas trasy będą o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t na oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym np. oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji wszystkich 100 obwodnic został oszacowany na 28 mld zł. Mamy na to zabezpieczone środki finansowe w ramach Krajowego Funduszu Drogowego. W chwili obecnej w realizacji znajduje się już 15 inwestycji, z czego obwodnice Wąchocka, Smolajn i Brzezia są w fazie budowy.

85 obwodnic znajduje się na etapie przygotowania, uzyskiwane są niezbędne decyzje administracyjne, w tym przede wszystkim decyzje środowiskowe. Realizacja obwodnic w ciągu dróg krajowych jest bardzo ważna i kluczowa ze względu na likwidację wąskich gardeł na sieci drogowej oraz poprawę warunków podróżowania, jak również eliminację negatywnego wpływu hałasu i spalin na mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu z centrów miejscowości. Trzeba też zaznaczyć, że jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chcemy to osiągnąć poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z zatłoczonych miejscowości. Przyświeca nam zasada: im mniej miejsc styku pojazdów, szczególnie tych ciężkich, z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, pieszymi czy rowerzystami, tym bezpieczniej. Dlatego budowane obwodnice pozytywnie wpłyną na tę sferę naszego życia. Przechodzę już do realizacji programu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na terenie tego województwa planowana jest realizacja pięciu obwodnic. Obwodnica jedna, ale dwóch miejscowości - części Olsztyna i Dywit. Druga obwodnica - miejscowość Gąski. Czwarta - miasto Szczytno. Piąta - Smolajny; jest to miejscowość w gminie Dobre Miasto.

Tu trzeba zaznaczyć, że województwo warmińsko-mazurskie będzie pierwszym województwem, w którym obwodnica w ramach tego programu zostanie oddana do użytkowania. Jesteśmy już w końcówce prac, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Smolajn. Mam nadzieję, że najbliższy kwartał pokaże, że ta droga, ta obwodnica zostanie oddana do użytkowania i będzie już komunikowała drogę krajową nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie pozostałe znajdują się co najmniej na etapie prac przygotowawczych. Jeżeli chodzi o prace przygotowawcze, to prowadzone są one w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które w przypadku tych umów jest poszerzone o elementy koncepcji programowej. Taki sposób przygotowania inwestycji wydaje się najbardziej efektywny i optymalny. W tym przypadku na pierwszym etapie określane są m.in. przebiegi dróg do obsługi przyległego terenu, ustala się typy oraz podstawowe parametry techniczne obiektów inżynierskich. Dodatkowo na tym etapie prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza, która stanowi podstawę do ustalania zakresu i rodzaju stosowanych urządzeń ochrony środowiska. Tak że inwestycje drogowe, które są w tej chwili realizowane, są prowadzone w sposób nowoczesny. Nie tylko po to, żeby korzystanie z samej drogi było bezpieczne i komfortowe, ale też po to, żeby wszystko to, co jest wokół - i to niezależnie od tego, czy to teren zurbanizowany, zamieszkały czy tereny leśne - było również do tej drogi w odpowiedni sposób dostosowane. Albo odwrotnie: żeby budowana droga była dostosowana i spełniała dużo szerszą (Dzwonek) funkcję niż tylko tę komunikacyjną. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wśród inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu budowy 100 obwodnic znalazła się obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych 58 i 63. W trakcie prac nad projektem mieszkańcom gmin Pisz przedstawiono wstępne warianty przebiegu trasy. Nie spotkały się one z akceptacją lokalnej społeczności, ponieważ zakładają przebieg obwodnicy przez tereny zurbanizowane. W ocenie mieszkańców Pisza warianty te nie pozwalają zrealizować głównego celu budowy obwodnicy, jakim jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. W zaproponowanym kształcie nie rozwiązują problemów komunikacyjnych miasta. W praktyce oznaczają też konieczność ingerencji w strukturę zabudowy miasta, w tym budynki mieszkalne.

Zbliżony wariant pojawił się w październiku ub.r. na mapach przygotowywanych przez projektantów z firmy TRAKT, które trafiły do Urzędu Miejskiego w Piszu. Niestety wariant ten wycofano jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji społecznych. Proszę bardzo.

Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o obwodnicę Pisza w ciągu dróg krajowych 58 i 63, to tak jak pan poseł wspomniał, aktualnie realizowane są prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej i elementami koncepcji programowej. Ja znam ten temat, ponieważ spotykałem się z panem posłem Jerzym Małeckim, ale też z innymi przedstawicielami, którzy są zainteresowani budową obwodnicy Pisza. Podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie. My naprawdę nie budujemy dróg wbrew społeczeństwu, tylko dla społeczeństwa. Zawsze staramy się interes społeczeństwa stawiać na pierwszym miejscu. Oczywiście w ramach tego opracowania musimy też analizować elementy środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. One wszystkie tworzą pewną całość, która później decyduje o tym, jaki wariant czy to obwodnicy, czy to danej drogi ekspresowej jest wybierany do decyzji środowiskowej. Jeżeli chodzi o obwodnicę Pisza, to postaramy się dochować należytej staranności, aby wybrać wariant, który przede wszystkim będzie wariantem realizowalnym. Czasami jest tak, że oczekiwania społeczne są słuszne, natomiast jeżeli chodzi o ich realizację, to są po prostu niemożliwe, bo występują przeszkody, np. środowiskowe albo techniczne, albo sam koszt jest na tyle wysoki, że przewyższa zakładane kwoty inwestycji. Natomiast zawsze do takiego tematu podchodzimy bardzo poważnie, starając się słuchać głosu społeczeństwa i w ramach konsultacji społecznych dokonywać jak najlepszych wyborów i jak najlepszych ocen. Tak że mam nadzieję, że jeżeli chodzi o obwodnicę Pisza, z tym tematem sobie poradzimy. Zdanie ostatnie związane jest z sytuacją inflacyjną, z wojną, która jest za naszą wschodnią granicą, przez co mamy widoczne zwyżki materiałów budowlanych. Działania Putina i tutaj są niestety bardzo widoczne i odbijają się na nas negatywnie. Natomiast dzięki decyzji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego dokonamy waloryzacji kontraktów już zawartych, tak aby wszystkie inwestycje, które są w realizacji, które są przygotowywane, nie zostały zatracone, nie zostały wstrzymane, nie zostały zatrzymane. Tak że mam nadzieję, że jeżeli chodzi o program budowy 100 obwodnic, wszystkie inwestycje będą szły zgodnie z naszym planem i zgodnie z naszymi założeniami z roku 2021.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 2377. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, - o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2358 i 2359.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 Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2360, 2367 i 2356. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Mamy wnioski formalne, ale przedtem, proszę państwa.

Wysoka Izbo! Wnoszę o przerwanie i odroczenie posiedzenia do czasu wyjaśnienia, czy pan minister Waldemar Kraska jest kłamcą lustracyjnym czy też być może zaledwie nie został zweryfikowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Korespondencja skierowana do jednego z historyków niezależnych wskazuje, że oświadczenia Waldemara Kraski w ogóle nie poddawano weryfikacji. Takie nasuwają się wnioski. Pani marszałek wie o tym z urzędu od poprzedniego posiedzenia Sejmu. Zachodzi zatem pytanie, czy złożyła wymagane prawem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Proszę bardzo, pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska.

Pani Marszałek! Panie Premierze!

Po pierwsze, nie mamy zabezpieczonego węgla. Rząd proponuję ułomną ustawę, która jest niewykonalna, a nad którą będziemy dzisiaj głosować. Po drugie, nie mamy zabezpieczonych dostaw gazu na najbliższą zimę. Rząd nie mówi prawdy Polakom. Chcielibyśmy, żeby rząd przedstawił jednolitą i pełną koncepcję zabezpieczenia systemu energetycznego dla Polaków.

Bardzo proszę, pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska.

Nie wiecie dziś, ilu macie ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy. Co więcej, doszliście już do takiej obłudy, że nagradzacie stanowiskami ministrów bez teki ludzi, którzy powinni dawno wylecieć z polityki.

Co więcej, Polacy klepią biedę, a wy rozdmuchaliście wydatki KPRM-u o kilkaset procent.

Dziękuję, panie pośle. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie. Otóż odpowiedzią i receptą na te problemy jest przede wszystkim szereg rozwiązań, które wprowadziliśmy.

Czy tego nie widzicie?

Podwyższaliście podatki, podwyższaliście VAT. Nie zrobiliście nic dla tych ludzi. My wprowadzamy wakacje kredytowe, 4 miesiące w tym roku, 4 miesiące w przyszłym. Państwo wtedy zdezerterowało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani poseł Katarzyna Kotula. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę, żeby dać czas klubom i kołom na przemyślenie tego. jak zagłosują dzisiaj w sprawie obywatelskiego projektu ˝Legalna aborcja. Bez kompromisów˝ Chcemy dać czas Prawu i Sprawiedliwości na wycofanie tego haniebnego wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się ponad 200 tys. obywateli i obywatelek. To jedyny projekt, który przywraca Polkom godność i poczucie bezpieczeństwa. Drogie Polki!

Proszę bardzo, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Wysoka Izbo! Z wczorajszej dyskusji o ustawie węglowej ponad wszelką wątpliwość wynika, że zimą tego roku w Polsce zabraknie węgla. Czy macie tego świadomość? Co chcecie w tym zakresie zrobić? Czy zabraknie również gazu? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałam przywitać siedzącą na galerii młodzież z Zespołu Szkół nr 5, z VII Liceum Ogólnokształcącego z Płocka i wolontariuszy, którzy pomagają walczącej Ukrainie i Ukraińcom. Witamy was.

Proszę bardzo, głosujemy nad wnioskiem o przerwę. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2375. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 2375? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2313-A. Proszę pana posła Mariusza Trepkę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie komisji dotyczące rządowego projektu ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, druki nr 2308 i 2313.

Jednocześnie w dodatkowym sprawozdaniu komisje przedstawiają poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Kto jest za przyjęciem 4. poprawki?

Sejm poprawkę przyjął. Kto jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2313, wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2357-A. Proszę pana posła Andrzeja Kryja o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie!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 Sejm w dniu 22 czerwca 2022 r. skierował ponownie projekt ustawy zawarty w drukach nr 2351 i 2357 do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po wnikliwym ich rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r. wnosi, aby Wysoki Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy, odrzucił poprawki 1., 2., 3., 4. i 5., przyjął poprawki 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., z tym że nad poprawkami 6., 7., 8., 11. i 12. należy głosować łącznie, oraz przyjął przedłożony projektu ustawy w całości. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2357. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w całości. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości? Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 3. poprawki? Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 4. poprawki? Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 5. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem 10. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2357, wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2363-A. Proszę pana posła Grzegorza Matusiaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Podczas drugiego czytania zgłoszono poprawkę. Komisja przedstawia również poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2363? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz Prawo ochrony środowiska. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 2362-A. Proszę panią poseł Ewę Szymańską o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz Prawo ochrony środowiska z druku nr 2352. Sejm na bieżącym posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r., zgodnie za art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2362 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2022 r., wnosi, aby Wysoki Sejm raczył odrzucić wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz wszystkie trzy poprawki, z tym że poprawki 2. i 3. należy rozpatrywać łącznie. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 2362. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości? Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2362? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. W dyskusji złożono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji po doręczeniu zestawienia poprawek. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem poddam ten wniosek pod głosowanie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji po doręczeniu zestawienia poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek przyjął. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone do druku nr 2361. Przystępujemy do trzeciego czytania. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 3. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 5,. 6. i 8. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawki odrzucił. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem 5. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 6. poprawki? Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem 8. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 10. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 11. poprawki? Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto jest za przyjęciem 13. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 14. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za przyjęciem 15. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2361, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? U kogo nie działa?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych. W dyskusji zgłoszono wnioski: o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu oraz o przystąpienie niezwłocznie do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 2298? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2275 i 2358) Proszę pana posła Leszka Galembę o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu komisji rolnictwa przedstawić sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2275.

Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 - za, przeciw - 438, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 3. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 4. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 5. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem 6. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Kto jest za odrzuceniem 7. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? U kogo nie działa?

Sejm odrzucił poprawkę.

Kto jest za odrzuceniem 11. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2342 i 2359) Proszę pana posła Jerzego Małeckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, druk nr 2342. Marszałek Sejmu zgodnie z regulaminem Sejmu skierowała w dniu 10 czerwca 2022 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wnosi, żeby poprawki 2. i 5. przyjąć, pozostałe poprawki odrzucić, a nad poprawkami 3., 4., 6., 8. i 10. głosować łącznie. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 440 posłów. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Senat proponuje zmiany o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 5. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 7. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie był za, przeciw - 441, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 11. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2343 i 2367) Proszę pana posła Tomasza Latosa o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2343 i 2367. Senat przedstawił 22 poprawki. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Kto jest za odrzuceniem 6. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 8. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 11. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę.

Sejm odrzucił poprawkę.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 Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek!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 Marszałek Sejmu skierowała w dniu 10 czerwca uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia.

Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan minister Paweł Szefernaker. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Ja chciałbym bardzo podziękować Wysokiej Izbie za to, że przyjęliśmy tutaj 2 tygodnie temu ustawę pomocową ponad politycznymi podziałami. Ustawa trafiła do Senatu. Ustawa ma charakter systemowy, te przepisy wychodzą bardzo często poza jej zakres przedmiotowy. W tej ustawie są również przepisy związane z zakupem interwencyjnym węgla właśnie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Te przepisy, które są w tej ustawie, mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa polskim obywatelom w zakresie ceny ciepła. To są przepisy, które mają pozwolić na to, aby jak najszybciej można było zakupić węgiel poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i zmienić sytuację na rynku węgla w Polsce, uruchomić zakupy interwencyjne. Niestety Senat przyjął poprawkę, która usuwa te przepisy. To jest hipokryzja, dywersja i sabotaż, proszę państwa. Rząd przyjął przepisy, które pozwalają na zakup tego węgla, i Senat te przepisy usuwa. Nienawiść do PiS-u przysłania wam zdrowy rozsądek.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 3. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2341 i 2360) Proszę panią poseł Annę Milczanowską o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2341.

Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. W uchwale Senat proponuje odrzucić ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Głosujemy.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Józefa Wojciechowskiego, reprezentowanego przez adwokat Katarzynę Witkowską z dnia 15 lipca 2020 r., poprawionego w dniu 24 sierpnia 2020 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka. Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka. Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Józefa Wojciechowskiego, reprezentowanego przez adwokat Katarzynę Witkowską z dnia 15 lipca 2020 r., poprawionego w dniu 24 sierpnia 2020 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka za czyn określony w tym wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

2 było za, przeciw - 431, 5 się wstrzymało. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Józefa Wojciechowskiego, reprezentowanego przez adwokat Katarzynę Witkowską z dnia 15 lipca 2020 r., poprawionym w dniu 24 sierpnia 2020 r. Przypominam, że uprawnione podmioty złożyły wnioski o uzupełnienie porządku dziennego: - Koło Parlamentarne Polska 2050 o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu systemu zarządzania kryzysowego oraz działań Rady Ministrów na rzecz jego wzmocnienia w związku z awarią w dniu 19.02.2022 r. numeru alarmowego 112 i nieprawidłowym działaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w całym kraju; - Koalicyjny Klub Poselski Lewicy o punkty: - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie konieczności wprowadzenia dotkliwych sankcji wobec władz Federacji Rosyjskiej oraz powiązanych z nią oligarchów, Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania Polski do udzielenia obywatelom Ukrainy ewentualnej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, zamieszkania oraz prac na terytorium RP, w przypadku eskalacji konfliktu z Federacją Rosyjską i napływu do Polski uchodźców z Ukrainy. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Głosujemy nad wnioskiem w sprawie uzupełnienia porządku dziennego o punkt dotyczący informacji na temat stanu systemu zarządzania kryzysowego. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy nad wnioskiem w sprawie uzupełnienia porządku dziennego o punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie konieczności wprowadzenia sankcji wobec władz Federacji Rosyjskiej oraz powiązanych z nią oligarchów. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy nad wnioskiem w sprawie uzupełnienia porządku dziennego o punkt dotyczący informacji w sprawie przygotowania Polski do udzielenia obywatelom Ukrainy pomocy w przypadku eskalacji konfliktu z Federacją Rosyjską i napływu do Polski uchodźców z Ukrainy. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Prezydium Sejmu, na podstawie art. 20 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 2377? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm podjął uchwałę Na tym zakończyliśmy głosowania.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Informacja bieżąca. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie analizy funkcjonowania Funduszu Medycznego, o przedstawienie której wnosił Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciele Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenia punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut.

Grupa zwiedza Sejm na zaproszenie posła Jana Dudy. Serdecznie wszystkich państwa witamy. Uprzejmie proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Dariusza Klimczaka. Dziękuję, pani marszałek.

Szanowni Państwo! Autorem idei powstania specjalnego funduszu, który by pomagał chorym dzieciom, szczególnie na choroby rzadkie, choroby, których leczenie nie jest refundowane, choroby onkologiczne, był ówczesny kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten pomysł w kampanii wyborczej podchwycił pan prezydent Andrzej Duda i go przedstawił Sejmowi. Ale dzisiaj ten fundusz jest. Zamiast realnej pomocy dzieciom chorym onkologicznie i na choroby rzadkie mamy niewykorzystane środki finansowe naprawdę ogromnej wielkości.

W roku 2021 w ramach Funduszu Medycznego przeznaczono na to tylko 21% całego budżetu. Według najnowszego raportu Najwyżej Izby Kontroli dysponent Funduszu Medycznego nie zrealizował w ubiegłym roku czterech z ośmiu zadań tego funduszu, co świadczy o słabości instytucjonalnej Ministerstwa Zdrowia. W 2021 r. zrealizowano przede wszystkim zadania z lat ubiegłych, a ich faktycznym wykonawcą był NFZ. Wszystkie nowe zadania wprowadzone ustawą o Funduszu Medycznym, które wymagały pracy urzędników, były w całym ubiegłym roku przygotowywane, uzgadniane.

NIK, Najwyższa Izba Kontroli zaleca niezwłoczne rozpoczęcie realizacji wszystkich zadań funduszu, a tym samym zasilenie systemu ochrony zdrowia środkami zgromadzonymi na rachunku tego funduszu. Oczywiście ministerstwo deklaruje, że niewykorzystane środki przejdą na kolejny rok. Mija połowa roku, a my nie wiemy nic. Nie wiemy, na co te pieniądze, w jakich proporcjach, a przede wszystkim kiedy zostaną przekazane. Szanowni Państwo! Nasz apel jest apelem o to, aby znowelizować tę ustawę i w przejrzysty sposób zaplanować proces legislacyjny. Dzisiaj jest Dzień Ojca.

Zebrała 5 mln zł, ale musi nazbierać drugie 5 mln zł. Leżą pieniądze, niewykorzystane, a to dziecko leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jak to się dzieje, że Ministerstwo Zdrowia, że ten rząd nie potrafią tych pieniędzy zadysponować? Dlaczego tak się dzieje, że wciąż trwają negocjacje nad refundacją najdroższego leku świata?

Czy to państwa nie boli? Mnie to bardzo boli. Dlatego dołączam się do wielu organizacji pacjenckich, występujących do ministerstwa z prośbą o dokonanie pilnych zmian w Funduszu Medycznym i efektywne wydawanie tych środków. Pod koniec roku 2021 Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Ta nowelizacja miała poszerzyć zasięg finansowania o szczepienia przeciwko HPV, diagnostykę genetyczną, molekularną w onkologii, ale niestety do dzisiaj ten projekt nie ujrzał światła dziennego. Ministerstwo, kiedy pytamy w interpelacjach, bardzo nieprecyzyjnie odpowiada na nasze pytania. W naszym przekonaniu należy niezwłocznie podjąć pracę nad nowelizacją ustawy o Funduszu Medycznym, tak aby fundusz spełniał (Dzwonek) swoje zadania, niósł faktyczną pomoc polskim pacjentom i poprawił dostęp do diagnostyki i leczenia najtrudniejszych chorób. Pragniemy, żeby był uwzględniony głos pacjentów. Rodzice, z którymi rozmawialiśmy, nawet dysponują swoim czasem. Bardzo prosimy o uwzględnienie tej kwestii w imieniu naszego klubu, ale przede wszystkim w imieniu tych małych, chorych pacjentów, którzy czekają na finansowanie ich leczenia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana ministra Marcina Martyniaka. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym powiedzieć, że Fundusz Medyczny to jest koncepcja wieloletnia i to było od samego początku podkreślane.

Natomiast na pewno nie będzie to tego typu kwota, bo oznaczałoby to wydatkowanie całości środków przeznaczonych na ten rok. A więc czekamy na finalną decyzję w oparciu o analizy, które w chwili obecnej są tworzone w Ministerstwie Zdrowia.

To oznacza, że popyt i pewnego rodzaju potrzeba są tutaj jak najbardziej widoczne. Ogłoszenie listy rankingowej będzie miało miejsce w najbliższym miesiącu. Mam tu na myśli lipiec. Jeśli chodzi o plany w zakresie subfunduszu infrastruktury strategicznej, to w III kwartale jeszcze tego roku będzie ogłoszony konkurs w zakresie wsparcia szpitali onkologicznych.

Możliwe, że jeszcze w tym roku, pod koniec tego roku pojawi się jeszcze jeden konkurs subfunduszu infrastruktury strategicznej. I chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną ważną rzecz. To, że środki nie zostały wydatkowane w tym roku czy w roku poprzednim, nie oznacza, że ta alokacja zostanie przetrawiona, przejedzona czy też zostawiona w bliżej nieokreślonym celu. To są środki wieloletnie, infrastrukturalne projekty wymagają wieloletnich ram czasowych.

Oczekuje na swoją kolej w Komitecie Stałym Rady Ministrów i procedowanie w ramach tego organu. Wejście w życie tej uchwały warunkuje ogłoszenie kolejnych konkursów.

Jeśli chodzi o plany na najbliższe 2 lata w zakresie subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, to jest to właśnie wydatkowanie tych niemal 350 mln zł oraz 700 mln na wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych. Kolejny, trzeci subfundusz, subfundusz rozwoju profilaktyki.

Między innymi z tego powodu - przecież Fundusz Medyczny, tak jak słusznie pan poseł zauważył, jest projektem, którego inicjatorem jest pan prezydent - i z potrzeby zanalizowania rozwoju obszaru profilaktyki został uruchomiony chyba niecałe 2 tygodnie temu program ˝Zdrowe życie˝ pod patronatem pana prezydenta we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, PZU oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych.

I kwartał, 3 miesiące - 275 mln. Łatwo policzyć, że będzie to ponad miliard złotych w tym roku.

Z czego to wynikało, szanowni państwo? Wynikało to z tego, że systemy ochrony zdrowia w innych państwach również się zlockdownowały, po prostu.

A więc możemy oczekiwać zdwukrotnienia albo nawet zwielokrotnienia środków, które będą przeznaczane na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju. Opracowano listę technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. To jest konieczność przejrzenia wszystkich list lekowych, to jest praca wielomiesięczna, która jest ukierunkowana na dobro pacjenta, dlatego że te leki muszą być ukierunkowane i jak najlepiej dobrane. To nie może być praca wykonana w sposób bardzo pobieżny i niedokładny.

Wnioski zostały złożone również dla pięciu leków. Finalnie objęto refundacją dwa z nich. Już mówię.

Ponadto opracowano drugą listę w zakresie TLI, oczywiście zgodnie z terminem ustawowym, gdzie znalazło się już 11 technologii lekowych. Minister poinformował już podmioty odpowiedzialne o tym, które technologie lekowe znajdują się na tej liście, i o możliwości złożenia wniosku.

Dla porównania pod koniec maja mamy bardzo podobny wynik.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość w ramach tego czwartego subfunduszu, jesteśmy na dobrej drodze - ten wątek też był poruszony przez pana posła - w rozmowach z kancelarią pana prezydenta i (Dzwonek) rozmowy są na etapie finalizacji w zakresie wprowadzenia nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Puentując, chciałbym powiedzieć, że ten fundusz jest czymś, czego dotychczas w Polsce nie było. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że duża, ogromna część alokacji dotyczy kwestii infrastrukturalnych, a jak powiedziałem na wstępie, te środki nie mogą być wydatkowane w ciągu roku, bo nie wyobrażam sobie, żeby inwestycje, nawet te o wartości ponad 300 mln zł, były realizowane w ciągu jednego roku. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze zapisać się do głosu? W takim razie zamykam listę mówców.

Otwieram dyskusję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak, to prawda, że fundusz działa prawie 2 lata. Tak, to prawda, że mamy wiele zastrzeżeń do działalności tego funduszu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykorzystanie środków. Ale są też racje, i to wcale nie takie małe, po stronie pana ministra. To jest fundusz o rachunku ciągnionym, a nie budżetowym, czyli nie rok do roku, ale w perspektywie 10-letniej, i musimy o tym pamiętać. Większość zadań tych subfunduszy, a jest ich przecież cztery, nie ma charakteru doraźnego, bo ten fundusz nie ma w ogóle, panie pośle, charakteru doraźnego.

To po pierwsze. Ona wynika z Prawa farmaceutycznego, które służy do tego, żeby ustalić cenę na rynku polskim, i to są długie negocjacje. Cieszę się, że ten fundusz już ruszy, i mam nadzieję, że to, co pan minister nam przedstawił, wreszcie zacznie skutkować - w sprawach infrastruktury, w sprawach modernizacji podmiotów leczniczych, w rozwoju profilaktyki.

Chodzi o kadry medyczne.

Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Najwyższy czas, żeby Polska przestała być krajem zrzutka.pl. Najwyższy czas, żeby przywrócić godność tym rodzicom, którzy muszą błagać, żebrać, zbierać nakrętki, żeby uratować swoje dzieci. Fundusz Medyczny powstał po to, żeby pomagać właśnie chorym dzieciom, żeby pomagać ludziom chorym na choroby rzadkie, żeby pomagać dzieciom chorym na choroby onkologiczne, żeby finansować oryginalne, rzadkie terapie albo operacje za granicą. Po to powstał fundusz. Wy z tego funduszu zrobiliście pewną zabawkę, po to żeby pokazywać, że więcej pieniędzy wydajecie na służbę zdrowia. W momencie, w którym przekazujecie te pieniądze, rok po roku, rolujecie je. Byłyśmy wspólnie z panią Moniką Wielichowską na kontroli w Ministerstwie Finansów. Dowiedziałyśmy się, że w roku 2022 również pieniądze nie zostaną wydane, a na rok kolejny zostanie w sumie przeznaczonych już 5,3 mld niewykorzystanych pieniędzy. które zostaną zrolowane na kolejny rok. W ten sposób, jeżeli będziemy tak sumować, to za kilka lat okaże się, że mnóstwo pieniędzy jest przeznaczonych na zdrowie, bo nie są wydawane na to, na co powinny zostać wydane. Nie może być tak, że rodzice, którzy mają dziecko chore na SMA, żebrzą. Nie może być tak, że mamy pieniądze, tylko nie sięga się po nie, ponieważ ktoś chce sobie budować statystyki dotyczące tego, ile w przyszłym roku wyda na ochronę zdrowia. To jest wielkie oszustwo. Najwyższy czas skorzystać z pieniędzy, które są (Dzwonek), na to, na co są przeznaczone.

Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zacznę od tego, że kilkadziesiąt milionów złotych, które mogłyby być przekazywane na terapie genowe dla dzieci z SMA rokrocznie, nie stanowiłoby dużego uszczerbku dla budżetu państwa. Pani Marszałek!

Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Panie Ministrze!

A przecież teoretycznie to z inicjatywy pana prezydenta powstała ta ustawa. Wiem, ile państwo pomogli w napisaniu tej ustawy i przeprowadzeniu jej przez parlament. Ale czy to nie byłoby honorowe, żeby pan prezydent lub jego przedstawiciel dzisiaj tutaj był? I czy państwo pytali, czy ktoś zechce tutaj przyjść? Pan nie odpowiedział w pierwszej rundzie - mam nadzieję, że w drugiej rundzie pan odpowie - na zasadnicze pytanie: Jaka jest konkretna liczba pacjentów, którzy do tej pory skorzystali z Funduszu Medycznego, ile terapii lekowych do tej pory zostało sfinansowanych w ramach Funduszu Medycznego i ilu pacjentów korzysta aktualnie z nowych opcji terapeutycznych? Jeżeli pan dzisiaj nie jest w stanie jej przedstawić, bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja.

Szczęść Boże! Wracam do pytania, które stawiałem już z tej mównicy i nie uzyskałem odpowiedzi. Pytania o biografię ministra Waldemara Kraski. Kto w tym resorcie zarządza zdrowiem, życiem, również majętnością Polaków, kto podejmuje decyzje ważące na życiu i przyszłości Polaków, nie powinien być postacią bez biografii. A taką postacią jest Waldemar Kraska.

Każdy z nas, kto pamięta, kto przeżył już jako dorastający czy dorosły człowiek lata 80., miał coś do opowiedzenia światu o tym, po której stronie wtedy był. Waldemar Kraska nie odpowiada na pytania. Zatem ponawiam je i proszę o odpowiedź na piśmie: Jaka jest ścieżka kariery edukacyjnej, zawodowej, naukowej Waldemara Kraski przed rokiem 1989? Jaką służbę odbywał? Jakie szkolenia przechodził? Jaki być może mundur mu przysługuje?

Panie pośle, proszę już usiąść i nie przeszkadzać. Proszę nie utrudniać pracy. Panie pośle, proszę zaczynać. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Fundusz Medyczny nie działa.

Pytanie: Czy pieniędzy w ochronie zdrowia jest już za dużo? Otóż nie. Portale są pełne zbiórek na terapie, za którymi stoją dramatyczne historie o zdrowiu i nieszczęściu także młodych Polek i Polaków. I to jest szczególnie bulwersujące. Pan prezydent i rząd PiS wmawiali Polakom, że życie ludzkie jest dla nich najważniejszą z wartości. Okazało się, że mijali się z prawdą, ponieważ kiedy trzeba było ratować to życie i zdrowie, przejść od słów do czynów, to posłowie i ministrowie z PiS odwrócili wzrok i trzymają 3,5 mld zł na kontach.

Panie ministrze, dziś pan reprezentuje całą tę władzę i wmawia nam, że wszystko jest dobrze. Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego tysiące ludzi błaga na portalach o pomoc? Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Nie ulega wątpliwości, że służba zdrowia po okresach rządów Platformy Obywatelskiej, PSL, SLD była na takim poziomie, że należało natychmiast podjąć działania, żeby ją ratować. Przypomnę państwu, że w 2015 r. wydawaliście na ochronę zdrowia 74 mld zł. Teraz jest ponad 126 mld zł.

Szanowni państwo, jeżeli chcecie rozmawiać merytorycznie o Funduszu Medycznym, to przyjmijcie do wiadomości, że jest to program 10-letni.

W ubiegłym roku np. na leczenie dzieci, o których pan poseł mówił, wydano ponad 527 mln zł, na starcie tego programu. Kolejne działania są daleko zaawansowane.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Powstanie Funduszu Medycznego miało zupełnie inne podłoże niż troska władzy o bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków. Miał być lekiem na fale krytyki, był odpowiedzią na wpadkę prezydenta z ostrym cieniem mgły i przekazaniem 2 mld zł na telewizję Kurskiego zamiast na walkę z rakiem. No bardzo dobrze brzmiał w kampanii, bardzo dobrze brzmiał PR-owsko, ale dzisiaj rodzice nadal muszą zbierać pieniądze na leczenie dzieci, choć PiS obiecał, że będzie inaczej. Nie dość, że nie ma dodatkowych pieniędzy w budżecie Ministerstwa Zdrowia, to jeszcze te, które zostały przesunięte do funduszu, są po prostu rolowane. Fakty są takie, że w 2021 r. z Funduszu Medycznego wydano zaledwie 21% z całego 4-miliardowego budżetu. Ministerstwo Zdrowia oczywiście zapewnia, że niewykorzystane środki mają przejść na kolejny rok, a to oznacza, uwaga, że w tym roku do przeznaczenia będzie ponad 7 Fakty są takie, że dzisiaj niewielu pacjentów skorzystało z możliwości leczenia nowoczesnymi terapiami z funduszu. Jest to związane zarówno z niepełnym wydatkowaniem ulokowanych do tego funduszy, jak i z długim procesem decyzyjnym, który niestety opóźnia dostęp pacjentów do leczenia. Mam pytania do pana ministra: Ilu pacjentów skorzystało dziś z refundacji najbardziej nowoczesnych terapii w ramach funduszu? Jaka jest planowana alokacja środków, które zostały z poprzednich lat? Dlaczego droga ubiegania się o taką refundację (Dzwonek) jest utrudniona i generuje zbędne opóźnienia w dostępie pacjentów do leczenia?

Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! We wrześniu 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o Funduszu Medycznym, w której zagwarantowano rządowi olbrzymie pieniądze na jak najwcześniejsze wykrywanie i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, chorób rzadkich. I co ministerstwo zrobiło za tak gigantyczne pieniądze? Gdy rodzice, lekarze, parlamentarzyści prosili i błagali ministra zdrowia i rząd o dofinansowanie czyjejś drogiej terapii i ratowanie życia, zawsze słyszeli jak mantrę, że rząd nie ma pieniędzy, bo gdyby je miał, toby je dawał. Teraz rząd ma te pieniądze, ale nie daje ich ciężko chorym pacjentom, bo dla niektórych polityków pacjent to koszt i problem w statystyce, a nie potrzebujący pomocy człowiek. Apeluję do pana ministra zdrowia, żeby wytłumaczył pacjentom i rodzinom tych pacjentów, także tym rodzinom, które niestety nie doczekały terapii swoich dzieci, dlaczego pieniądze przekazane na ich leczenie, przekazane panu ministrowi, nie zostały wykorzystane i zostały zmarnowane. To jest skandal.

10 lat - niektóre dzieci tego nie doczekają. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Gdy podejmowaliśmy decyzję o stworzeniu Funduszu Medycznego, chcieliśmy przede wszystkim pomagać ludziom, pomagać tym, którzy niestety nadal muszą zbierać te środki w różnego rodzaju zbiórkach, wiedząc, że czas jest dla nich najważniejszy. Proszę o podanie informacji na temat negocjacji z firmą mającą ten lek. Ile one trwały? Czy w procesie negocjacji środowiska pacjentów miały jakąkolwiek możliwość wypowiedzenia się? Dlaczego zostały one przerwane? Kiedy możemy liczyć, że zostaną przywrócone? Czy w innych krajach można to robić szybciej, skuteczniej? W Polsce jak zwykle mamy problem. To jest 3,5 mld wstydu, bo te pieniądze powinny po prostu pracować. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jak w ogóle śmiecie coś takiego z tej trybuny mówić? Ten fundusz miał poprawić los pacjentów z chorobami rzadkimi. Dlaczego w 2021 r. wydano zaledwie 21% budżetu? Dlaczego wydawano środki z zaledwie jednego z czterech subfunduszy? Jakie były osobowe koszty zarządzania tym funduszem w tym czasie? Ci ludzie walczą o zdrowie swoich dzieci. Przyzwoitości troszkę. Właśnie przyzwoitości. Naprawdę nie grajmy nieszczęściem dzieci. Jasne. Pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na początek chciałam podziękować klubowi, który zgłosił tę informację bieżącą, bo to jest bardzo ważny temat. Nawet zaczęło się merytorycznie w odróżnieniu od poprzednich informacji, które były z różnych klubów. Temat jest bardzo ważny.

Tak, ograniczyć, bo pewnie w żadnym kraju nie udałoby się tego całkowicie znieść, bo mówimy o bardzo wielkich pieniądzach.

Pewnie to, co najważniejsze, to kadry.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Rozpoczął pan przede wszystkim od subfunduszy, nie przede wszystkim, ale po prostu, po kolei idąc, od subfunduszu na modernizację szpitali.

Tutaj akurat nie trzeba było żadnych wielkich przygotowań, bo tu się szpitale nie przygotowywały do tego, tylko państwo się przygotowywaliście do ogłoszenia konkursu. Jest to konkurs, który powstał dla szpitali nie tylko pediatrycznych, ale także zakwalifikowanych do poziomu czwartego, piątego i szóstego. W takim układzie mam pytanie do pana ministra: Kiedy pozostałe szpitale z poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego też będą mogły skorzystać z tego Funduszu Medycznego, ponieważ mówiło się, że to jest na modernizację wszystkich szpitali?

Powtarza się niestety sytuacja, że beneficjenci są prawie zawsze ci sami i są to beneficjenci, którzy nie są szpitalami, tak jak powiedziałam, z pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam przed oczami taką scenę, jak umierał Jan Paweł II i nie mógł oddychać.

Mamy czas i to jest proste, ale nie jest proste dla tych, co nie mają czasu. To jest po prostu skandal, żeby mając miliardy złotych, nie pomóc ludziom, rodzinom, którzy potrzebują pomocy. Opowiadanie tutaj, że to jest jakiś atak, że to jest jakieś wyobrażenie, na które nie ma miejsca, bo to jest polityka. Jaka polityka? Nie macie kompetencji bądź nie macie sposobu na to, żeby te pieniądze wydać rozsądnie. Pan minister mówi, że przez kilka miesięcy muszą przejrzeć ileś tam rzeczy. A co innego robicie? To jest skandal. Opowiadanie, że to wszystko można przesunąć, jest niedorzeczne. Rozumiem, że nie ma pieniędzy, że możemy szukać pieniędzy, ale jak leżą miliardy, a nie możemy pomóc ludziom, nie możemy nauczyć lekarzy tego, co robią (Dzwonek) za granicą, nie możemy sprzętu sprowadzić odpowiedniego, to na to nie mam już słów. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, Koalicja Polska. Nie widzę. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050. Nie ma. Bardzo proszę, panie pośle.

Szanowni Państwo! Mówimy o bardzo newralgicznym i ważnym Funduszu Medycznym. Jestem akurat osobą, która od wielu lat jest prezesem organizacji pozarządowej, która setki tysięcy złotych zebrała w różnego rodzaju zbiórkach i przekazała na leczenie dzieci. Nie pamiętam dyskusji w ogóle na ten temat. A kiedy my, pan minister, pan prezydent wychodzimy z pomysłem, że będą dodatkowe pieniądze, fundusz powstaje, powstaje w październiku roku 2020, jest pandemia, a tak potężny fundusz trzeba usprzętowić w statuty, w regulaminy.

Wtedy nie ma czasu przeglądać właśnie tych wniosków, bo wy zawracacie głowę. Wróćmy do meritum. Panie Ministrze!

Dlatego musimy pomagać drugiemu człowiekowi. Pan poseł Marek Hok, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze Nieobecny! Wysoka Izbo!

A mianowicie są to: subfundusz rozwoju profilaktyki - od początku roku 2020 wydatkowano z tego subfunduszu 0 zł, subfundusz modernizacji podmiotów medycznych - od początku wydatkowano 0 zł, subfundusz infrastruktury strategicznej - od początku wydatkowano 0 zł. A tymczasem czekają tysiące, setki, miliony ludzi, Polaków na pomoc medyczną. W subfunduszu profilaktyki były również badania w kierunku onkologicznej profilaktyki.

W roku 2020 zachorowały 3862 pacjentki, zmarły 2137. Gdybyśmy szczepili, co było obiecane w Funduszu Medycznym, dzieci, dziewczęta i chłopców, ten problem by się kończył.

Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Nie ma. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, pani poseł.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Planowaliśmy przeznaczać na to rocznie ok. 600 tys. zł. Czy sądzi pan, że kwestia pandemii w ubiegłym roku, który był praktycznie pierwszym rokiem działania Funduszu Medycznego, była przyczyną tego, że podmioty nie sięgały po te środki?

Czy podjęliście jakieś decyzje, aby konsultanci krajowi zachęcali do korzystania ze środków funduszu? Inwestycje mają zawsze swój bieg, to wiemy.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Stworzyliście fundusz, który teoretycznie ma pomagać, teoretycznie ma dawać możliwość sfinansowania bardzo drogich leków, bardzo drogich terapii.

To bardzo dużo pieniędzy. Jakie kwoty w tym roku zostaną wydatkowane w ramach Funduszu Medycznego? Rodzice zbierający kolejne pieniądze, kolejne złotówki, kolejne miliony. Czy zamierzają państwo zrobić cokolwiek, żeby umożliwić rodzicom, żeby nie musieli zbierać kolejnego miliona złotych na bardzo drogie terapie ratujące życie i zdrowie swoich dzieci, żeby ten podatek po prostu znieść? To jest strasznie nieuczciwe, że po pierwsze, leki nie są refundowane w ramach Funduszu Medycznego, a po drugie, dodatkowo jeszcze dorzuciliście podatek. Zapraszam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Fundusz Medyczny jest oczywiście niesamowicie ważny. Powstał za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jest on drugim pod względem częstości występowania, po raku piersi, nowotworem złośliwym u kobiet na świecie, a w Polsce odnotowuje się ok. 3 tys. zachorowań na raka szyjki macicy rocznie.

Poproszę o przedstawienie szczegółów tej nowelizacji. Drugą kwestią, o którą chcę zapytać, jest to, że najbardziej innowacyjne terapie są finansowane przez Fundusz Medyczny, który gwarantuje skrócenie czasu od momentu zarejestrowania leku w Unii Europejskiej do momentu jego refundacji w Polsce. Proszę o przedstawienie takiej ścieżki refundacji. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rozmawiamy dzisiaj o Funduszu Medycznym, o funduszu widmo. Dzisiaj jest smutny dzień dla pacjentów i dla pracowników ochrony zdrowia.

Niestety rządzący nie myśleli o chorych dzieciach.

Telewizja Kurskiego otrzymała każdego roku po 2 mld zł i wydała te pieniądze. Raport NIK-u potwierdza zarzuty, że w Funduszu Medycznym nie sporządzono w 2021 r. planu rzeczowo-finansowego. Nie przeprowadzono też naboru do subfunduszy modernizacji podmiotów leczniczych, infrastruktury strategicznej i rozwoju profilaktyki. Państwo z PiS-u mówicie dzisiaj, że trzeba rozmawiać. Nie, dzisiaj trzeba ratować ludzi. Drodzy Rodzice!

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po raz pierwszy powstał Fundusz Medyczny.

Wtedy będzie dużo lepiej. Po raz pierwszy powstała strategia onkologiczna. Państwo tego nie zrobiliście.

Taka jest sytuacja i taka jest prawda.

Jak będzie można z tych subkont skorzystać? Zapraszam, pani poseł.

Pani Marszałek!

O ich zdrowie i życie walczą ich rodzice, opiekunowie, społeczności lokalne. To jest poważna choroba. Trzeba wspierać rodziny, ponieważ nie możemy liczyć na Fundusz Medyczny. Fundusz Medyczny był obiecywany pacjentom, był gwarantowany po to, żeby leczyć te dzieci.

Jedną z nich jest właśnie SMA.

Z dnia na dzień pogarsza się ich stan zdrowia. Terapia genowa stanowi dla tych dzieci wybawienie i szansę na normalne życie. Im dziecko szybciej dostanie lek, tym szybciej będzie mogło zostać wyleczone i tym mniejsze spustoszenie poczyni choroba w jego organizmie.

Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość.

Temat jest trudny. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

4 maja w szpitalu powiatowym w Wieluniu na świat przyszedł Jaś Rychlik, który został objęty, tak jak każde rodzące się w Polsce dziecko, badaniami przesiewowymi, na które szansy nie miały noworodki za czasów Platformy Obywatelskiej. Są to obligatoryjne badania, które od kilkudziesięciu miesięcy przeprowadzane są w Polsce. Pragnę zapytać, czy zakres tych badań będzie w najbliższym czasie poszerzony o kolejne schorzenia.

Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Warto przypomnieć, że Najwyższa Izba Kontroli negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Funduszu Medycznego. To jest dla nas bardzo ważna informacja. Druga bardzo ważna informacja dotyczy tego, na jaką kwotę były finansowane świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju. Szanowni państwo, to było tylko 60 988 tys. zł.

Mamy do czynienia z człowiekiem, który był w komunistycznym wywiadzie, który może upozorować swoją śmierć, może zmienić tożsamość i nigdy nie zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Żądam również informacji w tej sprawie.

Wydano wyłącznie 37,4% tego planu. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze, proszę państwa, proszę nie oszukiwać społeczeństwa, że mamy do czynienia z listą leków i listą pacjentów. To nie tak.

Nieprawda. Fakt jest taki, że jest bardzo dużo potrzebujących, ale jest bardzo dużo skomplikowanej procedury. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma istotne znaczenie, ponieważ zgłoszenie produktu, jego wykupienie, jego przeznaczenie do danej choroby to jest skomplikowana procedura. NIK też o tym napisał, że te procedury są bardzo skomplikowane, i nie jest to tak, jak się leczy powszechne choroby. Potrzeby są ogromne. Chciałam spytać, czy pani posłanka korzysta z tego portalu, żeby pomagać pacjentom, bo ja korzystam i wysyłam kwoty, o które proszą.

Dziękuję. Pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście Fundusz Medyczny - na początku tak się wydawało - był wielką nadzieją dla wielu zdesperowanych rodziców, którzy każdego dnia walczą o przyszłość swoich chorych dzieci. Ja też chciałem się zwrócić w imieniu wszystkich rodziców, których dzieci są chore na SMA. Rząd niestety nie podjął i nie podejmuje decyzji dotyczącej refundacji tego leku, a zebranie 9 mln, a w tej chwili blisko 10 mln, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć, to jest niesamowite wyzwanie.

Panie Ministrze!

Rodzice dostali następny cios w plecy, bo muszą zebrać dodatkowe 700 tys. czy 800 tys. zł. Ale możecie w tej chwili załatwić to, aby te najdroższe terapie nie były objęte tą stawką. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Celem utworzenia Funduszu Medycznego było utworzenie dodatkowej możliwości finansowania, dodatkowych źródeł finansowania różnych działań z zakresu ochrony zdrowia: profilaktyki, diagnostyki, leczenia. Środki, którymi dysponuje Fundusz Medyczny, są niemałe. Dotychczas nie były w pełni wykorzystane, ale wiemy, że przechodzą na kolejny okres. Panie ministrze, czy któryś z obszarów finansowania objętych celem działania Funduszu Medycznego będzie szczególnie priorytetowy dla Ministerstwa Zdrowia w najbliższych miesiącach? Dziękuję. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Gdy podczas kampanii wyborczej pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie projektu ustawy o Funduszu Medycznym, pomyślałem: to jest genialne posunięcie. Bo wszyscy obserwowaliśmy, jak w mediach społecznościowych, ale także tych tradycyjnych pojawiały się ogłoszenia, rodziny apelowały o zbiórkę pieniędzy, żeby pomagać najbliższym, którzy popadli w zdrowotne tarapaty. Takie doświadczenie to w każdym przypadku mała wojna. Taki mały konflikt, jaki teraz obserwujemy w Ukrainie. Wtedy liczy się czas, każda chwila.

To tak, jakbyśmy my dzisiaj, patrząc na zmagania Ukrainy, nie wysyłali tam amunicji, nie wysyłali piorunów, nie wysyłali krabów. To jest bezduszność, to jest brak empatii, to jest brak serca. Dziękuję. Pani poseł Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Chciałam podkreślić bardzo ważną rzecz: że rząd Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny rząd po 1989 r. dokonał wielkich, przełomowych zmian w zakresie opieki zdrowotnej i w kontekście podniesienia nakładów finansowych właśnie na opiekę zdrowotną w różnych obszarach.

W ramach tych zwiększonych nakładów wdrożono szereg różnego typu programów, m.in. właśnie ten fundusz. Panie ministrze, mam pytanie w związku z tym.

Czy intensywność prac rady zapewnia efektywne realizowanie roli doradczej i jak wygląda to właśnie z perspektywy Ministerstwa Zdrowia? Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Codziennie tysiące rodzin walczą o życie swoich dzieci. Codziennie wielu dorosłych walczy o swoje życie. Przeżywają codzienne dramaty. Nie stanowią statystyki. To realne sytuacje, problemy, wylane łzy i utracone nadzieje.

Przekazują środki, podejmują walkę. A co w tym czasie robi PiS? Kisi miliardy w Funduszu Medycznym. PiS tłumaczy, że ma czas na wydanie tych pieniędzy. Powiedzcie to tym, którzy czasu nie mają, dla których czas ma konkretny wymiar, dla których czas można kupić często za miliony złotych. Te pieniądze są w budżecie - są one zamrożone, ale są.

Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chyba nie ma na tej sali posła, który nie spotkałby się z taką sytuacją w swoim biurze, do którego by nie przyszli jacyś rodzice czy też inne osoby, ludzie, którzy właśnie proszą o jakieś wsparcie. Do mojego biura wielokrotnie takie osoby przychodziły. Otóż chciałem dopytać, bo z jednej strony są te leki - rzadkie, jednostkowe - z drugiej strony jest kwestia doboru tych leków. Nie jestem lekarzem, więc trudno mi tu coś powiedzieć. Jak to wygląda, ta kwestia właśnie tych leków rzadkich?

Bardzo proszę, pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W ostatnim czasie w szybkim tempie likwidowane są oddziały szpitalne w wielu szpitalach, np. Kowary - ginekologia i położnictwo oraz chirurgia, Strzelin - ginekologia i położnictwo, Ząbkowice Śląskie itd. Szpital w Kowarach świadczył usługi nie tylko dla mieszkańców Kowar, ale dla całego powiatu karkonoskiego oraz tysięcy turystów przebywających w Karkonoszach. W tym szpitalu są lekarze, pielęgniarki, a poziom leczenia i opieki oceniany jest wysoko. Mimo to zapada decyzja o ograniczeniu jego działalności. Szpital wojewódzki w Jeleniej Górze od lat ma zaniżone kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie jest w stanie zapewnić leczenia mieszkańców Kowar, powiatu karkonoskiego i wszystkich potrzebujących turystów. Jak długo trzeba będzie czekać na SOR-ze na udzielenie pomocy w nagłych przypadkach? A tak jest w górach. Mieszkańcy Kowar są bardzo zaniepokojeni decyzją właścicieli szpitala o znacznym ograniczeniu jego działalności - szpitala, który od zawsze był miejscem ich leczenia i opieki medycznej. Brak pieniędzy bądź niewystarczająca ich ilość nie może być głównym powodem ograniczenia działalności. Dlaczego nie bierze się pod uwagę faktu, że działalność szpitala jest podstawowym wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa medycznego, a nie zwykłą działalnością komercyjną? Dlaczego w takich sytuacjach jak ta w szpitalu w Kowarach nie ma wsparcia z Funduszu Medycznego? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Dominika Chorosińska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sytuacja pandemiczna wpłynęła na znaczne pogorszenie zdrowia psychicznego zarówno dzieci, jak i młodzieży. Borykamy się z problemami kadrowymi w obszarze psychiatrii dziecięcej. Moje pytanie do pana ministra: Czy środki z Funduszu Medycznego będą mogły być wykorzystywane na utworzenie dodatkowych centrów psychiatrycznych i szkolenie kadr? Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Krytyka Funduszu Medycznego nie wzięła się znikąd. Największe kontrowersje budzi fakt, że pieniądze z niego nie są w pełni wykorzystywane, za to są zamrażane i przenoszone na kolejny rok budżetowy.

To świadczy o słabości Ministerstwa Zdrowia i złym zarządzaniu. Jeżeli nie wiecie, na co wydatkować niewykorzystane pieniądze na zdrowie i życie Polaków, należałoby zwrócić szczególną uwagę na choroby rzadkie. Odbywa się ona nierefundowanym w Polsce lekiem, którego koszt przekracza aż 9 mln zł.

Rodziców chorego na SMA Wiktorka Szczechowiaka z mojego regionu, z gminy Węgierska Górka ta zmiana kosztować będzie kolejne 700 tys. zł. To kolejna kłoda rzucona pod nogi rodzicom dzieci chorujących na rdzeniowy zanik mięśni. Co stoi na przeszkodzie, żeby niewykorzystane środki finansowe z Funduszu Medycznego wykorzystać na leczenie chorób rzadkich w Polsce? Czy będą (Dzwonek) przewidziane pieniądze z Funduszu Medycznego na terapię genową SMA? Pani poseł Małgorzata Janowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Marcin Duszek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Działania strategiczne dotyczące dodatkowych źródeł finansowania, o których dziś rozmawiamy, wymagają czasu i przede wszystkim spokoju. Spokoju, którego gwarantem od kilku lat dzięki zaufaniu naszych wyborców jest polski rząd. Dzięki temu skutecznie podnosimy nakłady i naprawiamy krok po kroku polską służbę zdrowia. Trudne zadanie, ale pod naszymi rządami, jak widać, możliwe do realizacji. Dziękuję panu ministrowi za dzisiejsze wystąpienie i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, za wprowadzanie spokoju, który dzisiaj pan minister wprowadza, ale przede wszystkim - wizji naprawy systemu służby zdrowia.

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Na 1 tys. osób chorych na razie dopiero 100 osób otrzymuje refundację za lek, a to niewiele, chociaż zgłosili się błyskawicznie wszyscy. Jest to choroba genetyczna, im wcześniej się zadziała, tym naturalnie rokowania są lepsze. Jakie jest stanowisko ministerstwa? Jest oczekiwanie, że to będzie właśnie ten lek. Pytanie dotyczące drugiej choroby, hemoglobinurii. W obydwu sprawach pisałam interpelację. W sprawie hemoglobinurii otrzymałam odpowiedź, że będzie refundowany, ale z tego, co wiem, chyba jeszcze nie jest.

Serdecznie witamy w Sejmie. A teraz głos zabierze pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Przede wszystkim dziękuję za to, że mogę zabrać głos, ponieważ wcześniej byłem akurat na posiedzeniu komisji, gdzie byłem referentem. To będzie służyło, jak powiedział pan prezydent, ochronie dzieci, które do tej pory były pozostawione poza ramami Narodowego Funduszu Zdrowia ze względu na choroby rzadkie lub rzadkie choroby onkologiczne, w tym również właśnie wspomniane schorzenie SMA. Wszyscy przykładaliśmy do tego ogromną wagę, że to jest właśnie to nowe źródło, które daje pewną nadzieję. Proszę się nie dziwić, panie ministrze, słuchałem pańskiej odpowiedzi, która oczywiście wykazuje bardzo wiele elementów dobrej woli z pańskiej strony, ale proszę się nie dziwić, że jeżeli tam jest 3,5 mld zł, a tutaj jest taka presja, jak pan słyszał, z różnych stron na biura poselskie i również na nas osobiście, że pytamy o to, co można w tej materii zrobić, jakie programy państwo macie. Jakie rekomendacje np. ma rada funduszu w tej sprawie? Dobrze byłoby usłyszeć, czy rada funduszu w tej sprawie proponuje jakieś rekomendacje w tej sprawie. Czy państwo również ze strony tego funduszu zechcieliście powiadomić np. szpitale powiatowe?

Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Dariusza Klimczaka. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować każdemu parlamentarzyście, każdej posłance i każdemu posłowi, którzy wzięli udział w tej bardzo ważnej dyskusji. Dziękuję tym, którzy docenili wagę tematu, który poruszamy. Jestem przepełniony nadzieją, że ona zaowocuje dobrymi zmianami, które uratują wiele żyć.

Kiedy fundusz powstał, powstała także nadzieja. Dzisiaj w przypadku każdej choroby liczy się czas. Mówili o tym zarówno poseł Rusiecki, jak i poseł Dyduch. To niezwykle trafne określenie problemu, z którym się stykamy. Mówili o tym poseł Rutnicki, posłanka Rosa, ale także posłanka Płonka.

Procedury dotyczące Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji także należy zmienić. O negocjacjach wspominał pan poseł Jarosław Rzepa. Dziękuję mu za zwrócenie uwagi na tę kwestię, bo uważam, że my, Polacy nie jesteśmy gorsi od innych narodów. Potrafimy negocjować i mam nadzieję, że tę umiejętność posiadają także osoby, które zasiadają w rządzie, pracują w Ministerstwie Zdrowia.

Według zapowiedzi w ramach Funduszu Medycznego ma być finansowana diagnostyka genetyczna i molekularna. To samo zadanie zostało wpisane do działań w Planie dla Chorób Rzadkich, o którym tutaj była mowa. Czy celem projektu jest de facto pokrycie finansowe innych zobowiązań, jakie rząd ma wobec pacjentów? Według zapowiedzi diagnostyka ma objąć tylko populację dzieci. Podczas tej debaty docierało do mnie pytanie, co z dorosłymi. To także jest niezwykle ważny problem, o którym mówią organizacje pacjenckie.

Ono się delikatnie przewinęło w tej dyskusji. Ile do tej pory kosztowało funkcjonowanie tej rady? Ile odbyło się spotkań tej rady? Jaki był efekt ustaleń rady i gdzie ta rada się spotyka? Dotarła do mnie informacja, że były wyjazdowe posiedzenia tej rady. Jakie są przede wszystkim efekty jej pracy? Posłowie zadawali pytanie: Jakie rekomendacje rada wykonywała? Chciałbym prosić o szeroką informację na temat działalności tej rady. Upominamy się o wszystkie dzieci cierpiące na choroby rzadkie, o te dzieci, które z różnych powodów nie mają dostępu do terapii. Te 10 lat, o których tutaj wspomniano. Dzisiaj liczy się każda minuta, każda godzina, każdy tydzień.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym powiedzieć, że padły tutaj dość polaryzujące określenia dotyczące Funduszu Medycznego. Z jednej strony pojawiła się nadzieja, która przebiła się w ostatniej wypowiedzi pana posła Klimczaka, ale pojawiały się również takie zwroty jak ˝fundusz widmo˝ czy nawet ˝zabawka˝

Wydaje mi się, że jednak nie.

Jeśli chodzi o SMA, które bardzo często przewijało się w wypowiedziach i pytaniach państwa posłów, stanowczo i jednoznacznie chcę podkreślić, że wszystkie dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni w Polsce są leczone. Jest to lek Spinraza.

Mało który kraj robi badania przesiewowe na SMA.

Druga kwestia: wyłapujemy, mówiąc kolokwialnie, każdy przypadek tego typu schorzenia, tego typu choroby.

Już mówię, co z VAT-em. VAT był wprowadzony na okres pandemii na wszystkie leki ze zbiórek.

Pozwolę sobie go zacytować: NIK dostrzega wysiłek włożony w zapewnienie organizacyjnego i personalnego przygotowania Ministerstwa Zdrowia do realizacji tych zadań, w szczególności polegających na opracowaniu i przygotowaniu procedur związanych z funkcjonowaniem poszczególnych subfunduszy, przeprowadzaniem procedur naboru do nowo powstałego Wydziału Funduszu Medycznego Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, z czym wiązała się konieczność przeprowadzenia analiz, jak i prac planistyczno-koncepcyjnych oraz kontaktów z interesariuszami. To też trzeba jasno powiedzieć. Nie, działaliśmy na zasadzie: wszystkie ręce na pokład. Wydaje mi się, że warto również ten fakt przytoczyć.

Pozwolę sobie przytoczyć taką ścieżkę, która dotyczy subfunduszu inwestycji strategicznych: przygotowanie dokumentacji konkursowej, kryteria oceny, regulamin konkursów i wzory umów, przeprowadzanie naborów, wnioski, ocena złożonych wniosków, procedura ustanowienia poszczególnych inwestycji w drodze uchwał Rady Ministrów, zawieranie przez Ministerstwo Zdrowia umów z inwestorami, ogłaszanie przez inwestorów poszczególnych postępowań w zakresie wykonawców robót, realizacja robót i dopiero na końcu ponoszenie wydatków przez inwestorów. Proszę państwa, to jest łańcuch, który wymaga niestety czasu. Tak jak mówiłem podczas pierwszej mojej wypowiedzi, procesy inwestycyjne trwają.

Było pytanie dotyczące tego, czy Fundusz Medyczny będzie również kierunkował się na inne obszary wsparcia. Jeśli chodzi o rozwijanie samych subfunduszy, to nie, natomiast w proponowanych przepisach nowelizacji ustawy, która w niedługim czasie, mam nadzieję, zostanie przedstawiona opinii publicznej, mamy zaplanowane rozwinięcie pewnych obszarów. Jeśli chodzi akurat o kadry, te kadry będą finansowane z środków z innych źródeł, podobnie zresztą jak centra zdrowia psychicznego, na co również jest kompleksowy plan, mówiąc kolokwialnie, zazębiający się.

Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Banaszek dotyczące naszych priorytetów w ramach Funduszu Medycznego, jest to onkologia.

Były pytania dotyczące Rady Funduszu Medycznego. Owszem, Rada Funduszu Medycznego, która jest organem ekspercko-opiniodawczym dla Funduszu Medycznego, jest w bezpośrednim i stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i Kancelarią Prezydenta. Te posiedzenia odbywają się regularnie. Mają charakter merytoryczny i ekspercki, podkreślam: merytoryczny i ekspercki, bo pojawiły się odnośnie do tego jakieś sugestie, więc odnoszę się do tego w sposób jasny i bezpośredni. Wszystkie rekomendacje, które wypracuje rada, poddawane są później dalszym dyskusjom nie tylko w ramach kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, ale również w rozmowach z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta.

Było również pytanie dotyczące poziomów i wsparcia szpitali od pierwszego do trzeciego poziomu. Rzeczywiście subfundusz inwestycji strategicznych jest ukierunkowany bardziej na ośrodki referencyjne.

Do tego subfunduszu - za chwilkę, mam nadzieję, się ten konkurs pojawi, jeśli Rada Ministrów przyjmie tę uchwałę - takie szpitale będą mogły aplikować. Była jeszcze kwestia dotycząca negocjacji z producentem leku Zolgensma, bo wrócę jeszcze kompozycją klamrową do początku mojej wypowiedzi. Te negocjacje trwają. Wczoraj zresztą było posiedzenie komisji ekonomicznej, na którym również ten wątek był omawiany. Dlatego proszę się jeszcze wstrzymać w tym zakresie.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349)

Wysoka Izbo! Prezentowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw reformuje, zmienia jeden z elementów istniejącego systemu wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego, a konkretnie zmienia sposób obliczania wypłacanych odszkodowań.

Po pierwsze, każdy wywłaszczony otrzyma nieco więcej, niż wynosi wartość rynkowa jego nieruchomości, czyli otrzyma pewien bonus do wartości tej nieruchomości, z której jest wywłaszczany. W rozumieniu osobistej wartości netto - to pojęcie z dziedziny finansów osobistych - jego osobista wartość netto wzrośnie.

To pierwsza zasada. I to trzeba ustalić: ona jest najważniejsza. Każdy wywłaszczany dostanie nieco więcej, niż wynosi wartość nieruchomości, z której zostaje wywłaszczony. Zasada druga, pomocnicza. Każda szkoda, która w wyniku wywłaszczenia została wyrządzona, każda szkoda, którą wywłaszczany w wyniku wywłaszczenia poniósł, będzie zrekompensowana. Nawet jeżeli ta szkoda z jakiejś przyczyny jest większa niż wspomniana wartość nieruchomości plus pewien bonus. Za przypadek podlegający szczególnej ochronie, który należy stosować ze szczególną wrażliwością, uważamy przypadek, w którym wywłaszczana osoba mieszka na tej wywłaszczanej nieruchomości, czyli kiedy w wyniku inwestycji ktoś zostanie pozbawiony swojego dachu nad głową.

Te trzy zasady to są zarazem trzy zmiany w stosunku do stanu obecnego. Bo jaki jest stan obecny, obowiązujący w Polsce od wielu, wielu lat, niewprowadzany przez ten rząd, stosowany w przypadku wielu dotychczasowych wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego, wywłaszczeń pod autostrady, wywłaszczeń pod inwestycje związane z EURO 2012? W nim podstawą, główną zasadą było to, że odszkodowanie wynosi samą wartość rynkową wywłaszczanej nieruchomości. Nie było tu żadnego bonusu, nie było żadnego dodatku. Po pierwsze, sam fakt, że ktoś przymusowo musi pozbyć się swojej nieruchomości, nie planował sam jej sprzedawać. Jest to pewna dolegliwość trudno wycenialna materialnie, ale niewątpliwie musimy przyjąć, że ona występuje. Po drugie, w przypadku osób, które zamieszkiwały na tej nieruchomości, ta dolegliwość jest znacząco większa. Jest cały szereg dodatkowych kosztów z tym związanych: koszty pośrednictwa w zakresie nieruchomości, koszt obsługi prawnej, koszty przeprowadzki, które w tym systemie, w cudzysłowie, gołego odszkodowania w wysokości wartości rynkowej nie są rekompensowane.

Nie było tego, co wprowadzamy teraz, czyli roszczenia o pokrycie szkody rzeczywistej, gdyby jakieś szkody, chociażby tego rodzaju, o którym tu mówiłem, w wyniku wywłaszczenia się pojawiły. Przytłaczająca większość wywłaszczanych mogła więc czuć się poszkodowana z powodu bycia wywłaszczonym. Ale oczywiście, tak jak każda moneta ma dwie strony czy każdy kij ma dwa końce, była pewna grupa, nieliczna, która dzięki zastosowaniu tzw. zasady korzyści, zasady kuriozalnej i zasadniczo niewystępującej w Europie poza Polską, odnosiła w wyniku bycia wywłaszczonym na inwestycje celu publicznego ogromne zyski. Jaki rodzaj własności był szczególnie preferowany czy szczególnie premiowany w ten sposób przez, było nie było, polskie państwo? Nie własność działalności gospodarczej, nie własność jakiegoś drobnego zakładu rzemieślniczego, nie własność domu czy mieszkania, w którym ktoś mieszka, tylko własność dużych obszarów, dziesiątków hektarów ziemi o niskiej wartości.

Ta zasada była oczywiście absurdalna logicznie i po prostu, po ludzku niesprawiedliwa. Stąd ten wielokrotny, idący w setki procent, nieraz ponad 1000%, zysk dla nielicznych w wyniku bycia wywłaszczonym na inwestycje celu publicznego zniknie z systemu prawnego, nie będzie więcej funkcjonował, za to wszyscy dostaną więcej niż wynosi wartość rynkowa ich nieruchomości.

To jest ta podstawowa zmiana. Ona dotyczy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, jak również całego szeregu specustaw inwestycyjnych, wszystkich ustaw, które regulują zasady wywłaszczeń i wycen tych wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego. W ustawie poza tym znajdują się przepisy dotyczące już tylko Centralnego Portu Komunikacyjnego, ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Chcemy tu zaproponować rozwiązania, które pozwolą oferować mieszkańcom w ramach programu dobrowolnych nabyć korzystniejsze niż do tej pory warunki dobrowolnego wykupu nieruchomości.

Można np. siać, zbierać plony z tej nieruchomości, można ją wykorzystywać w swojej działalności rolniczej. Dotyczy to specyficznej grupy rolników, którzy - tak wynika z konsultacji społecznych, z rozmów, z postulatów strony społecznej - są już blisko wieku emerytalnego, nie są najmłodsi i sprzedają swoją nieruchomość.

Podkreślam, żeby też dobrze to zrozumiano, iż mówimy tu nie o rencie w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych, tylko o rencie w rozumieniu prawa cywilnego, zobowiązania cywilno-prawnego.

Szanowni Państwo! Jeszcze jedna uwaga do tej ustawy. Jak państwo tutaj już słyszeli, jak mówiłem, ona jest korzystna dla wszystkich, dla ogółu społeczeństwa, natomiast jest pewna wąska grupa osób, która na nim straci. Taka osoba straci w tym sensie, że zamiast dostać 700%, 800%, 1000% wartości swojej nieruchomości, zamiast na byciu wywłaszczonym 10-krotnie się wzbogacić, dostanie 120% np. wartości nieruchomości i środki na pokrycie szkody. Mówimy tu o kwotach idących w miliony i dziesiątki milionów. Wiem, że są specjalne organizacje, powiedzmy, że są one społeczne, które wspierają te kancelarie. Wiem, że one wysyłają do państwa posłów pisma. Czytając zapytania, interpelacje, czasem widzę w nich jednobrzmiące sformułowania żywcem wyjęte z pism tych organizacji. Bardzo proszę tu o ostrożność i rozwagę.

Bardzo proszę państwa posłów, żebyście podchodzili do tego rodzaju głosów z krytycyzmem, ze zdrowym rozsądkiem i oceniali, czy warto godność, powagę posła Rzeczypospolitej angażować w ochronę tego rodzaju interesów. Wysoka Izbo! Przedstawiana ustawa moim zdaniem stanowi kwintesencję tego, czym powinna być polityka publiczna. Powinno chodzić tu o popieranie nie wąskich grup interesu, ale ogółu społeczeństwa, o wprowadzanie w życie zasad sprawiedliwości społecznej, ale też, można powiedzieć, sprawiedliwości bezprzymiotnikowej, po prostu sprawiedliwości, o to, żeby był realizowany interes publiczny polegający na tym, żeby pewne dobra publiczne dostarczać wszystkim, np. drogi, linie kolejowe, lotnisko, sieci przesyłowe energetyczne, gazociągi, rurociągi, całą infrastrukturę, która nam wszystkim potrzebna jest do życia, i jednocześnie równoważyć to interesem, dobrem danej jednostki, danej osoby, która gdzieś ma kawałek gruntu, która gdzieś ma dom. Gdzieś trzeba takie obiekty budować, gdzieś trzeba je lokalizować. Odbywać się to będzie zawsze zgodnie z przepisami konstytucji, za słusznym odszkodowaniem, godziwym, nieco większym - podkreślam: nieco, ale większym - od wartości rynkowej tej nieruchomości.

Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie przedłożonej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zaprezentować nasze stanowisko wobec przedłożenia rządowego zawartego w druku nr 2349.

Pan minister tutaj przytoczył niektóre przykłady. Powtórzę. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości zamieszkałych i przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności zakładu, fabryki, wysokość odszkodowania stanowi wyłącznie wartość nieruchomości. Ona pomija - co było niejednokrotnie argumentowane - koszty przeprowadzki, koszty nabycia nowej nieruchomości, koszty przeniesienia działalności gospodarczej czy też odtworzenia produkcji rolniczej. Tak samo pan minister zwrócił uwagę, iż w dotychczasowym reżimie prawnym rolnicy nie otrzymują dzisiaj żadnej dodatkowej rekompensaty z tytułu utraty tej nieruchomości, która jest ich miejscem pracy. Z kolei w przypadku wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, komercyjną odszkodowania odpowiadają wyłącznie wartości rynkowej gruntów. Przechodząc teraz do proponowanych przez rząd regulacji, które Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście popiera, przede wszystkim podkreślę to, iż celem projektowanych zmian jest usunięcie tej społecznej niesprawiedliwości występującej w aktualnie obowiązującym systemie odszkodowań i odwołanie się szerzej do praktyki europejskiej szeroko stosowanej w wielu państwach naszego kontynentu. Chodzi o zastąpienie tej istoty, czyli zastąpienie zasady korzyści, nowymi regulacjami, które mają charakter taki, iż zapewniają słuszne odszkodowanie, również w takim zakresie, że przede wszystkim zdecydowanie bardziej respektują równość podmiotów wywłaszczonych wobec prawa, która się przejawia w powiązaniu wysokości odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości, z uwzględnieniem szczególnych sytuacji, zwłaszcza dotyczących wywłaszczenia nieruchomości mieszkaniowych. Pan minister już wcześniej wskazał, iż w tej nowej regulacji rząd rekomenduje następującą praktykę, aby do wartości nieruchomości w każdym przypadku był dodawany bonus pieniężny, który stanowiłby zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, realizacji czynności prawnych, które dotychczas nie były refundowane.

W przypadku obiektów budowalnych ten bonus wzrasta do 20% wartości lokalu powyżej wyceny, która oczywiście jest dokonywana według wartości rynkowej, na podstawie operatu.

Będzie mógł z tego skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie powoduje zawsze, w każdym przypadku, również w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego, wysokie szkody, których ta klasyczna, podstawowa skala 10% może nie pokryć. Można tutaj z naszej strony (Dzwonek) jeszcze dodać szereg innych argumentów. Ale raz jeszcze powtarzam, iż Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera rekomendowane zmiany zawarte w tym projekcie. Dziękuję za uwagę. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Gdy czytamy uzasadnienie tego projektu ustawy, która zmienia cały system, jak już było tu wspomniane, przede wszystkim odszkodowań w przypadku przymusowych wywłaszczeń, wyłania się nam nowy, wspaniały świat, taki z lekka orwellowski, tylko szczęśliwych ludzi, którzy są obdarowywani przez państwo większą dozą estymy i większym wynagrodzeniem, niż na to zasługują. Tylko nie wiedzieć czemu protestują w całej Polsce. Wprawdzie ustawa dotyczy regulacji w ogóle, ale z niej wyłania się pazerne, chciwe państwo, które nie liczy się z ludźmi, które nie liczy się z własnością, które nie liczy się z tradycją i kulturą, i trwałością siedlisk. A co sprawiło, jaka okoliczność, że w tej chwili regulujemy cały system w taki sposób, budzący trwogę u obywateli? Oto, co to sprawiło - nowy wspaniały świat ministra Horały trojga posad, który pokazuje nam świetlaną przyszłość i który wyzuwa z siedlisk i z własności na taką skalę, która w historii Polski nigdy nie miała miejsca. Szacuje się, że jest to ok. 20 tys. ha na megalotnisko z megadeweloperką wokół plus szprychy tzw. kolejowe. Na mapie wygląda to tak, jak gdyby gospodyni zabrała się do kapusty i ją dokumentnie posiekała, łącznie z ludźmi, którzy na tej ziemi są.

Tak się składa, że sprawiedliwe i słuszne odszkodowanie, zgodne z naszymi konstytucyjnymi zasadami, proponował, czy tylko wymusił, Bank Światowy, który finansował np. inwestycje przeciwpowodziowe. Jako klub Koalicji Obywatelskiej będziemy wnosili, skoro mamy do czynienia z systemowym rozwiązaniem, o wprowadzenie tej reguły, która pozwala na odtworzenie siedlisk, która pozwala na słuszne i sprawiedliwe traktowanie obywateli - będziemy wnosić o wprowadzenie tego do tej ustawy, do polskiego porządku prawnego. Oczywiście jeśli chodzi o tę ustawę, o to rozwiązanie w tej chwili - które jeszcze reguluje wszystkie inne specustawy, bo w Polsce mamy te kwestie rozproszone - będziemy wnosili o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu i zabranie się za rzeczywiste, sprawiedliwe i zgodne z konstytucją regulacje, które wymuszą partnerskie i pełne szacunku traktowanie swoich obywateli. Ja nie chcę się tu wypowiadać, bo nie jest to przedmiotem dzisiejszej debaty, na temat kwestii zasadności tego projektu, ale mówię o zasadności i sprawiedliwości traktowania obywateli. I proszę nie żonglować znaczeniem słów, bo zasada korzyści nie mówi o żadnych korzyściach, tym bardziej tych niesłusznych, o których pan mówi i zarzuca manipulację innym. Wartość rynkowa nie jest wartością rynkową tak naprawdę i nie pozwala na odtworzenie nieruchomości, bo wartość odtworzeniowa to jest minus zużycie, także robocizny.

W związku z tym wnosimy w imieniu Koalicji Obywatelskiej wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, a jeśli on nie znajdzie uzasadnienia, poparcia w Wysokiej Izbie, będziemy wnosić w drugim czytaniu przede wszystkim o wysłuchanie publiczne, bo to się Polkom i Polakom należy w tej sprawie.

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Witamy serdecznie w Sejmie. Bardzo proszę, pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy zakładają zreformowanie obszaru regulacji dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w celu zapewnienia zgodności w wyższym niż obecnie stopniu z zasadą słusznego odszkodowania określoną w przepisie art. 21 ust. 2 konstytucji. Najważniejsze rozwiązania to odszkodowanie za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycję celu publicznego. Do takiej wartości dodany będzie bonus pieniężny, który wyniesie bazowo 10% wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 20% dotyczyć będzie wartości budynku zlokalizowanego na nieruchomości oraz wartości lokalu mieszkalnego. Bonus pieniężny będzie zryczałtowanym ekwiwalentem kosztów przeprowadzki i czynności prawnych. Aby zapewnić słuszny charakter odszkodowania, przewidziane zostały dodatkowo dwa zabezpieczenia dla osób wywłaszczonych. Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym, niż to wynika z odszkodowania, a jeżeli wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, przysługiwać będzie zwiększenie tego odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej. To dość dobrze wyglądające założenia i sama idea wydaje się słuszna, gdyby nie fakt, że ustawa ta dotyczy m.in. inwestycji budzącej tak ogromne społeczne, gospodarcze i finansowe kontrowersje.

Mieszkańcy Baranowa i innych okolicznych miejscowości zwrócili się nawet o pomoc do rzecznika praw obywatelskich. Nie przeprowadzono bowiem analiz środowiskowych, w tym przede wszystkim w sprawie hałasu związanego z funkcjonowaniem ogromnego portu lotniczego. Jak czytamy w sprawozdaniu rzecznika praw obywatelskich, właściciele działek, którymi interesuje się CPK, skarżą się na iluzoryczny charakter przeprowadzanych konsultacji społecznych oraz brak wiarygodnych informacji. Nie jest nadal znany zasięg oddziaływania różnych uciążliwości związanych z planowanym lotniskiem. Zdarza się, że na teren nieruchomości znajdującej się w obszarze wstępnie zapowiadanych wywłaszczeń pod CPK bez zgody właścicieli wchodzą przedstawiciele inwestora, aby przeprowadzić inwentaryzacje przyrodnicze. Wywołuje to uzasadnione obawy mieszkańców co do podstawy prawnej wejścia na ich grunt, zwłaszcza że bez zgody właścicieli sporządzana jest dokumentacja fotograficzna działek i zabudowań, czytamy w dokumencie przedstawionym przez rzecznika praw obywatelskich. Zdaniem RPO działania związane z procesem nabyć i wywłaszczeń pod budowę wystawiają na szwank naczelną zasadę zaufania obywatela do państwa. Zakładane w ustawie odszkodowania będą miały charakter swoistego rodzaju ryczałtu, który będzie składał się w części odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości i bliżej niezdefiniowanej górki lub - jak chcą autorzy tego projektu - tzw. bonusu. Projektowane zmiany budzą mnóstwo wątpliwości natury społecznej i prawnej. W szczególności aktualne może być postawione pytanie: Czy odszkodowanie oparte na modelu ryczałtu jest zgodne z konstytucyjną zasadą, która uprawnia właściciela wywłaszczonej nieruchomości do odszkodowania odpowiadającego słusznemu wynagrodzeniu? Wątpliwości te budzą i będą szczególnie uzasadnione w przypadku wywłaszczanych nieruchomości nabytych w celach inwestycyjnych. Projektowane zmiany nie wprowadzają również dostatecznych mechanizmów, które pozwoliłyby na rzetelną ocenę rzeczywistej szkody poniesionej przez właściciela nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia. Wprawdzie projekt nowelizacji ma uruchomić ścieżkę sądowej kontroli prawidłowości wysokości odszkodowania, jednak zgodnie z deklaracją autorów nowelizacji roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości wywłaszczanych mają zostać ograniczone wyłącznie do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej. Eksperci mają co do tego mnóstwo wątpliwości. Nawet żeby nie wiem jak pan kręcił i (Dzwonek) owijał w bawełnę, fakty są takie, że macie manię stawiania sobie wielkich pomników w imię manii wielkości, które historia - głęboko w to wierzę - odpowiednio oceni. A ta kontrowersyjna inwestycja jest już potężnym kosztem, którego ciężar bez względu na wysokość odszkodowań przenosicie na społeczeństwo, które wam tego nie zapomni. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Tomczak, Koalicja Polska.

Boże mieszkańcom podrzeszowskiej Jasionki i innych miejscowości, przez które wytyczył pan minister szprychy rozmaite tego wielkiego projektu! Polska, wielki projekt, który realizujecie z jednej strony tak, że ciągnie się to latami, a jeszcze nie nabrał jakichś rzeczywistych konturów poza, rzecz jasna, wydrukami z kont zatrudnianych urzędników, a z drugiej strony zdążyliście już zaalarmować całą Polskę, postawić mieszkańców wielu miejscowości wobec perspektywy transformacji, a może rewolucji w ich życiu. W teorii zdaje się proponowanie rozmaitych wariantów przebiegu tych tras miało jakoś odprężać tę sytuację.

Pasjonują nas technika i technologia przyszłości, lotnictwo, kolejnictwo, byle prędkie.

Podrzeszowska Jasionka, Zamość po sąsiedzku na Lubelszczyźnie, Izbica, w Krasnymstawie bunt już całkiem nieźle zorganizowany. To jest niepokojące, że zmierzacie do celu, który jest oczywiście tak szczytny, że stanowi rodzaj szantażu moralnego wobec nas. Każdy, kto będzie kwestionował jego zasadność, ten właśnie wkłada kij w szprychy nomen omen i nie idzie z postępem. Po prostu nie szanujecie prawa własności. Nie chcecie z ludźmi negocjować, nie chcecie się z nimi spotkać, nie chcecie zaproponować im godziwej wypłaty za bardzo często ruinę życia, które dopiero zbudowali, np. przyjeżdżając z zagranicy, repatrianci z Zielonej Wyspy postanowili jednak postawić na Polskę, tu wychować dzieci i teraz mają to wszystko stracić. Bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Natomiast, nie zmieniając swojego zdania na temat CPK czy innych pałaców pychy budowanych przez PiS, muszę powiedzieć, że ta ustawa idzie w pewnym sensie w stronę uporządkowania i uczytelnienia systemu odszkodowań.

Dlatego też ten założony system, który tu jest, racjonalnie porządkuje system odszkodowań - to trzeba przyznać. Są czasem trzy kompletnie różne operaty. Wprowadza dobre wzorce z krajów zachodnich i to widać w uzasadnieniu tego projektu. Zapobiega nadużyciom, więc chroni w pewien sposób interesu podatników, ale też próbuje, przynajmniej wychodzi naprzeciw sprawiedliwemu i godnemu podejściu do interesów właścicieli, chociaż tutaj mamy poważne zastrzeżenia, bo będziemy składać poprawki, które ten interes właścicieli o wiele bardziej uwzględnią. uwzględniając też - i to jest faktycznie nowość - inne straty, otwierając drogę do roszczeń przed sądem, a więc w domyśle też możliwość układania się, ugód ze Skarbem Państwa co do innych kosztów, np. właśnie przestojów w produkcji. Ta ustawa również, i to jest na jej plus, zauważa sytuację osób w nieruchomościach o bardzo niskiej wartości, tzw. babinki w chatynce. Jest mnóstwo takich osób, które już w tej chwili np. na wywłaszczanych rezerwach pod drogi. Abstrahując od CPK, już w tej chwili ten problem bardzo często występuje. Ten mechanizm mówi, że korzystniejszy wariant wybiera się automatycznie, to znaczy, że te osoby nie muszą się procesować, bić o to, tylko one to dostaną. Oczywiście tyle w teorii. Natomiast, jak podkreślano na tej sali, cała ta inwestycja, cały CPK jest bardzo wrażliwym społecznie i kontrowersyjnym projektem.

Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Zamykam listę. Bardzo proszę, jako pierwszy pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw to projekt, który dotyczy wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości na różnego typu inwestycje. Panie ministrze, bardzo bym prosił o pisemną odpowiedź na pytanie, jaka kwota przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań w 2022 r. i jaka część tej kwoty dotyczy odszkodowań związanych z realizacją CPK.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pewnego dnia przychodzi do obywatela pismo i w jednej chwili odbiera obywatelowi wspomnienia z dzieciństwa lub plany na przyszłość związane z tym konkretnym miejscem. Urzędnik tak zdecydował i nasze plany nie mają znaczenia. Otrzymujemy zadośćuczynienie, które zazwyczaj nie jest satysfakcjonujące. Kupujemy mieszkanie lub inny dom, budujemy nowe plany na przyszłość i w pewnej chwili otrzymujemy kolejną wiadomość, że nastąpiła zmiana, że nie będzie wywłaszczenia, że możemy jednak zostać w swoim domu, tylko że musimy szybko oddać otrzymane pieniądze. Czy w takich sytuacjach konsekwencjami błędnych decyzji nie powinien być obarczony podmiot winny tej sytuacji? Mało tego, projekt przewiduje ściganie w takich sytuacjach spadkobierców, osób, które być może nigdy nie wiedziały o wypłacie takiego świadczenia. Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Niemczyk, Koalicja Obywatelska. Pani poseł Ewa Kołodziej, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami to skandaliczne rozwiązanie. Powstał on tylko i wyłącznie na potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który od początku budzi ogromne emocje i wiele kontrowersji. Do mojego biura poselskiego zgłaszane są liczne prośby od mieszkańców o pomoc w zaniechaniu tak szkodliwych działań ze strony rządu. Fakt przymusowego pozbawiania ludzi nieruchomości, domów, miejsc pracy na tak ogromną skalę oraz skutki, które on wywoła, są dla nich niewyobrażalne. Dodatkowo z przedstawionego projektu wynika, iż odszkodowania za przymusowe wywłaszczenia będą skrajnie zaniżone i niekorzystne dla osób pozbawionych swojego majątku. Zatem zwracam się do autora zmian tych przepisów pana Marcina Horały z pytaniami. Dlaczego nie szanuje pan art. 21 konstytucji, który mówi o słusznym odszkodowaniu w przypadku wywłaszczenia na cele publiczne? Dlaczego przepisy w zakresie wywłaszczeń w obecnym brzmieniu są korzystne tylko i wyłącznie dla inwestora? Czy naprawdę CPK musi być realizowane tak ogromnym kosztem społecznym? Nie ma pana posła. Pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! To, co robi pan, panie ministrze, jest skandaliczne. Pierwszym skandalem jest to, że to właśnie pan przygotowuje ten projekt ustawy, a jest pan osobą osobiście odpowiedzialną za to, żeby na CPK i te megalomańskie 10 szprych wydać jak najmniej. A drugim skandalem jest to, w jaki sposób pan mówi o dotychczas obowiązujących przepisach, z których może wynikać, że osoby, które obawiają się o utratę swojego dorobku życia, są jakimiś cwaniakami, bo mają się dorobić w jakiś szczególny sposób na tych wywłaszczeniach. Czy jest pan w stanie powiedzieć - nie, pan dobrze wie - czy przykładowy właściciel gospodarstwa ogrodniczego w podłódzkich Brzezinach nie znajdzie podobnego gospodarstwa za pieniądze, które od was otrzyma, i nie wybuduje nowego?

Dziękuję bardzo. Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Jest to działanie siłowe, powiedziałabym brutalne, bo pozbawia się właścicieli ich własności wbrew ich woli. Dlatego, szanując konstytucję, należałoby dołożyć wszelkich starań, aby to działanie było jak najmniej bolesne dla właścicieli, bez poczucia krzywdy. Tymczasem rząd skupia się głównie na tym, aby jak najtaniej, jak najszybciej nabyć nieruchomości do spółki CPK, bo to głównie o to chodzi, mamiąc ludzi bonusami. To jest absolutnie pułapka. Ludzie nie dadzą się na to nabrać, bo to jest dla nich krzywdzące. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Będziemy przypominać konstytucję, bo w art. 21 postanowiliśmy, że Rzeczpospolita chroni własność i prawo dziedziczenia. Przejrzałem konstytucję. Tu nie ma nic o ochronie najbardziej wymyślnych projektów inwestycyjnych takiego czy innego rządu. Ma pan pecha, bo mógł pan się zabrać za budowanie kolei dużych prędkości, portu lotniczego wtedy, gdy mieliśmy deflację, dziś mamy inflację. Propozycja, z którą pan przyszedł do Wysokiej Izby, nie gwarantuje aktualnym właścicielom, że w wyniku odszkodowania, które pan proponuje, będą mogli odtworzyć posiadane nieruchomości. Dowód? Wczorajsza ˝Polityka˝ i artykuł. Dlaczego nie zostały podpisane kontrakty drogowe? Dlatego że wykonawcy ocenili, iż ponieśliby straty na poziomie 25-30%. Pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jeżeli ma być tak pięknie, jak pan mówi, po wprowadzeniu tej ustawy, to dlaczego mieszkańcy Baranowa i Wiskitek panu nie wierzą?

Nie ufają wam. Zmieniamy zasadę definiowania konstytucyjnego pojęcia słusznego odszkodowania za naruszenie chronionego w ustawie zasadniczej prawa do własności, własności nieruchomości, które stanowią fundament dobrobytu Polaków. Dlaczego przedmiotem dyskusji nie jest redefiniowanie odszkodowania w sposób, który zagwarantuje odtworzenie stanu posiadania? Polski system opiera się na wartości rynkowej. Ustawodawca założył, że wywłaszczony ma prawo odkupić podobną nieruchomość, ale po tym, po takich masowych wywłaszczeniach (Dzwonek), te nieruchomości będą znacznie droższe i nawet przy 20% bonusu nie będzie można ich kupić w danej okolicy. Dziękuję bardzo. Pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałabym na konkretnym przykładzie pokazać, jak wspaniale traktujecie Polaków.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówimy o dorobku życia ludzi, czasami dorobku wielu pokoleń. Panie ministrze, trochę pokory. Chciałem pana zapytać, czy miał pan odwagę stanąć przed mieszkańcami Katowic, Mikołowa, i skonsultować z nimi tę propozycję. Odbyły się spotkania, miał pan szansę. Ci ludzie boją się, że za te pieniądze za tydzień czy za dwa nie będą mogli wybudować sobie domów, że nie będą mogli znaleźć sobie miejsca na ziemi, w Polsce, bo ceny galopują, inflacja galopuje, a pan tutaj daje (Dzwonek) malutki bonusik dla tych ludzi, którzy tracą dorobek życiowy. Dziękuję bardzo.

Proszę przybyć i być wyposażonym w dokumentację tej szprychy na tym odcinku. Proszę skonfrontować się z rzeczywistością.

Ma pan zaproszenie na posiedzenie zespołu parlamentarnego.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak w tym projekcie zabezpieczycie państwo kwotowo osoby, których nieruchomości zostaną zabrane pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, osoby z gminy Baranów, gminy Teresin, gminy Wiskitki, ale też z tych miejscowości, przez które będą przechodziły szprychy? Wywłaszczenie to naprawdę bardzo trudny i wrażliwy temat. Jak państwo zrekompensujecie to ludziom? To są też straty moralne. To dorobek życia tych ludzi od wielu, wielu pokoleń. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ta ustawa to dowód waszej arogancji lub niekompetencji, zależy, z której strony na to spojrzeć. Panie Ministrze! Czy jest pan w stanie stanąć w prawdzie i przyznać, że próbujecie stworzyć sobie furtkę do łatwiejszego wywłaszczania własności ludzi pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego? Prawo obowiązuje na terenie całej Polski, a nie tylko tam, gdzie zechce tego pan minister Horała. Brzmi to bardzo pięknie, ale czy nie widzicie, że te same przepisy znajdą zastosowanie w przypadku, gdy deweloper wykupi ziemię pod budowę mieszkań, a gmina będzie musiała go wywłaszczyć np. pod budowę drogi? Nowe, zwiększone odszkodowanie nie trafi z budżetów samorządów do ludzi, ale do kieszeni deweloperów. W mniejszych miasteczkach może to doprowadzić do kuriozalnej sytuacji, gdzie odszkodowanie będzie większe niż budowa całej inwestycji. Panie Ministrze! Czy to błąd, czy świadomie wspieracie deweloperów? Jak zamierzacie temu zapobiec? Ustawa w tym kształcie jest zwykłym bublem, który natychmiast trzeba wyrzucić do kosza.

Koszty tej inwestycji i wynagrodzenie dla zarządu CPK rosną szybciej niż trawa na łące w Baranowie. Przestańcie budować na ludzkiej krzywdzie. To było ostatnie pytanie. Bardzo proszę.

Inwestują w państwa, docierając do państwa, a państwo w ogóle.

Bardzo proszę, czy mogę prosić o spokój na sali.

Natomiast stworzenie organizacji, która zatrudnia ekspertów, której eksperci występują w mediach, którzy piszą pisma, ja też te pisma dostaję. Dostaję pismo od organizacji, a potem dostaję od państwa pismo, które jest słowo w słowo przepisane z pisma tej organizacji. No więc w tym sensie inwestują swój czas i swój wysiłek w dotarcie i wykreowanie tego rodzaju tez. Szanowni Państwo! Dlatego protestują, tak jak przy każdej inwestycji. Proszę mi wskazać inwestycję, np. budowę autostrady za czasów Platformy Obywatelskiej, co do której nie byłoby protestów. Oczywiście tych budów było mniej i one przebiegały znacznie wolniej, więc łączna zebrana suma, masa krytyczna tych protestów była mniejsza, to prawda. Bo rozmach inwestycji był mniejszy. Proszę o spokój, pan minister. No cóż, pozostaje mi się tylko nie zgodzić z tymi tezami. Wartość rynkowa to jest wartość rynkowa, a zasada korzyści to jest zasada korzyści. Zabrakło mi jednego argumentu.

Tego po prostu nie rozumiem i dziwię się państwu, że swoją twarz, swoje nazwisko dajecie obronie tego rodzaju rozwiązań. Pani poseł Karolina Pawliczak z Lewicy mówi, że nie przeprowadzono analiz środowiskowych i jednocześnie trzy zdania później mówi, że mieszkańcy są zaniepokojeni tym, że pracownicy inwestora wchodzą na ich nieruchomości, żeby przeprowadzić badania środowiskowe. No to albo to, albo to. To już chociaż proszę nas nie oskarżać o dwa zupełnie sprzeczne działania jednocześnie. Tak, są wykonywane badania środowiskowe: 14 miesięcy w przypadku samego lotniska i węzła i mniej więcej ponad rok w przypadku każdej innej inwestycji, już nawet nie setki, ale tysiące przyrodników. One wszystkie będą miały odzwierciedlenie w raporcie oddziaływania na środowisko, który będzie załączony do wniosku o decyzję środowiskową. Więc naprawdę bardzo proszę nie powtarzać tutaj ewidentnych, łatwo weryfikowalnych kłamstw, że nie są prowadzone analizy środowiskowe. Zresztą żadna inwestycja bez takich analiz nie może powstać, po prostu. Takie jest prawo w Polsce. Przecież nie wynagrodzenia oparte na ryczałcie, tylko bonus 10 lub 20% do wynagrodzenia opartego na wartości rynkowej, operat szacunkowy, tak jak i obecnie. Jeżeli obecnie ktoś dostaje samą wartość rynkową, sam operat szacunkowy, a dostanie operat szacunkowy plus 10 lub 20%, to jak można mówić, że straci na tym rozwiązaniu, jak dostanie o 10-20% więcej, niż dostawał wcześniej? Ograniczenie wyłącznie do szkody rzeczywistej, i to jest merytoryczny głos. Dlaczego to prawo roszczenia ograniczamy do szkody rzeczywistej, a nie do utraconych korzyści? Utracone korzyści to są przyszłe pożytki z prowadzenia działalności czy użytkowania w jakiś sposób danej nieruchomości. Jeżeli ktoś dostaje odszkodowanie, które pokrywa wartość tej nieruchomości, plus jeszcze pewien bonus, to założenie jest takie, że może nabyć sobie podobną w charakterze nieruchomość i wtedy z tej nowej nieruchomości czerpać pożytki mniej więcej takie same jak z tej starej.

Zresztą pojęcie utraconych korzyści jest bardzo nieprecyzyjne, podlegające bardzo daleko idącym różnicom interpretacyjnym i wprowadzenie takiego roszczenia odszkodowawczego do systemu prawnego powodowałoby cały szereg problemów i nieprawidłowości w sądach, więc oparcie o operat szacunkowy, wartość rynkową i szkodę rzeczywistą - dobrze zdefiniowane pojęcie w prawie jest znacznie lepsze. Natomiast znów, jak się jest. Bo państwo krytykują, np. państwo przedstawiciele posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, ale też Lewicy. Lewica też w Polsce rządziła, wtedy kiedy te przepisy już obowiązywały. Więc państwo nas oskarżacie, że danie prawa do dochodzenia szkody rzeczywistej to jest za mało, to jest źle, jeszcze utraconą korzyść, natomiast państwo, jak rządziliście, mieliście większość w Sejmie, mieliście możliwość uchwalania zmian, to nie daliście jakoś tych utraconych korzyści, ba, nawet nie daliście szkody rzeczywistej, tak jak my chcemy dać prawo do jej dochodzenia.

Tego wymaga prawo, tak się prowadzi proces inwestycyjny. Najpierw studium korytarzowe, które podlega konsultacjom, w którym przedstawiane są korytarze, w których będą się mieścić poszczególne przebiegi, potem, i to jest obowiązek inwestora, trzeba wyznaczyć kilka przykładowych przebiegów, po to żeby każdy z tych przebiegów móc bardzo dokładnie zbadać pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym, przekalkulować. To się nazywa analiza wielokryterialna. Trwa to rok, nieraz 2 lata w przypadku niektórych inwestycji, po to żeby z tych przebiegów wybrać optymalny, który różne aspekty równoważy w taki sposób, żeby ewentualne szkody społeczne, koszty i szkody dla środowiska były możliwie jak najmniejsze. To jest zresztą bardzo dobra praktyka, pozwalająca na wybranie optymalnego przebiegu. Otóż nic bardziej mylnego.

To korzyść 2 godzin, a nie minut, jak był łaskaw powiedzieć pan poseł. Znów nic bardziej mylnego.

Program inwestycyjny CPK, pomijając wszystkie jego aspekty, jest również największym w historii Polski programem konsultacji społecznych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Samorządy również prowadzą inwestycje celu publicznego. Nie wiem, czy z aż taką szczegółowością uda się zagregować i zebrać te dane. Obecnie jesteśmy wyłącznie na etapie dobrowolnych rozmów i ewentualnych dobrowolnych umów cywilnoprawnych.

Zmieniamy tylko zasadę wyliczania wynagrodzenia czy odszkodowania. Mówił o sytuacji, w której po wywłaszczeniu z nieruchomości odstąpiono od realizacji inwestycji celu publicznego i osoba, która dostała odszkodowanie, teraz ma zatrzymać tę nieruchomość i zwrócić odszkodowanie. Otóż tak się nie dzieje. Faktycznie, jeżeli inwestycja celu publicznego, na którą dokonano wywłaszczenia, nie została zrealizowana, osobie wywłaszczonej przysługuje prawo - ale prawo, nie obowiązek, może z niego skorzystać lub nie - zwrotu tej nieruchomości, z której została wywłaszczona. To jest decyzja własna tej osoby, która wywłaszczeniu podlegała, w sytuacji gdy cel wywłaszczenia nie został zrealizowany.

Jest słuszne, czyli odpowiadające społecznemu przeznaczeniu prawa własności i odpowiadające poczuciu sprawiedliwości.

Ktoś traci własność, dostaje za to odszkodowanie w wysokości jej wartości plus pewne wynagrodzenie za dolegliwości, szkody, dodatkowe koszty, które w wyniku tego wywłaszczenia poniósł, czyli ani nie traci, ani też oczywiście się wielokrotnie nie wzbogaca. Obydwa te rozwiązania trudno byłoby uznać za słuszne w myśl przepisu konstytucji.

To wszystko dodatkowe koszty, dodatkowa szkoda. Dzięki naszym zmianom będzie miał prawo do ich pokrycia, a w dotychczasowym reżimie prawnym nie miałby takiego prawa i nie dostałby tych środków. Pani poseł Zofia Czernow mówi, że ludzie nie dadzą się nabrać, bo to jest dla nich krzywdzące.

Pan poseł Cezary Grabarczyk przyniósł konstytucję na trybunę. Faktycznie, jest to system oparty nie na wartości odtworzeniowej, tylko na wartości rynkowej - tak jak system, który obowiązywał, podczas gdy pan był ministrem, realizował inwestycje infrastrukturalne i przeprowadzał wywłaszczenia na inwestycje celu publicznego. Wtedy też pan nie oferował wartości odtworzeniowej. Tak samo nie jest ona oferowana w Niemczech, we Francji, Włoszech, w Portugalii, na Litwie, w Bułgarii, Holandii i przytłaczającej większości innych państw Unii Europejskiej. System oparty na wartości rynkowej jest dominujący. Na drugim miejscu jest wartość podatkowa albo katastralna, której w Polsce nie mamy. Tak, były konsultacje.

Dziękuję uprzejmie za zaproszenie na posiedzenie zespołu parlamentarnego.

Pani poseł Bożena Żelazowska pyta, jak zabezpieczymy kwotowo osoby wywłaszczane, jak zrekompensujemy to ludziom.

Zachęcam do skorzystania z programu dobrowolnych nabyć. Można negocjować. Można przyjąć cenę lub jej nie przyjąć, jeżeli jest niesatysfakcjonująca.

W dyskusji zgłoszono wniosek. Bonus za szybsze wydanie jest i pozostanie. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy na następnym posiedzeniu Sejmu.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda o przedstawienie uzasadnienia projektu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku nr 2335, który ma na celu uregulowanie w Kodeksie pracy możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej oraz możliwości przeprowadzania przez pracodawców samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Jeśli chodzi o pracę zdalną, to jest ona świadczona przez pracowników w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 na podstawie przepisów specustawy COVID-owej z 2020 r. W ciągu ostatnich ponad 2 lat pandemii zarówno pracownicy, jak i pracodawcy chętnie korzystali z pracy zdalnej wprowadzonej specustawą, dostrzegając jej zalety.

Z uwagi na fakt, że praca zdalna przewidziana w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś nadzwyczajnych, jakimi jest sytuacja COVID-owa, konieczne było wypracowanie regulacji, które zabezpieczałyby interesy obu stron stosunku pracy. Dlatego też podjęliśmy pracę wspólnie z partnerami społecznymi zarówno w zespołach Rady Dialogu Społecznego, jak i na plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania. Można się spodziewać, że uregulowanie na stałe tej formy wykonywania pracy może zachęcić większą liczbę pracowników do jej świadczenia w miejscu zamieszkania z uwagi na większą dostępność pracy, którą można będzie wykonywać poza zakładem pracy, np. w miejscu zamieszkania, łącząc pracę z opieką nad osobami niesamodzielnymi, czy też na inne rozwiązania, które w tej sytuacji poprawią sytuację rodzin, jeśli chodzi choćby o opiekę nad dziećmi, czy osób, które są wykluczone, choćby komunikacyjnie. Projektowane regulacje zastąpią obowiązujące przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, które okazały się zbyt mało elastyczne. Niektóre rozwiązania prawne dotyczące telepracy zostały jednak przyjęte do nowych kodeksowych przepisów o pracy zdalnej. Jeśli chodzi o zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości, zmierzają one do stworzenia podstaw dla pracodawców do prowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Będzie to jednak dopuszczane tylko wtedy, gdy przeprowadzenie takiej kontroli będzie niezbędne do ochrony określonych dóbr. Prace legislacyjne nad ustawą w tym zakresie zostały podjęte w związku z licznymi postulatami ze strony pracodawców, których pracownicy wykonywali czynności zawodowe, będąc pod wpływem substancji czy środków negatywnie wpływających na ich sprawność psychofizyczną. W tych przypadkach pracodawcy nie mieli możliwości przeprowadzenia samodzielnej weryfikacji takiego stanu, stąd też te zmiany, które proponujemy. Dzisiaj te kwestie były i są uregulowane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tak że te zmiany, które wprowadzimy do Kodeksu pracy, również te kwestie uregulują. Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, które są zawarte w tym projekcie, kilka z nich bardziej szczegółowo omówię. Jeśli chodzi o pracę zdalną, wprowadziliśmy definicję pracy zdalnej. Pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę, zatem będzie przewidywała to wprost umowa o pracę, albo już w trakcie zatrudnienia w formie zmiany warunków umowy o pracę, co do której nie będzie wymagana forma pisemna. Umożliwia się polecenie pracownikowi pracy zdalnej przez pracodawcę w szczególnych przypadkach, np. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, przy zastrzeżeniu dotyczącym złożenia przez pracownika bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie.

Wtedy regulamin będzie ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Umożliwia się wykonywanie pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo nie ma regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej.

Wprowadza się także możliwość przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa, chronienia informacji oraz zasad postępowania w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień.

Ważną zmianą jest wprowadzenie okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Z uwagi na jej szczególny charakter nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej, np. obowiązek zapewnienia materiałów i narzędzi pracy. Projekt, tak jak wspomniałem, przewiduje również rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście będziemy się posiłkować działem dziesiątym Kodeksu pracy, z wyłączeniem m.in. obowiązku organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami, zasadami BHP, obowiązku dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego czy obowiązku dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w formie zdalnej. Z uwagi na specyfikę i charakter zadań realizowanych przez funkcjonariuszy nieuzasadnione byłoby wprowadzenie w ustawach pragmatycznych służb całości rozwiązań związanych z pracą zdalną, które są zaproponowane w Kodeksie pracy.

Określenie przesłanek do wprowadzenia przez pracodawcę takich kontroli, którymi będą ochrona życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrona mienia, a także określenie zasad, na jakich pracodawca będzie te kontrole przeprowadzał. Nałożenie na pracodawcę obowiązku niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy w jego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu wskazująca na stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu. Nałożenie na pracodawcę obowiązku niedopuszczenia pracownika do pracy również w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał ww. środki w czasie pracy. Uregulowanie procedury przeprowadzania przez Policję badania w celu ustalenia obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Wprowadzenie możliwości odpowiedniego zastosowania przedstawionych rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy cywilnoprawnej, oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, jeżeli współpracują z tymi podmiotami. Uzupełnienie katalogu przesłanek uzasadniających pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej w przypadku stawienia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywania takiego środka w czasie pracy. Te rozwiązania zawarte w Kodeksie pracy będą miały też zastosowanie do przedsiębiorców niebędących pracodawcami organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą. Ze względu na specyfikę stosunku służbowego w projekcie ustawy zaproponowano również odrębne regulacje w zakresie badania na zawartość alkoholu lub na obecność innego, podobnie działającego środka w organizmach funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W zakresie pracy zdalnej oznacza to, że projektowane przepisy zastąpią w dniu wejścia w życie ustawy obowiązujące przepisy specustawy COVID-owej. W związku z tym pracodawca, ze względu m.in. na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będzie mógł wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na podstawie Kodeksu pracy.

W związku z tym zwracam się do Wysokiej Izby o dalsze procedowanie nad ustawą, o skierowanie jej do komisji kodyfikacyjnej i o szybkie procedowanie nad nią. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwsza pani poseł Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Tak jak pan minister mówił, ten projekt jest rozwiązaniem dotyczącym dwóch tematów, ma osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, ma on umożliwić pracodawcom, oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Pan minister, przedstawiając nam projekt, użył kilka razy słowa ˝kompromis˝, powiedział, że ten projekt był konsultowany z różnymi środowiskami. Chyba właśnie słowo ˝kompromis˝ jest bardzo ważne w zakresie dwóch regulacji.

Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję. Panie pośle, ja bardzo proszę. Panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Natomiast jeżeli chodzi o regulacje dotyczące pracy zdalnej, to tak jak powiedziałam, ta praca się sprawdziła i wydaje się, że potrzebne jest stałe uregulowanie jej w przepisach prawa.

Jeżeli chodzi o badanie na obecność alkoholu czy innych środków, ten kompromis jest potrzebny z tego powodu, żeby w przypadkach, kiedy jest to konieczne, pracodawca miał takie instrumenty i mógł badać przy wszelkich ograniczeniach dotyczących ochrony wolności, dotyczących ochrony danych.

Drugi kompromis to właśnie praca zdalna.

Lewiatan jest to organizacja, która skupia pracodawców, więc te stanowiska są przedstawione.

To rozwiązanie jest potrzebne i kierunki, które w tym projekcie są przedstawione, są przez nas, przez Prawo i Sprawiedliwość, popierane. Liczymy na to, że uda się ten projekt szybko przeprocedować i te przepisy z korzyścią i dla pracodawców, i dla pracowników szybko wejdą w życie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który jest zawarty w druku sejmowym nr 2335. To oczywiste, bowiem rzeczywistość zmienia się błyskawicznie. Pod wpływem gospodarczego przymusu, ale także pod wpływem sytuacji geopolitycznej stoimy przed koniecznością zwiększania wielostronności i szybkości rozwiązań, dostosowując rynek pracy do bieżących wyzwań. Zaproponowane w projekcie z druku nr 2335 zmiany regulują przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników, tj. wprowadzają możliwość monitorowania trzeźwości pracowników. Nowelizacja Kodeksu pracy jest oczekiwana zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, w szczególności ze względu na konieczność uregulowania w Kodeksie pracy zasad wykonywania pracy zdalnej. Projekt obejmuje rozszerzenie Kodeksu pracy o rozdział IIc, który można zatytułować: Praca zdalna. Jego przepisy umożliwią pracownikom całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu, które wskażą, a także każdorazowo ustalą z pracodawcą. Porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej będzie można uzgodnić zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również przepisy dotyczące porozumienia się pracodawcy z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników w kwestii zasad wykonywania pracy zdalnej. Przyjęty regulamin powinien obejmować m.in. sposoby kontrolowania wykonywania pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę informacji. Propozycja nowelizacji uwzględnia również obowiązki, które będą leżały po stronie pracodawcy, czyli m.in. zapewnienie narzędzi i materiałów do pracy, a także instalację, serwis, konserwację sprzętu, pokrycie kosztów energii i usługi telekomunikacyjnej w zakresie potrzebnym do pracowania na odległość. Wysoka Izbo! W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Projektowana ustawa uwzględnia postulaty pracodawców i wprowadza taką możliwość w przypadkach, w których jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Taki sposób ma zagwarantować przeprowadzenie badania z jak najmniejszą ingerencją w dobra osobiste pracownika. Projekt zakłada, że regulacje dotyczące kontroli pracowników znajdą się w odpowiednich źródłach zakładowego prawa pracy, czyli w regulaminach pracy, zakładowych układach zbiorowych pracy, w stosownych obwieszczeniach pracodawcy. Wysoka Izbo! Po zapoznaniu się z projektem pojawia się jednak wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Doprecyzowania wymaga artykuł, który określa wyłączenia pracy zdalnej. Jak w praktyce w odniesieniu do wykonywania poszczególnych zawodów mamy rozumieć pojęcia: uciążliwe zapachy czy intensywne brudzenie? Pojawiają się sygnały, że projektowane przepisy mogą utrudnić pracodawcom prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Do zagadnień wymagających doprecyzowania należą także zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Należałoby także rozważyć zwiększenie wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej. Ponadto okres wejścia w życie ustawy jest zbyt krótki na tak daleko idące zmiany. Sprawą kluczową jest wydłużenie vacatio legis, myślę, że co najmniej do 3 miesięcy. Klub Koalicji Obywatelskiej, w imieniu którego występuję, wnosi o skierowanie projektu do dalszych prac w komisji kodyfikacyjnej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze! W imieniu klubu Lewicy pozwolę sobie przedstawić klubowe stanowisko. Sama ustawa powinna i ma dostosowywać polskie przepisy do dwóch dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie przewidywanych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Projekt ustawy przewiduje, by nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. To stanowczo za mało. Chyba że byłby przepis przejściowy, zgodnie z którym pracodawcy stosujący pracę zdalną na podstawie polecenia będą mieli zdecydowanie dłuższy czas na wdrożenie nowych zasad.

Pracodawcy, związki zawodowe i pracownicy dopiero teraz mogą zapoznać się z ostateczną jego wersją. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość wprowadzenia prewencyjnych kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie oraz wprowadzenia regulacji pracy zdalnej jako rozwiązania stałego. Poprzednia wersja projektu przewidywała, że nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 3 miesięcy od odwołania stanu epidemii, niezależnie od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Już wtedy pracodawcy apelowali o więcej czasu na przygotowanie się do zmian. Tymczasem najnowszy projekt nowelizacji przewiduje tylko 2 tygodnie na wdrożenie tych zmian w zakładach pracy. To stanowczo za mało zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, i związków zawodowych, które mogłyby uzgadniać wszelkie regulacje. Brak kompleksowych przepisów przejściowych, zwłaszcza w zakresie pracy zdalnej, zaproponowane wejście w życie nowych przepisów już po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw będzie dużym utrudnieniem, a wręcz będzie niemożliwe do wdrożenia w tak krótkim czasie. Jednocześnie w tym samym terminie uchylone zostaną COVID-owe przepisy umożliwiające pracodawcom jednostronne kierowanie pracowników do pracy zdalnej. Jedyną podstawą pracy zdalnej będzie zatem znowelizowany Kodeks pracy. Dla wielu pracodawców ten termin jest niemożliwy do wdrożenia. Wprowadzenie pracy zdalnej według nowej definicji będzie wymagało podjęcia przez pracodawców szeregu działań, w tym m.in. ustalenia zasad pracy zdalnej, przygotowania regulaminu pracy zdalnej, zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielami. W takim przypadku przedsiębiorstwa, które nie posiadają takich przedstawicieli albo zostali oni wybrani jedynie do wykonania określonych czynności, będą musiały najpierw takich przedstawicieli wyłonić w wyborach przeprowadzonych wśród załogi. Z reguły dzieje się tak w samorządach, a to wymaga czasu, opracowania nowych zasad BHP w związku ze zdalną pracą, przeglądu wewnętrznych regulacji związanych z ochroną danych osobowych i poufnością informacji oraz wprowadzenia ewentualnych zmian uwzględniających charakter nowej pracy zdalnej.

Można się spodziewać, że w większości firm i samorządów początkowy okres stosowania nowych przepisów będzie fikcją. Na ten moment żaden pracodawca nie wszedł w dialog z organizacjami związkowymi czy przedstawicielami pracowników, ponieważ patrząc zdroworozsądkowo, czekamy na ostateczny kształt regulacji. Jednocześnie przypominam, że kością niezgody w Radzie Dialogu Społecznego był właśnie zwrot kosztów pracy zdalnej, a brak ustawowych zasad jego ustalania sprawia, że będzie to kwestia ocenna i niejednokrotnie budząca duże wątpliwości. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Ministrze! Właściwym rozwiązaniem byłoby zatem odpowiednio długie vacatio legis powiązane z końcem stanu zagrożenia epidemicznego i upływem kolejnych 3 miesięcy. Ustawa mogłaby zatem wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ustania stanu zagrożenia epidemicznego. Do tego okresu pracodawcy mogliby nadal korzystać z COVID-owych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej. Nic nie uległoby tutaj zmianie wobec stanu obecnego. Mieliby wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian. Jeśli natomiast stan zagrożenia zmieniłby się w stan epidemii, to nadal obowiązywałyby obecne przepisy i do wejścia nowych rozwiązań musieliby znowu poczekać. Skoro bowiem rząd przez 2 lata nie uznał za właściwe uregulowanie pracy zdalnej w ramach Kodeksu pracy, to pracodawcy mogą jeszcze poczekać kilka miesięcy. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów mam przyjemność przedstawić państwu stanowisko mojego klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z druku nr 2335. Ten projekt - jak już było podkreślane - do Sejmu wpłynął 7 czerwca tego roku, a 8 czerwca został skierowany do pierwszego czytania. Projekt dotyczy stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr prewencyjnych, kontroli pracowników na obecność w ich organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Projekt ma też na stałe w Kodeksie pracy uregulować pracę zdalną na czas po pandemii. Prace nad tymi nowymi przepisami trwały od 2020 r., a wersji projektu było kilka. Pandemia pokazała, że praca zdalna jest potrzebna, toteż projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw tę pracę zdalną w części reguluje, bowiem jasno określa definicję pracy zdalnej, tryb uzgadniania pracy zdalnej, określa jej zasady, jasno mówi o prawie pracodawcy do kontroli pracy zdalnej w godzinach pracy pracowników. Jednak tutaj pracodawcy mają wiele zastrzeżeń i mam nadzieję, że zostaną one wzięte pod uwagę na dalszym etapie prac nad tym projektem. Dobrym rozwiązaniem zawartym w tym projekcie jest świadczenie pracy zdalnej jako wsparcie dla rodziców. Dzięki temu pracowniczka w ciąży czy rodzice wychowujący dziecko do 4 lat lub dziecko niepełnosprawne oraz pracownik - rodzic dziecka posiadającego odpowiednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będzie mógł wystąpić do pracodawcy o świadczenie pracy zdalnej. To są dobre rozwiązania zawarte w tym projekcie.

Często pracodawcy zgłaszają, że jest ono zdecydowanie za krótkie, że trudno będzie zapisy tych zmian wprowadzić w życie, jeżeli będzie ono trwało 2 tygodnie. Klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie za skierowaniem tego projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych. Bardzo proszę, panie pośle. Szczęść Boże ludziom pracy różnorakiej, a kto nie pracuje, niech też nie je! Gdy wziąłem ten projekt do ręki - on jest z uzasadnieniem z kategorii tych obszerniejszych - na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że chodzi o to, że chcecie ustawowo zastrzec, żeby ludzie nie pili w pracy zdalnej. Tam wyliczacie policjantów, strażaków, bezpieczniaków. Inna rzecz, czy w praktyce to się da wyegzekwować, ale wymyśliliście narzędzia egzekwowania. Kiedy jednak wczytałem się głębiej w ten projekt, uświadomiłem sobie, że to jest pandemia+, 2.0, turbo. Znaleźliśmy się w stanie głębokiej pandemii i parafrazując klasyka, zaczynamy się w tym stanie coraz lepiej urządzać.

Sterroryzowaliście naród i przetresowaliście nieźle i teraz oferujecie szeroki wachlarz rozmaitych udogodnień. To z pozoru brzmi całkiem fajnie. Mam problem, uzgodnię z pracodawcą, nie przyjdę do roboty, będę pracować przy komputerze na stołku w kuchni, ale w normalnym życiu, dopóki nie wkroczyliście na scenę dziejową, takie rzeczy załatwiane były jak człowiek z człowiekiem, w normalnych relacjach międzyludzkich. Wy doprowadziliście te relacje do stanu takiej abnormalności, że trzeba to regulować, i teraz dla niektórych to będzie dobra oferta i nie zauważą, że następuje transakcja.

Regulujecie - uświadommy to sobie - procedury, które umożliwią wkraczanie z alkomatem czy z rozmaitymi innymi tam urządzeniami, pobieranie próbek płynów ustrojowych do analizy, do ekspertyzy, czy przypadkiem funkcjonariusz, który się umówił z przełożonym, że zostanie w domu i będzie tam, prawda, sobie googlał w robocie, to oczywiście w ramach obowiązków służbowych, czy nie jest nawalony. Nie popieram oczywiście stanów nietrzeźwości i odmiennych stanów świadomości w jakiejkolwiek pracy, zwłaszcza tak odpowiedzialnej jak służby mundurowe - jawne, tajne, ale (Dzwonek) sprzeciwiam się instytucjonalizowaniu tej już nie furtki, ale całej bramy, którą władza ludowa pod pretekstem walki z pandemią i ułatwiania ludziom życia wkracza w naszą prywatność. Dlatego pójdę dalej, nie wnioskuję o przesłanie tego projektu do komisji tylko o wyrzucenia go do kosza. Wróćcie z czymś ludzkim. Jeżeli uważacie, że trzeba regulować, no to nie wprawiajcie mnie w podejrzenie, że szykujecie sobie po prostu nowe rozwiązanie na czas nowej pandemii, którą zapowiedzieli już premier Morawiecki i prezydent Biden.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zmiany w Kodeksie pracy są wyczekiwane i to przedłożenie jest bardzo istotne, tym bardziej że nasze rodzime rozwiązania prawne w tym zakresie prawa dosyć mocno i coraz bardziej odstają od Europy. Pracę zdalną doceniliśmy w czasie pandemii. Naprawdę nie trzeba siedzieć w biurze, żeby być efektywnym. Ta prawda jest znana od dawna w korporacjach, niedawno stała się oczywista również dla pozostałych sektorów. To, co z samej zasady ma być elastyczne, źle znosi usztywnione gorsety. W przedłożeniu widzimy bardzo mocne sformalizowanie modelu pracy zdalnej - ot, chociażby konieczność każdorazowego uzgadniania miejsca pracy zdalnej albo np. pewne zastrzeżenia co do wymiaru tej pracy. Np. na tzw. incydentalną pracę zdalną wskazano 24 dni w ciągu roku. To jest bardzo mało. Przed pandemią standardem tzw. pracy domowej był 1 dzień w tygodniu, a to daje 52 dni rocznie. Może to spowodować, że ta słuszna zmiana zadziała w sposób cokolwiek ograniczony. To jest bardzo ważny postulat od wielu lat zgłaszany przez organizację pracodawców. Pracodawca musi ocenić niezbędność tej kontroli dla życia i zdrowia innych pracowników albo innych osób. Jak taką niezbędność udowodnić? Bardzo, bardzo trudno będzie pracodawcy podjąć takie ryzyko, zważywszy na to, że będzie musiał liczyć się z reakcją pracownika, niekoniecznie reakcją w miejscu pracy tu i teraz, czasem reakcją w jakimś horyzoncie sądowym. Jeżeli dajemy pracodawcom takie narzędzie, które ma służyć bezpieczeństwu wszystkich, to niech ono będzie sprawne i niech będzie wszechstronne w użyciu. Reasumując, bardzo się cieszę, że wreszcie pracujemy nad Kodeksem pracy, tym bardziej że przed nami mnóstwo zadań dotyczących tego dokumentu. W kolejce czekają, przypomnę tylko, dyrektywa Parlamentu Europejskiego o sygnalistach - byliśmy zobowiązani do jej przyjęcia z końcem ubiegłego roku - dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy, dyrektywa o równowadze pomiędzy pracą a życiem poza pracą, ordynarnie nazywanej work-life balance. Mam nadzieję, że doczekamy się jak najszybciej wszystkich tych dokumentów tutaj, na sali plenarnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwsza pani poseł Wanda Nowicka, Lewica. Nie ma pani poseł. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rozmawiamy dzisiaj o projekcie ustawy z druku nr 2335 dotyczącym Kodeksu pracy. Mam bardzo krótkie pytanie i chciałbym, żeby pan był uprzejmy mi odpowiedzieć na nie pisemnie. Z jakimi związkami zawodowymi ten konkretny druk był konsultowany? Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mamy tymi zapisami załatwiony częściowo i uregulowany problem alkoholu i osób pod jego wpływem, które chcą przystąpić do wykonywania czynności zawodowych. Natomiast chciałem zapytać, co z całą gamą powszechnie stosowanych innych środków odurzających. Czy pracodawca powinien mieć możliwość pełnej i dokładnej kontroli osób, którym powierza się życie innych ludzi lub majątek często wart miliony złotych? Bardzo bym prosił pana ministra o odpowiedź na pytanie, jaka jest wizja resortu w tej sprawie. Pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Koalicja Obywatelska. Chciałam zadać dwa pytania. Po pierwsze: Na czym mają polegać warunki techniczne i lokalowe dla pracy zdalnej i kto je zapewnia? Czy chodzi o zakup odpowiedniego biurka, krzesła dla pracownika, czy może innych odpowiednich rzeczy, takich jak podnóżek albo podstawka pod monitor? W całej ustawie pojawia się pojęcie formy papierowej. Czym ona jest? Jak można papierowo złożyć oświadczenie? Mowa o takiej formie np. w odniesieniu do zapoznania się przez pracownika z procedurami ochrony danych osobowych albo szkolenia BHP. Zdaje się, że w polskim porządku prawnym mamy formę pisemną i formy równoważne, czyli kwalifikowany podpis elektroniczny czy formę dokumentową. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja.

Na szczęście dlatego, że do tej pory nie zdążyliście napisać tych wszystkich regulacji. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby to zepsuć.

Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po pierwsze, spójność obydwu tych części.

Rozumiem, że ono będzie dotyczyć różnych zagrożeń, które występują w mieszkaniu, a znajomość mieszkania przy pracy zdalnej, jeżeli ktoś pracuje z własnego domu.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050.

Pani Marszałek! Mam dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczy zmian, które wprowadzają państwo w umowach na okres próbny. Bardzo mocno formalizują państwo te umowy na okres próbny, w szczególności uzależniają państwo czas trwania takiej umowy na okres próbny od zamiaru pracodawcy zawarcia kolejnej umowy na czas określony. Troszkę tego nie rozumiem. Okres próbny to jest okres próbny i on ma obu stronom w stosunku pracy pokazać, czy nadają się nawzajem do tego, aby taki stosunek kontynuować. Drugie pytanie dotyczy vacatio legis. Proszę pamiętać, co wszystkie działy kadr, co wszystkie działy zarządzania zasobami ludzkimi przechodziły podczas pandemii, kiedy przepisy zmieniały się jak w kalejdoskopie i wszyscy kadrowcy, wszyscy płacowcy musieli odpowiadać na te bez ustanku zmieniające się przepisy.

To było ostatnie pytanie.

Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję wszystkim klubom za poparcie rozwiązań dotyczących pracy zdalnej, jak również umożliwienie pracodawcom badania trzeźwości. Jeśli chodzi o pytania, to jeszcze raz przypomnę generalną zasadę tych zmian, które wprowadzamy, dotyczącą pracy zdalnej. Ona ma się tak naprawdę opierać na porozumieniu między pracownikami i pracodawcą.

W tym przypadku pracodawca nie będzie mógł odmówić, a jeżeli odmówi, to będzie musiał uzasadnić, jaka jest przyczyna odmowy takiej pracy.

Z drugiej strony pracodawca w sytuacjach kryzysowych, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, przy COVID-zie, będzie mógł taką pracę powierzyć pracownikowi. Były też dyskusje dotyczące określenia kosztów. Ta dyskusja przewijała się również w pracach zespołu Rady Dialogu Społecznego.

Tak jak już powiedziałem, jest to kompromis między stroną pracodawców a związkami zawodowymi.

Pan poseł Gramatyka pytał o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz nie jest w tej ustawie. To jest następna ustawa dotycząca zmian w Kodeksie pracy, ale ona jest jeszcze w konsultacjach, tak że w tej ustawie, jeśli chodzi o okresy próbne, nie ma tych zapisów.

Bardzo dużo wątków dotyczących terminu wejścia w życie ustawy. Bo w pierwotnym projekcie było po 3 miesiącach zakończenia stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego. Tutaj na ten moment po wprowadzeniu krótkiego vacatio legis dalej działają przepisy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, czyli w dalszym ciągu pracodawca będzie mógł korzystać z rozwiązań, które są w tej chwili, ale skracając ten termin do 14 dni, ułatwiamy w tym przypadku osobom, o których mówiłem, czyli matkom wychowującym dzieci do 4 roku życia czy kobietom w ciąży, czy rodzicom, którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, że już będą mogli w krótkim okresie wystąpić do pracodawcy o powierzenie takiej pracy.

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy na następnym posiedzeniu Sejmu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696) Proszę pana posła Grzegorza Wojciechowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu.

Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Przedmiotem tej petycji było właśnie żądanie podjęcia inicjatywy w zakresie zmiany obowiązujących przepisów dotyczących egzekucji sądowej i administracyjnej. Zaraz to uzasadnię. A celem jest zwiększenie skuteczności dochodzenia. Projekt tego aktu prawnego został zamieszczony również w samym tekście petycji, z tym że efekt tej ustawy jest to już efekt pracy komisji i w szczegółach ten projekt nieco się różni od projektu, który został wniesiony, jednak merytorycznie jest to ten sam projekt. Do tego projektu w zasadzie do petycji raczej została sporządzona opinia Biura Analiz Sejmowych. Z tej opinii wynika również potrzeba zmian przepisów w zakresie egzekucji. Komisja petycji również wystosowała dezyderat do ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości w odpowiedzi na dezyderat wskazał także, że zmiana tych przepisów jest uzasadniona, i jednocześnie wskazał, że w najbliższym czasie nie są przewidywane zmiany. W związku z powyższym komisja petycji uznała, że złoży stosowny projekt ustawy. Projekt ustawy składa się w sumie z sześciu artykułów. Ideą tego projektu jest zwiększenie skuteczności egzekucji, zarówno egzekucji administracyjnej, jak też różnych innych egzekucji, bo tam są inne przepisy dotyczące egzekucji alimentów, a więc inne niż właśnie egzekucja alimentów.

Autor tej petycji złożył postulat, aby nie chronić w pełni wynagrodzenia minimalnego, lecz jedynie jego 85%. Wskazał przy okazji, że to minimalne wynagrodzenie jest coraz bardziej odległe od pewnych podstawowych minimalnych kosztów utrzymania czy też minimum socjalnego, czy też jeśliby w jakiś inny sposób nazwać tę minimalną wartość, która jest potrzebna do utrzymania się dłużnika.

Obecnie jest to 60% wynagrodzenia, natomiast autor proponuje zmianę do 50% wynagrodzenia.

Art. 5 wskazuje, że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w tych czterech artykułach w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i jest propozycja, aby vacatio legis w tym wypadku wynosiło 6 miesięcy. Również wpłynęły opinie dotyczące już tego konkretnego druku nr 1696 - od Konfederacji Lewiatan, od Narodowego Banku Polskiego, od NSZZ ˝Solidarność˝, od OPZZ, od Sądu Najwyższego. Wpłynęło również stanowisko rządu, może zacytuję fragment: Uwzględniając powyższe, Rada Ministrów pozytywnie ocenia komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, druk nr 1696, z tym jednak zastrzeżeniem, że obecny kształt wymaga dalszego dopracowania w taki sposób, aby uwzględniał pewne zastrzeżenia, które zostały wskazane przez ministerstwo. To tyle z mojej strony, pani marszałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, druk nr 1696. Projekt dotyczy zwiększenia skuteczności egzekucji sądowych i administracyjnych innych niż alimentacyjne oraz wprowadzenia zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunku bankowego i z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Proponowane zmiany mają za zadanie zwiększyć skuteczność powyższych egzekucji i stanowią uzupełnienie dotychczas podjętych działań legislacyjnych zmierzających do poprawy ich efektywności. Niska skuteczność egzekucji sądowych i administracyjnych jest spowodowana m.in. wzrostem wynagrodzenia minimalnego w ostatnich latach. Wysokość kwot wolnych od egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego powiązana z wynagrodzeniem minimalnym sprawia, że stale rośnie liczba dłużników, których nie można poddać skutecznej procedurze egzekucyjnej. Dochodzi do patologicznych przypadków zatrudnienia z wynagrodzeniem minimalnym, które jest wolne od potrąceń, oraz otrzymywania pozostałej części wynagrodzenia w sposób nierejestrowany. W wyniku tego rośnie liczba wierzycieli, którzy nie mają szans na odzyskanie utraconych pieniędzy. Tym samym obowiązujące obecnie przepisy tworzą podstawę prawną do ochrony wynagrodzenia za pracę, która w praktyce nie odpowiada współczesnym realiom gospodarczym oraz narusza zasadę równowagi pomiędzy prawami podmiotów dochodzących swych należności a zachowaniem praw dłużników. Przepisy w niezamierzony sposób faworyzują grono dłużników, czyniąc ich uprzywilejowanymi. Zaproponowane w projekcie rozwiązania zmierzają do ograniczenia skali niesprawiedliwości wobec równego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie zaś pozwalają dłużnikom na zachowanie środków niezbędnych do życia. Jednakże nowe przepisy powinny uwzględniać także sytuację życiową dłużników, stąd w toku dalszych prac legislacyjnych należy wyeliminować brak zróżnicowania między np. osobą samodzielnie utrzymującą z minimalnego wynagrodzenia za pracę kilkuosobową rodzinę a osobą z minimalnymi zarobkami pozostającą na utrzymaniu rodziców itp. Ponadto projekt zakłada, że kwota wolna od egzekucji z wynagrodzenia za pracę zostanie obniżona o 15%, zaś w odniesieniu do egzekucji z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego na rzecz członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej kwota wolna od zajęcia zostanie obniżona o ponad 33%. Zatem warto przedyskutować kwestię ujednolicenia tych dysproporcji. Reasumując, rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie ustawy pozwolą na ograniczenie możliwości unikania odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Pozytywnie wpłyną na sytuację prawną wierzycieli będących zarówno przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi. Biorąc powyższe pod uwagę, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość deklaruję poparcie dla niniejszego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Zwiefka, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt, nad którym dzisiaj dyskutujemy, przygotowany przez komisję petycji, jest szalenie istotny dla kilku grup. Bardzo istotny jest dla grupy dłużników, ponieważ ma wpłynąć na zmniejszenie kwoty, która dzisiaj jest chroniona przed egzekucją sądową czy też administracyjną. Z drugiej strony ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności egzekucji, by poprawić sytuację wierzycieli. To ma również ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu ostatnich lat skuteczność egzekucji systematycznie spada. Jeśli przyjmiemy, że w roku 2020 całość środków, które zostały odzyskane przez wierzycieli w drodze egzekucji, wynosiła ponad 9 mld zł, to w roku 2021 r. była to kwota o prawie miliard złotych niższa. To pokazuje, że wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także różnego rodzaju zabiegi polegające na pobieraniu wynagrodzenia w sposób niekoniecznie ujawniony, czyli tzw. płacenie pod stołem, powoduje trudności w odzyskaniu należności przez wierzycieli. Ma to oczywiście wpływ także na funkcjonowanie gospodarki, szczególnie w obrocie mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Niestety nie znalazłem nigdzie danych mówiących o procentowym udziale w odzyskiwaniu tych środków, kwot, które dotyczą należności dla Skarbu Państwa, kwot, które wiążą się z odzyskiwaniem należności dla przedsiębiorców czy też dla indywidualnych osób, a warto by poznać także te zależności. A zatem pracując nad przedłożonym przez komisję petycji projektem, powinniśmy zwrócić uwagę na balans pomiędzy interesem dłużnika a interesem wierzyciela, balans, który został w sposób dosyć wyraźny zaburzony na korzyść dłużnika. W o wiele trudniejszej, gorszej sytuacji znajdują się dzisiaj wierzyciele. Z drugiej strony, kiedy uświadamiam sobie, że ten projekt wpłynął do Wysokiej Izby końcem poprzedniej kadencji, a procedujemy nad nim dopiero dzisiaj, to ta sytuacja powoduje, że również inaczej patrzymy na kwestię minimalnego wynagrodzenia oraz pozycję dłużników. Wzrost inflacji, trudna sytuacja gospodarcza, wysokie ceny, mówiąc krótko: drożyzna, powodują, że bardzo często dłużnicy, ci uczciwi dłużnicy, mają istotne problemy z oddawaniem długu. Postawienie ich teraz w jeszcze trudniejszej sytuacji może spowodować rzeczywiście bardzo poważne problemy w ich życiu osobistym czy rodzinnym, bowiem często mają na utrzymaniu także inne osoby. To też musimy wziąć podczas naszych rozważań pod uwagę. Wspomniana została kwestia różnych procentowo ujęć, jeśli chodzi o zmniejszanie kwoty, która jest chroniona w przypadku wynagrodzenia za pracę, w przypadku wynagrodzenia za pracę więźniów czy w przypadku zajęć finansowych dotyczących kont bankowych bądź kont indywidualnych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych. Też musimy zastanowić się, czy ta różnica musi wynosić aż tyle, czy w ogóle powinna być jakakolwiek różnica, i w którą stronę to zrównanie powinno zdążać, czy w stronę tego mniejszego, 15-procentowego ograniczania, czy też tego większego, ponad 30-procentowego. Wiąże się to z pytaniami, które się pojawiają, a mają wpływ zarówno na grupę dłużników, jak i na grupę wierzycieli, ale także tych pracowników, którzy zajmują się ściąganiem należności. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska proszę o przesłanie tego projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Anna Maria Żukowska, Lewica. Wysoka Izbo! Pan poseł z PiS już przedstawił, właściwie przeczytał, całe uzasadnienie tego projektu, dlatego nie ma sensu do niego wracać i je powtarzać, bo właściwie słyszeliśmy je dwa razy, również od pana posła wnioskodawcy. Lewica zawsze skupia się na sytuacji osób najsłabiej uposażonych. I jeżeli ktoś zarabia pensję minimalną, to samo to sformułowanie, że jest to płaca minimalna, oznacza, że naprawdę nie jest to wysokie wynagrodzenie, nie są to duże zarobki, i to w czasie, kiedy mamy taką sytuację gospodarczą i raty kredytów rosną z miesiąca na miesiąc nieraz o kilkaset złotych.

Myślę, że musimy o tym porozmawiać. Myślę, że ten projekt powinien być lepszy i powinien przewidywać takie sytuacje, które muszą przeciwstawiać się wpadaniu Polek i Polaków w pętlę zadłużenia, która niestety często kończyć się może tylko na bezdomności. Tego byśmy chcieli zdecydowanie uniknąć. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Maliszewski, Koalicja Polska. Nie ma pana posła. Pan poseł Krzysztof Tuduj, Konfederacja. Wysoka Izbo! Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję złożoną przez osobę fizyczną. Celem tej ustawy jest zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej poprzez zmianę czterech ustaw: Kodeksu pracy, Kodeksu karnego wykonawczego,

Regulacja będzie miała pozytywny wpływ właśnie na wierzycieli, zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Konkretnie przedłożenie zawiera propozycje zmiany przepisów umożliwiających prowadzenie egzekucji należności innych niż alimentacyjne na wyższym poziomie w zakresie kwot wolnych od potrąceń, w ramach egzekucji z wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia skazanego lub osadzonego, oraz z rachunku bankowego i rachunku prowadzonego w SKOK. W przypadku wynagrodzenia za pracę kwotę wolną od egzekucji stanowi obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych i rachunkach w SKOK były wolne od potrąceń do wysokości 50%, a obecnie jest to 75%. Jako były specjalista do spraw windykacji uważam te rozwiązania co do zasady za słuszne. Ludzie powinni brać odpowiedzialność za zobowiązania, jakie zaciągają, spłacać swoje długi, oddawać pieniądze, jakie pożyczyli.

Przy tak galopującej inflacji, wzroście cen projekt będzie uderzał w osoby, które starały się odpowiedzialnie prowadzić własne finanse, ale takiego wzrostu rat kredytu nie były sobie w stanie wyobrazić. Reasumując, to przedłożenie, które rząd na pewno poprze, najbardziej pomoże bankom. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pan poseł Tomasz Zimoch, który przedstawi stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050. Panie Ministrze! Chciałoby się zakrzyknąć: W obywatelach moc! Bo oto 30 lipca 2019 r. pan Kamil Łagocki złożył w Sejmie petycję w interesie publicznym. Uważał, że w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej istnieje potrzeba zmiany w Kodeksie pracy, Kodeksie karnym wykonawczym, Prawie bankowym oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Po raz kolejny warto podkreślić obywatelską siłę petycji. Sejmowe ukłony dla autora. Brawo, panie Kamilu! Zresztą nie pierwszy raz w tej kadencji Sejm przyjmie ustawę właśnie za sprawą petycji pana Kamila Łagockiego. W petycji zwrócił uwagę, że proponowany projekt jest istotnym uzupełnieniem podjętych dotychczas działań prawodawczych oraz całościowym rozwiązaniem problemów, które dostrzeżono także w orzecznictwie sądowym. M.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wskazano, iż skuteczna egzekucja prawa jest jednym z najważniejszych zadań demokratycznego państwa prawa. W opinii wnioskodawcy jedynie wskazanie nowych kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego na rzecz członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może w pełni zrealizować postulaty ustawodawcy. Projektowana ustawa bezspornie przyczyni się do zdecydowanej poprawy skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej. Autor petycji podkreśla, że statystyki dotyczące skuteczności egzekucji są niezadowalające.

Na problem małej efektywności egzekucji administracyjnej wskazywała również Rada Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022. Proponowana ustawa zdaniem pana Kamila Łagodzkiego zwiększy prestiż państwa oraz pozytywnie wpłynie na gospodarkę oraz dochody jednostek sektora finansów publicznych. Należy przy tym podkreślić, że celów zakładanych w tym projekcie ustawy nie można osiągnąć w inny sposób, zaś podejmowane dotychczas działania legislacyjne nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

Właśnie wtedy zrodził się pomysł tej konkretnej petycji. Raz jeszcze ukłony dla autora. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, w obywatelach moc. Bardzo dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do zadawania pytań. Jeżeli nie, to informuję, że zapisało się pięcioro państwa posłów, a właściwie pięciu panów posłów. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Rafał Adamczyk. Nieobecny. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozumiem, że pewien obywatel chce w możliwie szybki sposób odzyskać swoje pieniądze, i trudno mieć o to do niego pretensje. Czy jednak możemy skazywać miliony najuboższych Polaków na bezdomność, skrajne ubóstwo, czy nawet śmierć w wyniku np. zaniechania zażywania leków? Nie można odbierać ludziom środków, które zostały wyliczone jako minimum niezbędne do ich funkcjonowania. Czy można to robić zwłaszcza w okresie katastrofalnej inflacji oraz horroru, który polskie rodziny przeżywają w związku z niekontrolowaną w żaden sposób podwyżką cen żywności, ogrzewania oraz energii elektrycznej?

Długi na pewno trzeba spłacać, ale nie za cenę życia dłużnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Grzegorz Lorek. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Nigdy nie ma dobrego czasu. Zawsze coś się dzieje w kraju, na świecie i ten czas nie jest najlepszy. Tu bardzo dobre zdanie powiedział chyba pan poseł Tadeusz: to balansowanie między dłużnikiem a wierzycielem. To jest bardzo trudne do osiągnięcia, ale myślę, że trzeba się nad tym zastanowić. Każdy z nas, tak mi się wydaje, zna jakieś rozbite małżeństwo. Przychodzą ze sprawami alimentów, które nie są ściągane lub egzekwowane. Powstają gigantyczne problemy, długi. Wtedy ten problem jeszcze bardziej narasta, ślad się urywa, co też potęguje skalę tego zjawiska. Balansowanie między dłużnikiem (Dzwonek) a wierzycielem - myślę, że trzeba nad tym pomyśleć i że projekt jest wart uwagi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Cała Polska zadłużona. Kto nie odbierał monitów, kto nie odbierał telefonu, a może domofonu, z komornikiem po drugiej stronie, niech pierwszy rzuci kamieniem.

Jesteśmy na najlepszej drodze. Pytanie o tę płacę minimalną czy w ogóle przy okazji. Bo co innego jest płaca minimalna w Szczecińskiem, a co innego w Przemyskiem.

Bardzo dziękuję. Listę posłów zapisanych do pytań zamyka pan poseł Tomasz Zimoch. Panie Marszałku!

Bardzo dziękuję panu posłowi. Zapraszam na mównicę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Michała Wosia. Wysoka Izbo!

Niewątpliwie projekt jest pożądany, wprowadza pożądane rozwiązanie w zakresie skutecznej egzekucji prawa do sądu.

Natomiast chciałbym się odnieść do pewnych spraw, które padły z mównicy i które niekoniecznie mają walor prawdziwości. Odnosząc się do lewicowej wrażliwości, proszę pamiętać, że czym innym jest minimum socjalne, a czym innym jest płaca minimalna. Minimum socjalne jest określane przez jeden z instytutów badawczych podległych ministrowi rodziny i polityki społecznej na ok. 1200-1300 zł w ostatnich badaniach. I biorąc pod uwagę te liczby bezwzględne, propozycja obniżenia kwoty wolnej od zajęcia z minimalnej na 85% minimalnego wymaga też spojrzenia na tę propozycję w walorze kwotowym. A mianowicie, biorąc pod uwagę minimalną netto, mamy do czynienia z ok. 2200-2300 zł, a jeszcze więcej, biorąc pod uwagę różne zmiany podatków, natomiast po wzroście płacy minimalnej do 3450, przy uwzględnieniu zmian podatkowych i przy uwzględnieniu ewentualnego wejścia w życie tego projektu, czyli 85% płacy minimalnej, ta kwota i tak będzie wyższa. I to jest coś istotnego, co należy wziąć pod uwagę.

Szanowni Państwo! A mianowicie pod rozwagę trzeba wziąć na pewno poziom obniżenia tego pułapu, bowiem w jednym przypadku mamy obniżenie ze 100% minimalnej do 85%, czyli o 15 punktów procentowych. W związku z tym wymagałoby wnioskodawcy.

Drugą propozycją opracowaną we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej jest propozycja uwzględnienia walorów domu tej osoby, czyli czy ma dzieci na utrzymaniu, czy to jest jednoosobowe gospodarstwo, bo to sprawia, że jest jednak pewna różnica. W związku z tym można by rozważyć, czy czasem o określony odsetek nie powinno się wprowadzić pewnego mechanizmu, w którym kwota wolna od zajęcia ulegałaby podwyższeniu np. o 5 punktów procentowych. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Czy pan poseł przedstawiciel wnioskodawców zamierza zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Również na posiedzeniu komisji petycji była dyskusja dotycząca tego, czy płaca minimalna jest dobrym wskaźnikiem dotyczącym sytuacji danego człowieka, czy jest on w stanie spłacać, czy nie jest w stanie spłacać swojego zobowiązania bez naruszenia podstawowych potrzeb utrzymania, potrzeb życiowych.

W związku z tym mamy dezyderat. Ministerstwo odpowiada: tak, istotnie, tak jest. Przy pierwszej zmianie to zrobimy.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zawarty w druku nr 1696, do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 57. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Na razie wygląda na to, że nikt nie zgłosił się do oświadczeń. Jednak są państwo. Pani poseł Wanda Nowicka.

Marszałku! Wysoka Izbo! Dobiega końca posiedzenie. Nie ma w tej Izbie ani w żadnej izdebce na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej miejsca, w którym można by pilnie reagować na rozmaite zagrożenia, które pojawiają się na horyzoncie. W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym podyktować do protokołu, szanowni państwo, że niepokoi mnie przybycie do Warszawy - po raz kolejny w tym sezonie - pana Davida Harrisa, szefa czegoś, co nazywa się Amerykańskim Komitetem Żydowskim - American Jewish Committee. Myślę, że pan Harris może być już powoli nazywany bywalcem.

Od lat jest on też szermierzem interesu żydowskiego, działając głównie z drugiej strony globusa, z tamtej strony. Rzecz w tym, że to są - jak wiemy z doświadczeń historycznych - sprawy bardzo poważne. Potrącenie tej struny często wywołuje wilka z lasu i.

Myślę, że sprawa jest ciekawa i rozwojowa. Więc tak to bywa, że kiedy pytamy o te sprawy, to mówią nam, że to jest kurtuazja, dyplomacja, że nie należy tych wrażliwych spraw w stosunkach polsko-żydowskich psuć jakimiś krytycznymi uwagami, przesadną podejrzliwością. Potem, jak przychodzi co do czego, to wyjeżdżający - np. na drugą stronę globusa - oficjele warszawscy, prezydent belwederski czy premier składają wręcz wizyty ad limina w siedzibach organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. A zatem, choć nie mamy do czynienia z głową żadnego państwa ani nawet główką, to jednak czasami zdaje się, że ogon merda psem i że są to sprawy być może najbardziej istotne dla przyszłości i dla majętności Polaków.

Oczywiście chodzi o tzw. roszczenia, uroszczenia, czyli prawem kaduka wymuszane cesje majątkowe. To po prostu żądanie pieniędzy.

I teraz rząd PiS-u reklamuje, że teraz już będzie bardzo asertywny. Ostatnia kwestia. Ostatnia kwestia, panie marszałku. Zadaję pytanie, które oczywiście pozostanie dziś wieczór retorycznym, czy nasadzenie pana Kościńskiego, wielki powrót Kościńskiego do rządu, akurat na tak wrażliwy odcinek jak zbrojeniówka, zakupy zbrojeniowe, które jak wiadomo, mogą być przykrywką dla dowolnych gabarytów transferów finansowych, czy nie ma czegoś wspólnego jedno z drugim, z trzecim. Akt 447, wojna na Ukrainie, wymuszenia żydowskie wobec Polaków, być może transmitowane na Ukrainę. Szanowni państwo, moim zdaniem roszczenia wracają. I naprawdę to już postscriptum, moje jaskółki doniosły, że w Waszyngtonie ambasador Magierowski zaangażował się - oczywiście w tajemnicy przed polską opinią publiczną, nie wiem, czy jawnie dla całego rządu - w negocjowanie spłaty urojonych roszczeń żydowskich pod szantażem trwającym lata i że zostały one jakoś tam wstępnie wylicytowane na określoną sumę w miliardach. Warto dopytać się, panie pośle, tych jaskółek w tej kwestii. Mówię, że warto tych jaskółek troszkę bardziej szczegółowo się dopytać, bo kwestia jest, jeżeli faktycznie prawdziwa, to niezwykle interesująca.

Panie Marszałku! Rzecz jasna, nie zaniedbuję okazji, ale myślę, że marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ma nieporównanie poważniejsze narzędzia dochodzenia przynajmniej odpowiedzi na dobrze postawione pytania w tej sprawie. Więc dobrze postawione pytanie brzmiałoby i może zadam je w trybie doniesienia publicznego: Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej negocjuje z Żydami wypłacenie - w gotówce lub w naturze, w postaci transferów jawnych czy ukrytych, pod przykrywką operacji pomocy zbrojnej Ukrainie -jakichkolwiek kwot? Proszę zredagować, panie marszałku, w sposób dowolny, sobie właściwy te pytania, ale myślę, że tak ono by brzmiało. Ale obecny jest pan poseł Grzegorz Lorek. Proszę o wygłoszenie oświadczenia. Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niektóre wydarzenia w historii Polski są przeceniane, jak twierdził profesor Ludwik Stomma. Jednak na pewno nie należą do tej kategorii wybory lub plebiscyt, który odbył się 4 czerwca 1989 r. Poprzedziła je długa droga. Ów czerwiec nie był zjawiskiem odosobnionym. W Polsce historia galopowała od lutego 1989 r., kiedy ówczesny rząd rozpoczął rozmowy z opozycją przy tzw. okrągłym stole. Zostawmy na boku kulisty tych wydarzeń. Dość powiedzieć, że trwające od kwietnia obrady zaowocowały powtórną rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ˝Solidarność˝, zmianą ordynacji wyborczej oraz przyspieszeniem wyborów do Sejmu i po raz pierwszy do Senatu. Niektórzy historycy nazywają owe wybory pierwszym plebiscytem, który miał pokazać prawdziwe zaufanie do ówczesnych komunistycznych władz. Wybory, choć koncesjonowane i nie do końca wolne, pokazały jednoznacznie, że PZPR straciło legitymację do sprawowania władzy. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa, Bełchatowa czy innych miast regionu różnie wspominają tamten czas. Jedni pamiętają plakaty z Lechem Wałęsą firmującym swoim wizerunkiem kandydatów Komitetu NSZZ ˝Solidarność˝, inni plakaty, ulotki PZPR (Dzwonek), a jeszcze inni rzeczy o którym mówiły: nie bierzcie udziału w tych wyborach. Wszyscy jednak mówią zgodnie, że największe wrażenie robił plakat z uzbrojonym kowbojem ze znaczkiem ˝Solidarność˝, Garym Cooperem. Przekaz był jasny: jedyny sprawiedliwy w tym mieście. Nieżyjący już Zbigniew Mroziński, działacz związkowy, a później poseł III Kadencji NSZZ ˝Solidarność˝, nie był początkowo entuzjastą okrągłego stołu, jednak przyłączył się do ruchu mając nadzieję na zmianę. Startująca i wybrana z Tomaszowa Mazowieckiego Teresa Zalewska była pełna obaw, czy da sobie radę w Sejmie. Wspominał on: brakowało wszystkiego, ale nie determinacji do zmian. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz o wygłoszenie oświadczenia pana posła Krzysztofa Janusza Kozika, jeżeli jest obecny na sali. Jest. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niedawno przeżywaliśmy dwie ważne rocznice. 18 czerwca 1792 r. miała miejsce bitwa pod Zieleńcami, stoczona pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki a wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez gen. Morkowa. Miała ona miejsce rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Polskie oddziały liczyły ponad 15 tys. żołnierzy, natomiast rosyjski korpus ekspedycyjny - 11 tys. żołnierzy. Bitwa pod Zieleńcami była pierwszą od prawie wieku wiktorią polskiego wojska, porównywaną w tamtym czasie w odsieczą wiedeńską z 1683 r. Poza przewagą liczebną Polaków właściwie wszystko przemawiało na korzyść Rosjan. Mimo to armia polska odniosła zwycięstwo nad armią carów i zmusiła Rosjan do wycofania się. Nie sposób nie dopatrzyć się analogii w kontekście obecnej agresji Rosji na Ukrainę i kontestowania bytu suwerennego państwa. Oczy całego świata od 24 lutego br. zwrócone są na Ukrainę i miejmy nadzieję, że wojna w obronie kraju okaże się zwycięska dla naszych sąsiadów. Warto dodać, że w dniu bitwy pod Zieleńcami książę Józef Poniatowski w pisanym do króla Stanisława Augusta raporcie zwrócił się o wprowadzenie nowego odznaczenia wojskowego. Miało być ono formą podziękowania za męstwo, ale i chodziło o podniesienie morale wśród żołnierzy.

Wśród pierwszych 15 udekorowanych najstarszym orderem wojskowym na świecie spośród tych, które są jeszcze obecnie nadawane, znaleźli się m.in. generałowie: książę Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko i Józef Zajączek. Jak dotąd orderem odznaczono ok. 26 tys. osób. Statut przewidywał pięć klas orderu: Krzyż Wielki z Gwiazdą, Krzyż Komandorski, Krzyż Kawalerski, Medal Złoty i Medal Srebrny. Na wzór Orderu Marii Teresy oznaczenie uzyskało kształt krzyża, na którym widniał rok 1792 oraz herby: Korony - Orzeł i Litwy - Pogoń. Order Wojskowy Virtuti Militari, który zachował pięć klas i kształt krzyża, został przywrócony dopiero w wolnej Polsce, a jego dewizą stały się słowa: Honor i Ojczyzna. Te wymowne słowa były wiążące dla żołnierzy, bowiem dzięki takim postawom i takiemu hartowi ducha, jak podczas bitwy pod Zieleńcami, udało się pokonać wroga. Cenna lekcja historii powinna być stale aktualna i przekazywana z pokolenia na pokolenie, ponieważ, jak mawiał Jan Paweł II, naród, który traci pamięć, traci również swoją tożsamość. Tym bardziej w kontekście agresywnego zachowania Rosji wobec suwerennych sąsiadów musimy pamiętać o tym, że tylko wspólne działanie dla dobra naszego kraju może ustrzec nas przed różnymi zakusami obcych państw, w tym przed agresją zbrojną. Bardzo dziękuję panu posłowi. Oświadczenie teraz wygłosi pan poseł Maciej Kopiec, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wydawałoby się, że praca w spółkach Skarbu Państwa to wyróżnienie łączące zarabianie pieniędzy z honorem budowania dobra wspólnego - państwowych firm, które mają tworzyć siłę gospodarczą kraju. To dlatego stawia się wymagania merytoryczne ludziom, którzy zasiadają w radach nadzorczych spółek, żeby pilnowali prawidłowego ich funkcjonowania, by podatnicy spali spokojni o los majątku, bezpieczeństwo i gospodarkę kraju, w którym żyją. Tyle w teorii. Tak byłoby, gdyby nie rządzili nami oszuści. Jak to wygląda w księstwie klakierów PiS? Na potrzeby kształcenia żon, mężów, pociotków, cyngli Prawa i Sprawiedliwości, zwykle wyszkolonych jedynie w czyszczeniu partyjnych butów, władza sprawiła sobie uczelnię - Collegium Humanum. Można w niej, na receptę prezesa oczywiście, kupić sobie dyplom MBA potrzebny do zasiadania w płatnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Taki sam dyplom na normalnej uczelni robi się przynajmniej 2 lata, inwestując kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podobno zbieżność nazwisk z Ryszardem Czarneckim, europosłem oszustem z PiS, który wyłudzał pieniądze z Parlamentu Europejskiego, jest przypadkiem, choć twarz posła jest wykorzystywana do promocji szkoły, bywa on na każdej imprezie organizowanej przez uczelnię. Rektor tej uczelni może pochwalić się wieloma osiągnięciami, wśród nich - został oskarżony o plagiat w swojej pracy doktorskiej. Sprawa trafiła do komisji i została oddalona. A skąd ta pobłażliwość? Rektorem placówki, w której mieści się komisja (Dzwonek), był pan Paweł Czarnecki. Jak miło. Wśród absolwentów tej kuźni talentów same gwiazdy: Bartłomiej Obajtek, dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku, brat prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Antoni Duda, stryj prezydenta Andrzeja Dudy, obecnie pracujący w Radzie Nadzorczej PKP Cargo. Marcin Dec, wydawca w orlenowskiej Polska Press. Swoją drogą - w maju Polska Press przyznała Collegium Humanum tytuł uczelni roku i jest to tak samo słuszne i prawdziwe, jak przyznanie Kaczyńskiemu tytułu Człowieka Wolności. Żadna inna partia nigdy nie dokonała takiego powrotu do PRL-owskiej przeszłości i rzeczywistości, jak Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu posłowi. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ze stron internetowych poświęconych zaangażowaniu rządu na rzecz polskiej młodzieży wynika, że jednym z najbardziej zapracowanych członków Rady Ministrów jest pan minister Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. Jak wynika z rządowej propagandy, pan minister niezwykle ciężko pracuje, bo nieustannie w czymś bierze udział, ciągle gdzieś dyskutuje, politykuje, odbiera tytuły dla honorowych członków, a gdy doba pozwoli, to nawet jeszcze twórczo konsultuje i dialoguje. Moi młodzi wyborcy pytają jednak pana premiera, czy na pewno na takim pełnomocniku rządu i na takiej pracy pełnomocnika rządu zależy polskiej młodzieży, która chce się czuć podmiotowo w Unii Europejskiej. Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży, a każdy taki dedykowany rok jest dla Europejczyków okazją do pozyskiwania środków na różne działania w obszarze, który w danym roku jest promowany. Mogą być one pozyskiwane bezpośrednio ze środków unijnych, ale mogą też pochodzić z budżetów państw członkowskich, które w ramach tego roku opracowały własne programy skierowane do młodzieży oraz własne systemy grantowe. I tu (Dzwonek) można by oczekiwać, że rząd, który dla realizacji polskiej polityki młodzieżowej finansuje z budżetu własnego pełnomocnika, sfinansuje także konkretne działania na rzecz polskiej młodzieży albo przynajmniej, we współpracy z Komisją, umożliwi młodzieży skorzystanie ze środków europejskich. A tymczasem mija już połowa 2022 r., a rządowych programów i całej rządowej polskiej polityki młodzieżowej, wobec młodzieży, ani widu, ani słychu. Dlatego w imieniu moich wyborców mam do pana premiera uprzejmy apel, aby pan premier poprosił pana ministra pełnomocnika o to, by w natłoku spraw reprezentacyjnych znalazł także czas i pomysł na to, jak Polacy mogą skorzystać z tej pięknej inicjatywy Komisji Europejskiej, i zwrócił się też do pana ministra Czarnka, niech porzuci badania nad cechami niewieścimi, a zajmie się wysłaniem do Komisji Europejskiej wniosku o pieniądze dla polskiej młodzieży. Mam nadzieję, że Europejski Rok Młodzieży będzie rokiem wykorzystanych - a nie zmarnowanych - szans dla polskich młodych obywateli. Dlatego proszę pana premiera z tego miejsca o osobiste zaangażowanie w tej sprawie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Taka drobna uwaga: jeśli chodzi o pana ministra Czarnka, to jego badania idą w kierunku cnót niewieścich, a nie cech niewieścich, chociaż pewnie i jedne, i drugie mają blisko siebie różnego rodzaju inklinacje i konotacje. Bardzo prosimy pana posła Tomasza Zimocha. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Od początku kadencji staram się aktywnie włączać do godnego uczczenia pamięci i oddawania przez Sejm hołdu wybitnym Polakom. W 2021 r. zorganizowałem dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs literacki ˝Tadeusz Różewicz inspiruje˝ W roku bieżącym temat konkursu brzmiał: ˝Wanda Rutkiewicz inspiruje˝, bo przypomnę, że 14 października ubiegłego roku Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 rokiem Wandy Rutkiewicz w 30. rocznicę śmierci. Wanda Rutkiewicz, co podkreślił Sejm w uchwale, nie godziła się, by zdolne alpinistki były wyłącznie broszkami w męskich wyprawach. Góry były jej światem. Pozwalały na wyjątkowe doznania intelektualne i estetyczne. Wspinanie uznawała za twórczość. Rutkiewicz tworzyła wyjątkowe dzieła. W tym roku prace nadesłane przez uczniów szkół ponadpodstawowych oceniało grono jurorów w składzie: dr Joanna Lisiewicz - polonistka, teoretyk literatury, doświadczona nauczycielka języka polskiego, Anna Kamińska - pisarka, reportażystka, dziennikarka, autorka książek biograficznych, m.in. książki ˝Wanda. Historia Wandy Rutkiewicz˝, Agnieszka Uścińska - scenarzystka, reżyserka, absolwentka filologii polskiej, dziennikarstwa i studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Dzwonek), Paweł Lęcki - nauczyciel języka polskiego w II Liceum w Sopocie, który jest, jak sam mówi, jest fanem prac domowych, Leszek Cichy - wybitny himalaista, pierwszy zdobywca Mount Everestu zimą, geodeta, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Jurorem był także poseł Tomasz Zimoch. Każdy z jurorów wyłaniał najlepszą pracę i pięć wyróżnień.

Laureatka jest także uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Trzecie miejsce zajęła Julia Chmielowska - uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach za pracę pt. ˝Szczyt˝

Piąte miejsce dla Anety Klein z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Szóste miejsce zajęła Adrianna Żeromska z Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku za pracę pt. ˝Buty marki Wanda Rutkiewicz˝

Autorka najlepszej pracy otrzymała zgodnie z regulaminem nagrodę pieniężną w wysokości 2022 zł. Gratuluję laureatom. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Przesyłam ukłony nauczycielom, pod kierunkiem których pracowali w tym konkursie uczniowie. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Wielkie brawa dla jurorów. Wykonali tytaniczną pracę. Nie ukrywam, panie marszałku, Wysoki Sejmie, że jestem w siódmym niebie - moc w młodzieży. Wielkie podziękowania również dla Danuty Stenki, która w miniony poniedziałek w Sejmie prezentowała prace laureatów podczas uroczystości zakończenia konkursu. Zachęcam do obejrzenia relacji z tej uroczystości. A ponieważ postanowiłem, że będę organizował konkursy do czasu, kiedy będę sprawował mandat posła, mam nadzieję, że jeszcze jeden raz zaproszę uczniów do literackiej twórczości. Najlepsze prace w tegorocznym konkursie zebrałem w takie oto książeczce. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Wspaniała alpinistka i z pewnością zapoznam się z tą pozycją. Dziękuję za wspaniałe oświadczenie. Proszę bardzo. Szeregowy Pośle Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ z panem posłem Jarosławem Kaczyńskim oboje jesteśmy z tego samego, warszawskiego okręgu wyborczego, to chciałabym pana posła serdecznie zaprosić na wydarzenie, które odbywa się w Warszawie, czyli na sobotni marsz równości. Żeby uczestniczyć w tym pochodzie, nie trzeba być gejem, przecież ja też nie jestem lesbijką, a biorę udział w tych paradach. To jest po prostu piękne, kolorowe święto wolności i pokazanie, że każdy ma równe prawa w naszym pięknym kraju bez względu na to, kogo kocha. Na pewno spodoba się panu ta impreza. Ochroniarze mogą sobie wziąć wolne, bo to jest pokojowe wydarzenie. Możemy nawet, panie prezesie, tak się umówić, że jeżeli pan odwiedzi marsz równości, to ja przyjdę na miesięcznicę do kościoła. To może być okazja dla nas do otwarcia się na zupełnie nowe środowiska. Na zachętę mam dla pana prezesa mały upominek, czyli tęczowe sznurówki. Ponieważ widzę, że nie ma aktualnie pana posła na sali, to przywiążę je tutaj, do mikrofonu, i będą sobie czekały na pana prezesa, aż je odbierze. Proszę pamiętać: miłość nie wyklucza. Dziękuję.

Proszę bardzo, teraz pan poseł Waldemar Andzel. Wysoka Izbo! Moje oświadczenie jest dzisiaj na temat 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski i obchodów tego święta w Katowicach. W miniony weekend w Katowicach odbyło się szereg uroczystości związanych z obchodami stulecia powrotu Śląska do Polski i pierwszym Narodowym Dniem Powstań Śląskich. Przypominam, że 20 czerwca 1922 r. Wojsko Polskie pod wodzą gen. Szeptyckiego uroczyście wkroczyło do Katowic, co oznaczało powrót części ziem Górnego Śląska do Polski. Osobiście wziąłem udział w zasadzeniu dębu w nowo powstałej al. Polskiego Dziedzictwa Śląska, a także miałem okazję zobaczyć prezentację znaczka pocztowego z okazji tego okrągłego jubileuszu. Odbyła się rekonstrukcja wkroczenia Wojska Polskiego, w której uczestniczyłem, odbył się koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, jak również msza św. w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Obchody będą kontynuowane w ten weekend w Pszczynie. Dziękuję władzom województwa śląskiego i włodarzom miasta Katowice za możliwość celebrowania tej uroczystości. Wieczna cześć i chwała za walkę dla Polski dla bohaterów z Górnego Śląska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Ponieważ nie ma na sali pana posła Pawła Lisieckiego, który był zapisany właśnie teraz do wystąpienia, bardzo prosimy panią poseł Elżbietę Płonkę o wygłoszenie oświadczenia. Wysoka Izbo! W tym roku mija 50 lat, od kiedy bullą papieża Pawła VI została utworzona diecezja gorzowska, obecnie jest to diecezja zielonogórsko-gorzowska. Pod hasłem ˝Pokój wam˝ 13 czerwca br. odbyły się jubileuszowe obchody w sanktuarium diecezjalnym w Rokitnie. Z kolei główne uroczystości miały miejsce 18 czerwca w dniu odpustu ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, patronki naszej diecezji. Była to szczególna okazja do wspólnego świętowania w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej przez duszpasterzy, osoby świeckie, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie, jak również do dziękowania za dar trwania w kościele lokalnym już pół wieku. Nie sposób wymienić wszystkich osób zarówno duchownych, jak i świeckich, które na dobre zapisały się na kartach historii naszej diecezji oraz przyczyniły się do umocnienia wiary oraz miłości chrześcijańskiej. Niewątpliwie to ich ciężka praca u podstaw zarówno na polu katechetycznym, duszpasterskim, jak i administracyjnym przełożyła się na trwanie diecezjan w duchu chrześcijańskich wartości w różnych momentach dziejowych Polski. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Gorzowie Wielkopolskim. Przypadająca w tym roku 25. rocznica pobytu papieża Polaka w sercu naszej diecezji to powód do dumy i okazja do sięgnięcia pamięcią (Dzwonek) do historycznego dziedzictwa i słów, które skierował wówczas do zgromadzonych ponad 400 tys. ludzi. Papież Polak odniósł się do korzeni naszej diecezji, które sięgają misji jej patronów, św. Braci Międzyrzeckich, pierwszych męczenników Polski, Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, a więc początku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa i pierwszych lat polskiej państwowości. Nazywa się tych męczenników Braćmi Polskimi, chociaż byli wśród nich także cudzoziemcy. Jak podkreślił Jan Paweł II, ich śmierć męczeńska obok śmierci św. Wojciecha stoi niejako na progu milenium chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Wart podkreślenia jest także fakt, iż naszych korzeni należy dopatrywać się w historycznej diecezji lubuskiej, która została utworzona w XII w. Obejmowała ona wtedy ziemie leżące w rozwidleniu rzek Odry i Warty. Mając na uwadze burzliwe losy tamtych ziem oraz męczenników, którzy przelali krew za wiarę i wolność, jesteśmy zobowiązani do podtrzymywania pamięci, trwania przy wartościach oraz przekazywania cennej lekcji historii i poświęcenia kolejnym pokoleniom. Jak mówił wspomniany wcześniej św. Jan Paweł II, naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość. Powrót do korzeni i sięganie do źródeł są w obecnych czasach niezwykle istotne. To konkretny sygnał dla nas, abyśmy umieli docenić wartość pokoju i potrafili zabiegać o niego ponad podziałami na różnych płaszczyznach. Bardzo dziękuję, pani poseł. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.